Otwieram posiedzenie. Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Rafała Bochenka oraz Roberta Gontarza, którzy prowadzić będą protokół i listę mówców. W pierwszej części obrad sekretarzem będzie poseł Rafał Bochenek.

Wysoka Izbo! Bardzo proszę o powstanie. Wysoka Izbo!

Uczcijmy jego pamięć minutą ciszy.

Wysoka Izbo! 71 lat temu w więzieniu na Mokotowie strzałem w tył głowy zamordowany został mjr Zygmunt Szendzielarz ˝Łupaszka˝, dowódca 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Wraz z nim komuniści zamordowali trzech innych oficerów, towarzyszy walki: ppłk. Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy.

Informuję, że w związku z wygaśnięciem mandatu pana posła Łukasza Szumowskiego. Proszę państwa o spokój. Informuję, że w związku z wygaśnięciem mandatu pana posła Łukasza Szumowskiego na podstawie art. 251 § 5 Kodeksu wyborczego postanowiłam o wstąpieniu na jego miejsce pana posła Rafała Romanowskiego, który zgłosił się do ślubowania poselskiego. Proszę pana posła o zbliżenie się do stołu prezydialnego. Panie i panów posłów proszę o powstanie. Obecnie odczytam rotę ślubowania. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej˝ Stwierdzam, że pan poseł Rafał Romanowski złożył ślubowanie poselskie. Obecnie, proszę państwa, przystąpimy do stwierdzenia kworum. Bardzo proszę wszystkich państwa posłów o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu. Bardzo proszę.

Stwierdzam kworum. Rada Ministrów przedłożyła pilny projekt ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, druk nr 1989. W związku z tym, na podstawie art. 73 ust. 1 regulaminu Sejmu, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o pierwsze czytanie tego projektu ustawy. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłożyła sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, druk nr 1977. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół w łącznej dyskusji nad sprawozdaniami zawartymi w drukach nr 1927 i 1928. Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół w dyskusji nad sprawozdaniem w sprawie solidarności z obywatelkami Afganistanu. Prezydium Sejmu proponuje, aby w dyskusjach nad pozostałymi punktami porządku dziennego Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycje przyjął. Informuję, że Konwent Seniorów jednomyślnie zaopiniował propozycję rozpatrzenia na bieżącym posiedzeniu informacji w sprawie realizacji sztandarowych programów polityki prorodzinnej wprowadzonych przez rząd PiS, jak np. ˝Rodzina 500+˝, ˝Za życiem˝, ˝Dobry start˝, ˝Mama 4+˝, dodatkowe świadczenie trzynasta emerytura, oraz nowego, realizowanego w ramach Polskiego Ładu, świadczenia rodzinny kapitał opiekuńczy, o której przedstawienie wnosił Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Punkty porządku dziennego bieżącego posiedzenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów. Informacja w tej sprawie, a także wykaz ustaw, które Senat przyjął bez poprawek, dostępne są w Systemie Informacyjnym Sejmu. Proszę posła sekretarza o odczytanie komunikatów.

Dziękuję bardzo.

Pani Marszałek! Wnoszę o przerwę do godz. 12 celem przedstawienia przez premiera Mateusza Morawieckiego oficjalnego stanowiska rządu w sprawie Funduszu Odbudowy. Wprowadziliście najwyższą w Polsce inflację. zabraliście Polakom pieniądze tym polskim wałem, doprowadziliście do upadku setki, tysiące polskich małych, średnich firm. a dzisiaj ustami waszych prominentnych działaczy mówicie o wycofaniu się z Funduszu Odbudowy. 250 mld zł - na to czeka polska gospodarka, na to czekają polskie firmy, czekają samorządy. A wy co? A wy próbujecie okraść Polaków z pieniędzy, które im się należą. Dlaczego? Ponieważ padł wniosek formalny o przerwę w obradach, poddam ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach do godz. 12, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Z wnioskiem formalnym pan poseł Paweł Zalewski. Proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Lewicy składam wniosek o odroczenie obrad, zwołanie Konwentu i wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego powodów rezygnacji i dymisji ministra finansów. To bardzo poważna sprawa i myślę, że pan premier powinien Wysokiej Izbie wytłumaczyć, z jakich powodów pan minister finansów tę dymisję składa i co będzie dalej. Przypomnijmy tylko, że dzisiaj mamy do czynienia z wielką inflacją, szalejącą drożyzną, ze wzrostem cen prądu, wzrostem cen gazu. Oczywiście rządzący mówią: to wszystko wina Putina, wina Unii Europejskiej, ale niestety prawda jest trochę inna. Prawda jest taka, że to jest wina waszej polityki. W związku z tym dzisiaj wnosimy o to, ażeby pan premier powiedział, jak polski rząd zamierza uporządkować sprawy finansów publicznych po wprowadzeniu tego polskiego nieładu.

Zgłoszony został wniosek formalny o odroczenie obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił. Z wnioskiem formalnym pan poseł Paweł Zalewski, Polska 2050. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Od kilku tygodni jesteśmy informowani o agresywnych zamierzeniach Rosji wobec Ukrainy, o planach wojny, którą Rosja chciałaby przeprowadzić na wschodzie Polski, w najbliższym otoczeniu. Już na Białorusi stacjonuje ok. 30 tys. żołnierzy rosyjskich. W tym czasie polski rząd kontynuuje wojnę z Unią Europejską, pojawiają się głosy o tym, że mamy zrezygnować z Funduszu Odbudowy, co oznaczałoby tak naprawdę wycofanie się z istotnych obszarów działalności Unii Europejskiej. W tym czasie pan premier jedzie do Madrytu i popiera oficjalnie panią Marine Le Pen, która głosi w kampanii wyborczej, że chce wycofać Francję z NATO.

Powiedziałam, że zwrócę się do pana ministra spraw zagranicznych. A więc wniosek pański jest trochę przedwczesny, panie pośle. Ale rozumiem, że nie wycofuje pan wniosku o zamknięcie obrad? Proszę bardzo, wniosek przeciwny, pan poseł Korwin-Mikke. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jest taka piosenka Młynarskiego: ˝Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie, co by tu jeszcze spieprzyć? I teraz, w tej chwili, po wpędzeniu Łukaszenki w objęcia Rosji, chcemy dalej jeszcze coś spieprzyć. Ja proponuję, żeby wreszcie już nie działać, nie robić ruchów prorosyjskich, nie straszyć. Kto straszy Rosją, ten działa na rzecz Putina. Dziękuję, panie pośle. Ponieważ padł wniosek o zamknięcie posiedzenia, poddam ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za zamknięciem obrad, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W nawiązaniu do głosów, które tutaj już padły, chciałbym stwierdzić, że niestety Konfederacja musi powiedzieć: A nie mówiliśmy w sprawie unijnego funduszu zadłużenia, w sprawie zadłużania przez Unię Europejską wszystkich Polaków, w sprawie tworzenia nowych unijnych podatków? Mówiliśmy o tym. W tej sytuacji, w której rząd skapitulował w tej sprawie, a teraz nie wie, co z tym zrobić, czy się wycofywać, przyznaje nam po prostu rację. Każdy kryzys jest wykorzystywany przez eurokratów do zacieśniania ich władzy. Trzeba się temu jednoznacznie przeciwstawić i Polska powinna być tym państwem, które ten proces przeciwstawiania się Unii Europejskiej z jej dążeniami totalistycznymi zapoczątkuje. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (druk nr 1989) Proszę sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa pana Janusza Cieszyńskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy, a wszystkich państwa posłów... 2 minuty przerwy, żebyście państwo mogli wyjść z sali.

Bardzo proszę sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa pana ministra Janusza Cieszyńskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Bardzo proszę, panie ministrze. Wysoka Izbo! Chciałbym w imieniu Rady Ministrów przedstawić uzasadnienie odnośnie do rządowego projektu ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. To jest, szanowni państwo, niezwykle istotny projekt, ponieważ ze względu na zmianę standardu nadawania telewizji wymuszoną decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystania zakresu częstotliwości 470-790 MHz w Unii Europejskiej jesteśmy zmuszeni dokonać przesunięcia w paśmie, na którym nadawana jest naziemna telewizja cyfrowa, a co za tym idzie - przygotować instrumenty wsparcia, które pozwolą na zmitygowanie kosztów, które w związku z tym mogłyby ponosić gospodarstwa domowe. Wynika to z tego, że.

Wiem, że zawsze jest tak jak w tym momencie, że jeszcze ktoś coś, ale mówię i do prawej, i do lewej strony, i do środka: proszę o to, żeby pan minister mógł spokojnie wygłosić to, co ma do wygłoszenia. Tak że przepraszam. Spełniam pana marzenia.

Według szacunków Krajowego Instytutu Mediów ok. 2270 tys. gospodarstw domowych w Polsce po zmianie standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej przy tym sprzęcie, który obecnie posiada, utraci możliwość odbierania sygnału naziemnej telewizji cyfrowej, czyli wszystkiego, co dzisiaj mamy na tych kanałach.

W związku z tym proponujemy racjonalny mechanizm osłonowy dla tych gospodarstw domowych, które zadeklarują, że nie są w stanie poradzić sobie z wymianą we własnym zakresie. W naszej ocenie jest to sprawiedliwe działanie, ponieważ polskie państwo czerpie bardzo duże korzyści z tego, że eksploatuje częstotliwości, które zostaną uwolnione.

To wystarczy na zakup podstawowego dekodera, a taki dekoder umożliwi odbieranie naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie. Dystrybucja kuponów, które będą niezbędne, żeby z tego skorzystać, będzie się odbywała za pośrednictwem kanału on-line oraz - ze względu na to, że w większości dotyczy to osób starszych - za pośrednictwem placówek Poczty Polskiej. W naszej ocenie jest to racjonalne rozwiązanie, pozwalające na szybkie i sprawne osiągnięcie planowanych efektów. W związku z tym gorąco liczymy na to, że cała Wysoka Izba wesprze rząd w tym działaniu. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół.

Dziękuję bardzo. Panie Marszałku!

Ta decyzja jest podyktowana ustaleniami na poziomie Unii Europejskiej, ale jest to decyzja dobra.

Zmiana ta jednak wiąże się z koniecznością dostosowania części wykorzystywanych dzisiaj odbiorników do nowego standardu nadawania.

Kupno dekodera umożliwia w dalszym ciągu niezakłócony odbiór telewizji naziemnej. Również proponowane rozwiązania, jeśli chodzi o składanie wniosków, w przekonaniu Prawa i Sprawiedliwości są racjonalne i pokazują, że wnioskodawca zdaje sobie sprawę z tego, jak wygląda realna sytuacja, jak wygląda rzeczywistość. Jak pokazują badania, znakomita większość liderów technologicznych w gospodarstwach domowych, gdzie jest naziemna telewizja cyfrowa, to osoby nie tylko 60+, ale wręcz 70+, więc wyznaczenie operatora, czyli Poczty Polskiej i jej placówek, jako miejsca, gdzie obok systemu informatycznego można składać te wnioski, jest wyjściem naprzeciw potrzebom tych osób i umożliwia im skorzystanie z tej oferty. Również zapisane w projekcie ustawy zasady przyłączania się do tego programu sprzedawców, przedsiębiorców, którzy takie dekodery oferują, są czyste, przejrzyste i nie dyskryminują żadnych podmiotów z Unii Europejskiej albo z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podsumowując, klub Prawa i Sprawiedliwości popiera to rozwiązanie i apeluje do pań i panów posłów o głosowanie za tą ustawą. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę pana posła Grzegorza Napieralskiego, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Co najmniej od 5 lat wiemy już, panie pośle, panie ministrze, że taki system nadawania będzie.

Skorzystają również na tym młodzi ludzie, dlatego że będą lepsze usługi, jeżeli chodzi o naszych operatorów telekomunikacyjnych.

Bo, przypomnę jeszcze panu ministrowi, to my wywołaliśmy ten temat i pierwszą dyskusję, bardzo poważną debatę. Dziwi mnie to, bo przecież dziś tak naprawdę ministrem cyfryzacji - to musimy sobie uświadomić - w naszym kraju jest premier Mateusz Morawiecki, który powinien pilnować tak ważnych projektów jak ten i tak ważnych zmian, które są w naszym kraju. Mam nadzieję - pan premier zawsze z tej mównicy mówił o roli opozycji, o pomocy opozycji - że doceni starania Koalicji Obywatelskiej, która już dawno temu wskazywała, że jest taki problem. Chcieliśmy o tym rozmawiać i współpracować. Tymczasem, szanowni państwo, problem jest naprawdę bardzo poważny, dlatego że do końca nie wiemy, jak duży jest - bo nie jest to dzisiaj sprawdzone bardzo dokładnie - ten problem. Brakuje aktualnych i wiarygodnych danych.

Mechanizm wsparcia jest potrzebny, panie ministrze i panie pośle. Pan poseł sprawozdawca z PiS-u poszedł. Po pierwsze, nagradza tych, którzy czekali bardzo długo na wymianę dekodera, do ostatniej chwili. A co się stanie, panie ministrze, szanowni państwo, jeżeli ktoś był na tyle solidny, na tyle poważny, że kupił dekoder, wydał pieniądze, mimo że go nie było stać, ale je uzbierał, żeby móc oglądać swoje ulubione kanały, mieć dostęp do informacji, edukacji czy nawet rozrywki? Dodatkowo oczywiście ta ustawa jest bardzo skomplikowana w wielu miejscach, bo przykładowo mówi się, że pod groźbą odpowiedzialności karnej obywatel ma złożyć oświadczenie, że nie stać go na zakup dekodera. To oznacza, że akurat dziś nie mam 100 zł, więc składam, bo akurat nie mam.

Tego nie wiemy tak naprawdę, szanowni państwo, i warto, żeby o tym porozmawiać. Ale pojawia się kolejny problem, jeżeli chodzi o tę ustawę. Robi się wielki popyt na dekodery. Pytanie, czy będzie można je kupić.

Tego niestety nie wiemy. Z tej ustawy bije jeszcze jeden bardzo poważny problem. Mnie to absolutnie zastanawia. Dlatego że widać niechęć partii Prawo i Sprawiedliwość, obecnej władzy, do samorządów.

Przecież one na co dzień w tym miejscu pomagają. Widzi, że może być problem, że mogą być wyłudzenia, więc stara się to w tej ustawie zapisać, żeby np. nie było sprzedaży obwoźnej dekoderów. Jeżeli pan pozwoli, to będzie niecała minuta. Pomimo tych wszystkich zastrzeżeń znów opozycja staje przed dylematem: poprzeć ustawę złą, która jednak rozwiązuje część problemów, czy nie popierać jej ze świadomością, że nawet kawałka problemów nie uda się rozwiązać. Znów jest to dylemat mniejszego zła czy raczej co do zasady chodzi o słuszną ideę wsparcia ludzi realizowaną w sposób spóźniony, nieprzemyślany lub bałaganiarski. Jesteśmy za skierowaniem ustawy do dalszych prac w komisji w nadziei, że chociaż część oczywistych niedostatków tej ustawy da się poprawić w trakcie prac tej komisji. Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie ministrze. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Zapraszam. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! PiS i rząd obudziły się z zimowego snu i postanowiły znowu nas zaskoczyć. Mamy ustawę pilną.

Pewnie nasz rząd postanowił wystartować w zimowej olimpiadzie w kategorii załatwiania spraw na ostatnią chwilę. Rzeczywiście w tej kategorii możemy liczyć na medale i to złote. Wsparcie gospodarstw domowych oraz realizacji tego wsparcia w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Czy dowiedzieliśmy się o tym wczoraj, miesiąc temu? Nie, wiemy o tym od kilku lat, ale działamy dzisiaj. Ta pomoc ma być w postaci świadczenia na zakup dekodera telewizyjnego. Ma się to dziać na podstawie dokumentu potwierdzającego przyznanie dofinansowania. Dofinansowanie będzie przysługiwało jednej osobie z gospodarstwa domowego, jeśli sytuacja materialna gospodarstwa domowego tej osoby uniemożliwia samodzielne ponoszenie kosztów nabycia dekodera. Kto ma więc dostać według tej ustawy te 100 zł? Bo nigdzie nie jest podane żadne kryterium dochodowe.

Czemu nam nie ogłoszono, że powinniśmy sobie odkładać te 100 zł na uzbieranie na ten dekoder. Bardzo dobrze, że państwo z naszych podatków chce nam zafundować dekodery, ale czy zdąży to zrobić przez taki krótki czas, jaki został do zmiany ustawy. Bo jak się coś robi na ostatnią chwilę, okazuje się, że pojawiają się jakieś dziwne firmy handlujące wcześniej maseczkami, pewnie teraz się pojawią firmy handlujące dekoderami, może nawet będą to te same osoby.

Kolejny punkt. Osoby, które chcą te pieniądze dostać, mają składać oświadczenie, że sytuacja materialna im na to nie pozwala. Z kolei jeszcze jeden punkt. Minister będzie ustalał wysokość kwoty, jeśli ktoś oszuka, i jaką kwotę będzie oddawał. Maksymalny limit wydatków z budżetu ma wynosić 280 mln zł. To rzeczywiście żadna suma, skoro Bielan mówi, że my nie potrzebujemy tych europejskich pieniędzy, to te 280 mln to rzeczywiście bardzo mały wydatek. Mam jeszcze takie pytanie. Kiedy i w jaki sposób rozpocznie się kampania informacyjna, co i jak z tą ustawą. Aby starsi ludzie, bo słyszeliśmy tutaj przedstawicieli rządzących, którzy uważają, że to właśnie starsi będą potrzebować tego wsparcia, dowiedzieli się, jak nie zostać oszukanym w zakupie tego dekodera. Na razie ani w telewizji publicznej, ani nigdzie indziej nie ma żadnej kampanii reklamowej mającej ułatwić ludziom załatwienie tej jednak chyba skomplikowanej sprawy. Klub Lewicy oczywiście pewnie znów będzie musiał poprzeć kolejny bubel prawny. bo bardzo boimy się, że okaże się, że sposób, w jaki ta ustawa będzie wprowadzana i w jaki te dekodery będą trafiały do gospodarstw domowych (Dzwonek), będzie kolejnym bublem prawnym. Dziękuje serdecznie. Pani poseł Urszula Nowogórska, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. Będziemy widzieli panią poseł. O, widzimy. Dzień dobry, panie marszałku, pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Koalicji Polskiej, PSL, Unii Europejskich Demokratów i Konserwatystów Marka Biernackiego w sprawie rządowego projektu ustawy, zawartego w druku sejmowym nr 1989, o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Wysoka Izbo! W uzasadnieniu do ustawy czytamy: ˝Celem wprowadzenia programu jest złagodzenie skutków społecznych zmiany standardu nadawania przez zapewnienie gospodarstwom domowym możliwości nieprzerwanego odbierania telewizji naziemnej˝ Ustawa daje możliwość dofinansowania do zakupu dekoderów w wysokości do 100 zł i budżet państwa będzie kosztowało to maksymalnie 280 mln zł.

Ustawa trafiła do nas wczoraj, dlatego należałoby się zastanowić, dlaczego ustawa procedowana jest w trybie pilnym, skoro o zmianach nadawania wiemy od dawna i znowu procedujemy coś na kolanie, i znowu procedujemy coś za pięć dwunasta. Bo przecież wiemy o tych zmianach już co najmniej od 4 lat. Trzeba również uczciwie powiedzieć, że niektórzy ponieśli już wydatki związane z zakupem nowych dekoderów. Czy nie należałoby się zastanowić, panie ministrze, nad opracowaniem regulacji prawnych, które będą dawały możliwość refundowania tej kwoty dla osób, które dokonały zakupu wcześniej i nie czekały na sam koniec? Rodzi się też kolejna wątpliwość w zakresie zabezpieczenia danych wrażliwych osób, które zadeklarowały chęć skorzystania z dofinansowania. Jak będą zabezpieczone te dane? Chodzi o to, aby zabezpieczyć ludzi właśnie przed wyciekiem ich wrażliwych danych w niepowołane ręce, by te dane nie były przedmiotem handlu i wykorzystywania do niecnych celów, tym bardziej że opinia publiczna w ostatnim czasie słyszy o różnych nadużyciach w tym zakresie. Trzeba również powiedzieć, że świadczenie będzie realizowane w sklepach stacjonarnych, internetowych, przez platformy sprzedażowe, a także przez Pocztę Polską, o czym wspomniał pan minister. Chciałam zapytać pana ministra, czy pracownicy Poczty Polskiej z uwagi na dodatkowe obowiązki wynikające z konieczności wdrożenia tej ustawy będą mieli dodatkowe wynagrodzenie. Rodzi się kolejne pytanie: Jak wyeliminować nieuczciwe praktyki i jak zabezpieczyć np. seniorów przed naciągaczami i wizytami nieuczciwych osób w miejscach ich zamieszkania? I dlatego pytam w tym momencie: Czy minister spraw wewnętrznych i administracji i komendant główny Policji wyrazili swoje stanowisko w przedmiocie tej ustawy? Panie Marszałku! Panie Ministrze! Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska podnosi rękę za każdym projektem, który służy społeczeństwu, szczególnie osobom starszym, których dochody są na niskim poziomie, i oczywiście poprzemy ten projekt. Natomiast mam nadzieję, że wszystkie uszczegółowienia, które będą w dokumentach wykonawczych do projektu ustawy, będą zawierały regulacje odnośnie do wątpliwości, o których wspomniałam. Dziękuję bardzo, pani poseł. Zapraszam pana Krystiana Kamińskiego z koła Konfederacja. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Na początek akcent humorystyczny, i państwo sami na pierwszej stronie to napisali: Rada Ministrów uznała wyżej wymieniony projekt za pilny z uwagi na potrzebę zapewnienia dostępu do bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej osobom o najniższych dochodach niekorzystających z innych form uzyskania informacji, biorąc pod uwagę konieczność przekazywania obywatelom informacji związanych z epidemią COVID-19. Przecież to jest propaganda tak toporna jak ˝Wiadomości˝ w Telewizji Polskiej. Chcą państwo dołożyć 100 zł do dekoderów, ale nawet nie potrafią określić grupy beneficjentów. Zobaczmy art. 15 pkt 3: oświadczenie osoby uprawnionej o tym, że sytuacja materialna gospodarstwa domowego tej osoby uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia dekodera telewizyjnego. W związku z tym nie dziwi, co państwo dalej napisali: ostateczna liczba gospodarstw domowych, które skorzystają ze świadczenia, nie jest możliwa do oszacowania, zatem można przyjąć, że minimalna liczba gospodarstw, które wystąpią o przyznanie świadczenia, będzie mieścić się w granicach 2270 tys., natomiast maksymalna liczba gospodarstw, które wystąpią o przyznanie świadczenia, to 14 mln. Czyli jesteśmy w granicach między wydaniem 230 mln a 1400 mln i to państwo w swoim projekcie napisali. Dodatkowo państwo zakładają, że szacowane jest wydanie 280 mln na ten projekt, co, jak widać, państwo szacują, bo nie wiedzą, jakie to będą wydatki. Robimy program, gdzie na każde 50 zł 15 zł to są koszty obsługi. Jeszcze nie ma takiego drogiego programu w Polsce.

Wiedzą państwo co? Generalnie to chyba najgorzej ukrywane rozdawnictwo pieniędzy ze wszystkich. Nie dość, że wyrzucają państwo pieniądze na obróbkę tego całego programu, to jeszcze rozdają w jakiś bardzo infantylny sposób. Dlatego jako Konfederacja składamy wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu tego projektu. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Nie chcę znęcać się nad panem ministrem cyfryzacji i powtarzać tych wszystkich argumentów, które z tej mównicy zostały podniesione, dlatego zacznę może pozytywnie. Sama zmiana systemu nadawania generalnie nie budzi zastrzeżeń. Wiadomo, że chodzi o lepszą jakość programów, oczywiście techniczną, węższy zakres częstotliwości, większą możliwość kompresji, bardziej efektywne algorytmy, a co za tym idzie - więcej kanałów, uwolnienie pewnych pasm częstotliwości, które w przyszłości będzie można sprzedać. To, że wykorzystują państwo zasoby Polek i Polaków do ingerencji na rynku, to nie jest nic nowego, dlatego że robicie to co jakiś czas. Natomiast w tym przypadku ingerujecie na pewnej części rynku, tym samym naruszacie zasady uczciwej konkurencji, a to z kolei jest sprzeczne z zasadami pomocowymi Unii Europejskiej. Liczę na to, że ten element zostanie poprawiony. Wskazują państwo na jeden konkretny standard nadawania, tak jakby nie było żadnych innych standardów nadawania.

Budujecie kolejny system dziedzinowy za grube miliony złotych dla obsługi jednego świadczenia.

Nie wiadomo, gdzie one wyciekną, kto z nich zrobi jakiś użytek, jak będą chronione. Nie za bardzo wiadomo za co, ale przedsiębiorcy będą mogli płacić kary, nie za bardzo wiadomo, na jakich zasadach, nie za bardzo wiadomo, kto to ma egzekwować, ale bat oczywiście musi wisieć.

Koło Polska 2050 liczy na to, że na etapie prac w komisji przynajmniej kilka absurdów zostanie wyeliminowanych.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Robert Kwiatkowski, koło Polska Partia Socjalistyczna. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Zdaje się, że to jest ten przypadek. Zacznijmy litościwie od tych dobrych chęci.

Samo w sobie jest to dość korzystne.

Druga dobra rzecz, Wysoka Izbo, to chęć wsparcia w transformacji technologicznej najuboższych. Dalej już jest gorzej, ponieważ żeby to osiągnąć, wymyślono konstrukcję rodem z ministerstwa dziwnych kroków albo stworzono takich mechanizm, w którym łatwo wykazać błędy i potknięcia, ale nie sposób znaleźć zalet tego rozwiązania. Zapominacie, że co miesiąc tym samym ludziom, tym samym gospodarstwom domowym zabieracie 25 zł w postaci abonamentu. Czy nie lepiej byłoby połączyć jedno z drugim i zwolnić ludzi przez 4 miesiące z płacenia abonamentu?

Przecież media publiczne i tak w lwiej części są dzisiaj finansowane z budżetu. Ot i cała filozofia. Wydaje mi się, że trudno o prostsze rozwiązanie.

Będziemy wnosić poprawkę do tej ustawy.

Chodzi o zwolnienie z płacenia abonamentu dla każdego gospodarstwa domowego przez 4 miesiące. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do zadawania pytań. Ustalam czas zadawania pytania na 1 minutę. Do pytań zgłosiło się 14 osób. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej jest bardzo dobrym projektem. Dziękuję panu ministrowi i rządowi za przygotowanie go. Jest to kolejne wsparcie gospodarstw domowych w związku ze zmianami, które wprowadzane są w wyniku decyzji Unii Europejskiej. Ta dyskusja, która przed chwileczką się wywiązała, świadczy o tym, że państwo jako totalna opozycja potraficie skrytykować każdy projekt, nawet projekt wspierający polskie rodziny. Panie Ministrze! Kto wtedy rządził, to państwo doskonale wiecie. Panie ministrze, czy wtedy rząd przygotował jakikolwiek program wsparcia gospodarstw domowych? Jakie kwoty (Dzwonek) zostały na ten program wydatkowane? Dziękuję bardzo. Pan poseł Michał Szczebra. Przepraszam, Michale. Panie Marszałku! Jest takie powiedzenie: zima zaskoczyła drogowców. Cyfrowa telewizja naziemna zaskoczyła nieobecnego przez chwilę pana ministra Cieszyńskiego.

Czy ma pan jakiekolwiek dane?

Ostatnia sprawa. W mojej opinii zarobi znowu Poczta Polska. Tak jak na pulsoksymetrach i na innych usługach, które realizowała. Cały czas odpłacacie się za wybory kopertowe, które przyniosły tej spółce straty. Ile zarobi Poczta Polska na tej usłudze, na dostarczaniu kodów wszystkim zainteresowanym, którzy nie korzystają z poczty elektronicznej? Panie Marszałku! Panie Ministrze! W projekcie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej czytamy przy harmonogramie: świadczenie na zakup dekodera telewizyjnego uprawnia do otrzymania dofinansowania do zakupu jednego dekodera telewizyjnego w gospodarstwie domowym, umożliwiającego co najmniej odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC. Panie ministrze, co ten dekoder, oprócz tego ˝co najmniej˝ dotyczącego telewizji, będzie odbierał? Czy będzie można łączyć go z jakimiś innymi rzeczami związanymi z, nie wiem.

Proszę bardzo. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałoby się powiedzieć: pilny projekt ustawy, a nasuwa się pierwsze pytanie, od kiedy państwo wiedzieliście o tym, że zmieniamy system na inny.

Panie ministrze, konkretne pytanie: Dlaczego działacie państwo w takim chaosie, dlaczego wiedząc od kilku miesięcy o tym, że rozpoczynamy w ogóle takie prace, właściwie od miesięcy to już trwa, w takim trybie wprowadzacie dzisiaj takie rozwiązania?

Dziękuję serdecznie. Pan poseł Michał Urbaniak, koło Konfederacja. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Panie Ministrze!

Już w samym uzasadnieniu zakładają państwo, że ceny dekoderów w związku z waszym projektem mogą być wyższe, ale to nie szkodzi, bo przecież wy dokładacie tylko po 100 zł.

Wysoka Izbo! Stawiam pytanie, czy taka procedura notyfikacyjna została przeprowadzona. Kiedy złożono odpowiednie dokumenty i jakie było stanowisko organów unijnych? To są bardzo istotne elementy procesu legislacyjnego, który z konieczności fundują nam państwo w takim właśnie szalonym pędzie. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzień dobry, panie ministrze. W Ministerstwie Zdrowia zasłynął pan ze słynnych respiratorów. Pan minister Szumowski złożył rezygnację z mandatu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała panu ten przetarg z wiadomych powodów. No jak?

Przychodzi pan w ostatniej chwili, kiedy wiadomo, że te dekodery trzeba będzie wymieniać w ciągu 3 miesięcy. Bo był już handlarz bronią, był już instruktor narciarstwa.

Otóż jak patrzę na pana doświadczenia, a trudno nazwać pana człowiekiem sukcesu, biorąc pod uwagę to, co pan robił, to obawiam się, że 2 mln ludzi może zostać bez sygnału telewizyjnego. Pan poseł Jan Szopiński, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Cała ta ustawa sprowadza się do dwóch pytań. Po pierwsze, czy polska administracja faktycznie nie ma co robić? Po drugie, jeśli administracja pocztowa nie ma co robić, to ile tak słabo opłacani pracownicy poczty z owych 15 zł, które kasujecie ze 100 zł, otrzymają? Niech pan, panie ministrze, powie, ile ci pracownicy otrzymają tych pieniędzy. Natomiast mam dla pana bardzo logiczną podpowiedź.

Przecież każda osoba płacąca abonament mogłaby skorzystać na równych zasadach z dobrodziejstwa rządu. Panie ministrze, poproszę o odpowiedź tutaj wszystkim Polakom i poproszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo. Pan poseł Mieczysław Kasprzak, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Prosta sprawa, a tyle komplikacji, tyle uwag.

A rozwiązanie jest proste, poseł Kwiatkowski o tym mówił - zwolnić z abonamentu. Od 2 lat leży projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego mówiący o tym, żeby wszystkich Polaków zwolnić z abonamentu. Za 700 mln mamy wszystkich zwolnionych z abonamentu. Kiedy zgłaszaliśmy ten projekt, mówiło się, że brak pieniędzy, że telewizja nie przeżyje tego. Państwo w kampanii wyborczej bąkaliście coś pod nosem (Dzwonek), że trzeba ludzi zwolnić z abonamentu. I moje pytanie: Czy chcecie to zrobić czy nie? Dziękuję bardzo. Pani poseł Marta Wcisło, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Ustawa zwana pilną. Od 5 lat wiadomo, że w Polsce od czerwca tego roku ma się zmienić system nadawania telewizji cyfrowej. 4 miesiące przed tym wprowadza w trybie pilnym ustawę. Nie było takiej ustawy w przypadku ustawy COVID-owej, w przypadku ustawy dla przedsiębiorców, ale w przypadku ustawy o wymianie dekoderów jest. Ja się zastanawiam, dlaczego to akurat pan. Pan został wczoraj pełnomocnikiem do spraw naprawy Polskiego Ładu. Ja się boję o ten Polski Ład, a właściwie o obywateli. Ale pan budzi emocje, panie ministrze. Też się zaczynam bać. Bardzo proszę. Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze!

Czy te dane mają posłużyć później weryfikacji, kto płaci abonament, kto nie płaci? Bo przecież placówki pocztowe. Bo pełne dane będą dostępne u ministra cyfryzacji. Czy również temu w przyszłości posłuży zbieranie tych danych od osób, które otrzymają to dofinansowanie? To chyba jedno z zasadniczych pytań, jakie padły. Przepraszam, że oceniam, ale taka refleksja. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Moje pytanie jest proste i już było tu powtórzone, ale mimo wszystko je zadam. Proszę mi powiedzieć: Co ma być w tym dekoderze jeszcze innego? Jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, to ja się martwię, że te dopłaty dostaną tylko ludzie, którzy są związani z PiS. Tak zawsze jest, że. Może być to śmieszne, ale ja tak uważam, że w pierwszej kolejności. Mówię to dlatego, że nie mam za grosz zaufania do pana. A więc ja uważam, że PiS doprowadzi do tego, że będziemy płacić za wszystko (Dzwonek), za te... zapomniałam, kurde. dekodery, dekodery też.

Dziękuję bardzo. Pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! To, że w tym roku zmieni się standard nadawania telewizji naziemnej, było wiadomo już od dawna. Tymczasem ustawa określająca zasady przyznawania i realizacji świadczenia na zakup dekodera telewizyjnego procedowana jest dopiero teraz, a powinna wejść pod obrady odpowiednio dużo wcześniej. Z badań Krajowego Instytutu Mediów wynika, że ok. 2,3 mln polskich gospodarstw domowych nie jest przystosowanych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Co w sytuacji, jeżeli gospodarstwa domowe będą zmuszone kupić nowy telewizor, gdy okaże się, że wymiana samego dekodera nie wystarczy? Komplikujecie życie Polaków - jak zwykle, tradycyjnie. Dajecie 100 zł dopłaty do dekodera i jeszcze zobowiązujecie Polaków do składania oświadczeń. Mam nadzieję, że ta ustawa (Dzwonek) zostanie doprecyzowana w trakcie prac komisji, bo w proponowanej formie jest nie do przyjęcia. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jestem wielkim zwolennikiem tego, by wspierać gospodarstwa domowe, ale jestem przeciwnikiem chaosu i skomplikowanych przepisów. Państwo, rząd PiS-u doskonale wiedział, wiedział o tym od 4 lat, że jest taka sytuacja, i w zasadzie w ostatnim momencie przedstawiacie projekt ustawy. Takie sprawy załatwia się dużo, dużo wcześniej. System jest niejasny, jest skomplikowany. Oczywiście rozumiem, że państwo chcecie znowu wyjść i powiedzieć, że oto rząd PiS-u pięknie dba o gospodarstwa domowe, o mieszkańców i każdemu da 100 zł. Nie wiem, czy jest to dobre rozwiązanie. Co z osobami, które już zapłaciły tę kwotę?

Dziękuję bardzo. Panie ministrze, zapraszam. Ma pan trudne zadanie, ale mamy nadzieję, że da pan radę.

Bardzo dziękuję. Otóż tak. Państwo z opozycji chcecie zwolnić z abonamentu. Będzie niższy abonament, per saldo wyjdzie tak samo. Przeczytam, to państwo może się zreflektujecie, czy to na pewno jest taki dobry pomysł. Osoby od 75. roku życia lub od 60., jeżeli pobierają emeryturę. Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i rentę socjalną. Osoby pobierające zasiłki, osoby niesłyszące, niewidome i inwalidzi I grupy. Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego. Osoby bezrobotne, inwalidzi wojenni, wojskowi i weterani. To są osoby, które w projekcie Polskiej Partii Socjalistycznej - chapeau bas - będą wykluczone z otrzymania wsparcia, a to są, szanowni państwo, osoby, które w mojej ocenie przede wszystkim powinny z tych możliwości skorzystać. Państwo zadajecie szereg pytań, że jest jakieś oświadczenie, że jest odpowiedzialność. Oczywiście. że jest oświadczenie, że jest odpowiedzialność karna za złe oświadczenie. Tak, szanowni państwo, dlatego że my ufamy Polakom i wierzymy w to, że te osoby same najlepiej potrafią ocenić to, czy je na to stać, czy nie. Jak słyszę od parlamentarzystów z opozycji, którzy mówią, że złożą na to posłowie, to mam jedno pytanie: Czy państwu nie jest wstyd tak pytać? Naprawdę.

Dlatego myślę, że mieszanie tego naprawdę nie jest w porządku. Mówili też państwo o propozycjach komisji. Ale czy jest jakiś komisyjny projekt w tej sprawie?

Ja jestem zawsze otwarty na dyskusję. Przecież nawet podczas szczytu cyfrowego w Katowicach mieliśmy bardzo ciekawą komisję, rozmawialiśmy normalnie jak ludzie, a tutaj, jak są konkrety, państwo od razu idą w politykę. A na koniec co przyznajecie? Że to jest dobry projekt.

Państwo pytacie o dane wrażliwe. Jeżeli chodzi o adres, e-mail i numer telefonu, to praktycznie te dane wielu obywateli, 8 mln są w Rejestrze Danych Kontaktowych, w urzędach skarbowych, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w e-zdrowiu.

Pan poseł Gramatyka pytał czy właściwie stwierdzał, że ingerujemy w rynek. Szanowny panie pośle, ingerujemy w taki sposób, że w momencie, w którym zmienia się standard, przestaje działać jakiś konkretny standard i zmienia się na inny, to dajemy możliwość skorzystania właśnie z takiego standardu. To jest też to pytanie, które pan poseł Adamczyk i pani poseł Krzywonos zadali, mówiąc, że co najmniej HEVC. To, szanowni państwo, wynika z tego, że są takie dekodery, które obsługują kilka standardów na raz. Gdybyśmy wpisali tylko jeden, to właśnie wtedy w nieuprawniony sposób zaingerowalibyśmy w rynek. I jeszcze pytanie drugie czy też stwierdzenie pana posła Gramatyki, że to bat na firmy. Tak. Wie pan na jakie firmy? Na te, które dzisiaj na najpopularniejszym polskim serwisie aukcyjnym oferują dekodery, które od czerwca przestaną działać. Na te firmy jest wprowadzony bat. I przyznaję, biję się w pierś: powinien być wprowadzony znacznie wcześniej, bo to jest najzwyczajniej w świecie oszukiwanie Polaków, panie pośle, i powinien pan sobie z tego zdawać sprawę. Pani minister Józefa Szczurek-Żelazko pytała, jak to było w 2013 r., kiedy rządziła Platforma Obywatelska. Czy wtedy (Dzwonek), kiedy zmieniał się standard cyfrowej telewizji, było jakieś wsparcie od rządu? Było. Od rządu Włoch, od rządu Hiszpanii, Słowacji, Litwy, Węgier i Bułgarii, bo od rządu Platformy Obywatelskiej obywatele nie dostali nic. Dziękuję serdecznie. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. W związku z tym do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druki nr 1699 i 1975) Bardzo proszę pana posła Jarosława Sachajkę o przedstawienie sprawozdania komisji. Zapraszam, panie pośle. A panu ministrowi dziękuję serdecznie za udział w obradach.

Panie marszałku, nie ma nikogo z Ministerstwa Zdrowia, nie wiem, czy to ważne.

Po prostu nie ma nikogo z Ministerstwa Zdrowia.

Odsłucha. Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu połączonych komisji: Komisji Zdrowia oraz komisji rolnictwa sprawozdanie komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wówczas pani marszałek skierowała ten druk do połączonych komisji: komisji rolnictwa oraz Komisji Zdrowia. Komisja Zdrowia w dniu 25 stycznia przygotowała sprawozdanie komisji. Jest to druk nr 1975. Osiem poprawek zostało przyjętych, pięć poprawek zostało odrzuconych. Zgłoszono cztery wnioski mniejszości. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Nadal nie ma nikogo z ministerstwa. Przykro mi. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Bardzo serdecznie proszę pana posła Krzysztofa Szulowskiego z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o zabranie głosu. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani autorstwa posłów Kukiz’15 i Prawa i Sprawiedliwości, druki nr 1699 i 1975. Celem projektu jest znowelizowanie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani w zakresie kwestii dotyczących upraw i zbioru konopi innych niż włókniste w celu uzyskania surowca farmaceutycznego.

Przypomnę też, że parlament był w większości prawicowy i stało się to głosami przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości. Na podstawie obecnych przepisów po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste oraz żywica konopi innych niż włókniste mogą stanowić surowiec farmaceutyczny do sporządzania leków recepturowych. Dodatkowo kwestie te reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r. Natomiast obszar dotyczący sporządzania i wydawania produktów leczniczych, leków recepturowych jest obwarowany wymogami określonymi w szczególności w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Najważniejszą propozycją zawartą w projekcie jest ta, aby uprawy i zbiór konopi innych niż włókniste, z których będą sporządzane dopuszczone do obrotu produkty lecznicze, były prowadzone po uzyskaniu zezwolenia głównego inspektora farmaceutycznego przez polski instytut badawczy nadzorowany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Zezwolenia te będą wydawane w formie decyzji przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny po zasięgnięciu opinii komendy wojewódzkiej Policji. Istotna będzie kwestia sposobu zabezpieczenia upraw przed dostępem osób nieuprawnionych, w tym poprzez konieczność prowadzenia wykazów osób uprawnionych do wejścia i pojazdów uprawnionych do wjazdu.

Jest to technologia zdalnego radiowego nadzoru roślin, która wykorzystuje fale radiowe do odczytu i przesyłania danych zawartych na etykiecie naniesionej na każdą z uprawianych roślin, umożliwiając identyfikację każdej z tych roślin znajdujących się jednocześnie w polu odczytów. Klub Prawa i Sprawiedliwości wyraża poparcie dla projektu. Poprzez przyjęcie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, jak wspomniałem, zgodziliśmy się na wykorzystanie surowca z konopi innych niż włókniste jako surowca farmaceutycznego. Pora na to, aby surowce pochodziły z polskiej, w pełni kontrolowanej uprawy, a nie z zagranicy. Mamy zapewnienia, że Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu lub ewentualnie inna jednostka mają wiedzę, potencjał i infrastrukturę, aby taką uprawę prowadzić i pozyskiwać surowiec. Uzyskiwanie surowca w kraju sprawi, że nie będziemy musieli sprowadzać go z zagranicy. Pozwoli to znacznie obniżyć jego cenę, a więc i cenę leków recepturowych przepisywanych pacjentom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.

Witam pana ministra. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Sama idea usankcjonowania prawnego uprawy w Polsce konopi innych niż włókniste, czyli zawierających znaczną ilość THC, czyli tetrahydrokannabinolu, jest całkowicie słuszna. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zalegalizowała obrót lekami opartymi na marihuanie, ale jednocześnie nie umożliwiła krajowej uprawy konopi innych niż włókniste. Nie było w tym większej logiki. W tej sytuacji leki z marihuaną leczniczą muszą być sprowadzane z zagranicy. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest ich bardzo wysoka cena. Ustawa wskazuje instytucje, które powinny wydawać zezwolenia na uprawę w Polsce konopi innych niż włókniste, oraz dość szczegółowo określa minimalne wymogi infrastrukturalne, jakie powinno spełniać miejsce uprawy, i różnego rodzaju wymogi bezpieczeństwa, w tym sposób zabezpieczenia upraw przed kradzieżą. Kontrola działalności podmiotu zajmującego się uprawą miałaby być przypisana wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym. Przy okazji projektu ustawy autorzy proponują zmianę definicji konopi włóknistych dopuszczanych w Polsce do uprawy i wskazują, że są to rośliny z gatunku konopie siewne, w których THC nie przekracza 0,3% w przeliczeniu na suchą masę. Z punktu widzenia hodowców, plantatorów przemysłowo wykorzystywanych konopi włóknistych jest to zmiana bardzo korzystna.

Słabością ustawy jest wskazanie instytutów badawczych jako jedynego podmiotu mogącego starać się o uzyskanie pozwolenia na produkcję konopi indyjskich. Tłumaczenie autorów projektu i ministerstwa, iż ta regulacja wynika z podpisanych kilkadziesiąt lat temu przez Polskę zobowiązań, jest całkowicie nieprzekonujące i trudne do zweryfikowania. Wpisane w ustawę ograniczenie możliwości starania się o pozwolenie na uprawę konopi indyjskich przez podmioty inne niż instytuty badawcze de facto wskazuje z imienia i nazwiska Instytut Roślin Włóknistych i Zielarskich z Poznania. Należy przypuszczać, że jak w przypadku każdego monopolu brak konkurencji spowoduje, iż nie dojdzie do oczekiwanej skali obniżki cen leków zawierających marihuanę leczniczą. Jak wiemy, w Sejmie pojawił się równolegle projekt dotyczący tego samego tematu. Myślę tu o sygnowanym przez Lewicę poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1701. Projekt ten został przez większość sejmową odrzucony w pierwszym czytaniu. Podobnie jak omawiany tu projekt ustawy autorstwa Kukiz’15 projekt z druku nr 1701 miał na celu umożliwienie w Polsce uprawy konopi innych niż włókniste oraz nadzoru nad tymi uprawami, ale dodatkowo rozszerzał pole zainteresowania o inne aspekty uprawy i przerobu konopi zawierających znaczną ilość THC.

Błędem jest odrzucenie przez Komisję Zdrowia proponowanych poprawek, które mogły spowodować, że ustawa stałaby się kompilacją dwóch równoległych propozycji i rozwiązałaby inne pojawiające się przy okazji dyskusji o marihuanie leczniczej problemy. Między innymi chodzi tu o wprowadzenie do polskiego porządku prawnego pojęć: stan po użyciu tetrahydrokannabinolu i stan upojenia tetrahydrokannabinolem, analogicznych do pojęć: stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości, czy o możliwość refundacji części kosztów leków opartych na marihuanie leczniczej. Klub Koalicji Obywatelskiej ma świadomość niedoskonałości omawianej ustawy, jednak wobec braku możliwości uchwalenia przez ten Sejm lepszego prawa, biorąc pod uwagę przede wszystkim dobro pacjentów czekających na obniżenie ceny marihuany leczniczej, co nie nastąpi bez umożliwienia produkcji konopi innych niż włókniste w Polsce, klub Koalicji Obywatelskiej poprze projekt ustawy. Zapraszam. Wysoka Izbo! 13 stycznia br. parlamentarzyści i parlamentarzystki zajęli się trzema projektami ustaw dotyczących konopi, z czego dwa odnosiły się do medycznej marihuany. Mowa tutaj oczywiście o projekcie sygnowanym przez posła Jarosława Sachajkę z druku nr 1699 i o projekcie z druku nr 1701, który miałam przyjemność przedstawiać Wysokiej Izbie. Obydwu projektom przyświecał wspólny cel, a mianowicie ułatwienie legalnej uprawy marihuany medycznej w Polsce, której pilnie potrzebują pacjenci, aby terapia tym lekiem była bardziej dostępna, z tą różnicą, że zaprezentowane wtedy przeze mnie rozwiązania, który były efektem solidnej i sumiennej pracy w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Legalizacji Marihuany, dotykały tematu znacznie szerzej i z kilku ważnych perspektyw. Mam na myśli chociażby umożliwienie większej liczbie podmiotów legalnej uprawy konopi, zniesienie zakazu refundacji medycznej marihuany, umożliwienie prawnego wprowadzenia stanu po użyciu THC czy edukacji lekarzy i farmaceutów. Niestety podczas posiedzenia projekt ten został odrzucony, choć decyzja ta nie została poparta żadnym merytorycznym uzasadnieniem. Szkoda, bo nie zawierał on żadnych kontrowersyjnych zapisów, lecz stanowił konkretną odpowiedź na bolączki polskich pacjentów. Projekt sygnowany przez posła Sachajkę został skierowany do dalszych prac. Wtedy też zapowiedziałam, że nie będę się poddawać, będę dążyła do wprowadzenia dobrego prawa w zakresie medycznej marihuany. Dlatego podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia wspólnie z posłanką Marceliną Zawiszą zgłosiłam kilka istotnych poprawek do omawianego dzisiaj projektu ustawy, które mogłyby sprawić, że wcielenie jej w życie przyniesie nieco więcej korzyści, niż pierwotnie sam ten projekt zakładał. Przede wszystkim oprócz zmiany zapisów w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii zaproponowałyśmy, aby dokonać ich także w ustawie o refundacji leków. Miałby pojawić się w niej zapis o wydawaniu specjalnych zaświadczeń dla pacjentów leczących się medyczną marihuaną, aby uniknąć wszelkich nieporozumień i zbędnych konfrontacji z policją, która z góry zakłada, że ma do czynienia z nielegalną marihuaną. Takie zaświadczenie, czy elektroniczne, czy papierowe, to mała rzecz, a może pomóc pacjentom w wielu sytuacjach. Złożyłyśmy także poprawkę, która jasno stanowi, że nie popełnia przestępstwa ten, kto przetwarza lub przerabia na własny użytek produkty lecznicze przygotowane z konopi innych niż włókniste. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii wskazuje, że takie działanie jest zakazane, ale nie konkretyzuje, czy dotyczy to także medycznej marihuany. Dlatego najwyższy czas rozwiać wszelkie wątpliwości i doprecyzować tę kwestię prawnie. Podczas prac komisji zaproponowałyśmy także bardzo ważną poprawkę, która zniosłaby nareszcie zakaz refundacji medycznej marihuany. Terapia nią, zwłaszcza kiedy nadal musi być sprowadzana z zagranicy, nie jest tania. Pragnę podkreślić, że ta poprawka nie obligowałaby państwa do refundacji, ale pozostawiałaby ministrowi zdrowia prawną możliwość podjęcia takiego kroku i wskazania, w jakich przypadkach, przy jakich chorobach ta refundacja byłaby możliwa dla pacjentów. Powyższe poprawki z pewnością wzmocniłyby pozytywny wpływ projektu ustawy posła Sachajki z druku nr 1699 i w kilku istotnych kwestiach rozwiązałyby przede wszystkim problemy polskich pacjentów korzystających z terapii medyczną marihuaną. Ta ustawa to i tak jest dziś krok naprzód, ale moim zdaniem powinniśmy jako posłowie i posłanki, którzy pracują w tej Izbie, mieć odwagę zrobienia nieco większego ruchu, tak aby Sejm podszedł do tematu kompleksowo, z korzyścią dla pacjentów i polskiego rolnictwa. Z pewnością Lewica poprze ten projekt, ale też prosimy Wysoką Izbę o poparcie tych wniosków mniejszości wynikających z poprawek, które zgłaszałam w komisji i które przed chwilą omówiłam. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę pana posła Radosława Lubczyka, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

My mówiliśmy dość jasno, pytaliśmy, dlaczego nie mogą tego robić rolnicy, którzy też przecież mogliby mieć takie możliwości, dlaczego to jest przypisane tylko do tej jednej instytucji. Klub Koalicji Polskiej oczywiście będzie popierał tę ustawę, idzie to w dobrą stronę, a mam nadzieję, że kolejny krok to będą kolejne łagodzenia.

Ale, panie marszałku, ta ustawa nie budzi wielkich kontrowersji, stąd, jeśli pan marszałek pozwoli, ja jednak będę mówił o czymś innym.

Kolejna osoba, kolejny przypadek. Nie mam ze sobą rachunku, ale jeśli będziecie tu państwo, to ten rachunek za chwilę zorganizuję i wam pokażę.

To 1000% podwyżki za gaz. Gdzie wy jesteście?

To zaczynają być rzeczywiście tragedie ludzkie, a wy dalej nie macie żadnego planu działania. Działacie od ściany do ściany. Jaki jest pomysł na to, żeby tym ludziom pomóc? Te raty cały czas rosną galopująco. Może wam się wydawać, że 500 zł dla normalnej rodziny to jest nic, ale dla ludzi, którzy normalnie żyją od pierwszego do pierwszego to są strasznie duże wydatki. To naprawdę boli polskich obywateli. Zastanówcie się, co wy robicie, gdzie wy jesteście. Ludzie naprawdę są zdesperowani. Ludzie naprawdę są zdesperowani, panie pośle. Rozumiem, że do pana też przychodzą i zastanawiają się, skąd mają na to wszystko brać. Przecież widzimy tę drożyznę. Widzimy dzisiaj tę drożyznę. To są realne osoby, które do mnie przychodzą i płaczą. To wy rządzicie od 5 lat, doprowadziliście do takiej sytuacji. Zacznijcie rządzić, zacznijcie pomagać tym ludziom, bo są rzeczywiście problemy, za chwilę będą tragedie. Dzisiaj są nieszczęścia, za chwile będą tragedie. Bardzo dziękuję. Panie pośle, zawsze mam dylemat w takiej sytuacji, bo prowadzimy dyskusję na temat ustawy w sprawie marihuany.

żebyście nie krzyczeli do siebie: za dużo się napaliłeś albo coś takiego, bo to nie jest rozsądne. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowni Państwo! Znów zastanawiamy się, czy, w jaki sposób, z jakimi ograniczeniami, do jakich celów zalegalizować określoną substancję. Tymczasem powinniśmy się zastanowić, czy państwo w ogóle ma prawo i czy państwo powinno interesować się tym, co dorosły człowiek je, pije, przyjmuje, pali itd. Oczywiście, że tak. Jednym z przykładów jest alkohol. Alkohol to oczywiście substancja psychoaktywna, silnie uzależniająca, nadużywana bardzo szkodliwa. To jest oczywiście narkotyk, tyle że różni się od innych narkotyków tym, że jest legalny. No i powiedzmy o tym alkoholu. Poza powodowaniem śmierci bezpośrednio nadużywanie alkoholu prowadzi do wielu chorób śmiertelnych, prowadzi do rozbijania rodzin, uzależnienie od alkoholu powoduje mnóstwo przestępstw, w tym morderstw. Tymczasem wy skupiacie się tylko na substancjach, które w tym momencie są nielegalne, tak jakby zakaz używania substancji zatrzymywał używanie tej substancji. Statystyki pokazują, że to oczywiście nie działa. Teraz narkomania jest większa niż za czasów, kiedy narkotyki nie były zakazane.

Oczywiście skończyłoby się to tak jak w USA za prohibicji, kiedy nadal był używany alkohol tylko dodatkowo były mafie, morderstwa, rozboje, kradzieże. Dlaczego jest tak, że nikt nawet nie wspomni o zakazie i karaniu za alkohol, o prohibicji alkoholowej, a wszyscy bronią tego, żeby była prohibicja narkotykowa? To jest tyrania status quo, o której mówił Milton Friedman. To, żeby alkohol był legalny, opłaca się tym, którzy zarabiają obecnie na tym miliony, lobbują za tym, żeby był legalny, płacą łapówki, pilnują tego. Natomiast to, żeby pozostałe narkotyki były nielegalne, jest w interesie mafii narkotykowych, które lobbują, przekupują, przekonują, żeby narkotyki były nielegalne.

Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Mam zawszę tę sposobność występowania po osobie, po przedstawicielach koła, z którymi się dramatycznie nie zgadzam, ale ponieważ czasu mało, więc nie będę obalała tych tez, które przed chwilą usłyszeliśmy. I to dobrze, że jesteśmy w stanie rozmawiać o marihuanie leczniczej czy bardziej o terapiach związanych z leczniczą marihuaną bez fobii, bez przesądów, tylko w normalnym trybie. Co więcej, te trzy projekty, nad którymi się pochyliliśmy, to projekty pochodzące z trzech bardzo skrajnie różnych środowisk politycznych, a mimo to postulaty, które się w nich pojawiają, są bardzo do siebie podobne. I najważniejsze w tej ustawie jest to, że dzieje się to wszystko z ogromną korzyścią dla osób chorych, które tych terapii marihuaną leczniczą potrzebują.

To było absolutnie nieludzkie, więc dobrze, że to zmieniamy, pracując nad tymi trzema ustawami. Umożliwienie produkcji w Polsce to przede wszystkim dobry krok w kierunku chorych, dobry krok w kierunku polskiego budżetu, w kierunku polskich hodowców. Tak jak mówię, tak jak powiedziałam na początku, dobrze, że odrzuciliśmy fobie i pracujemy nad tym projektem. Najważniejsze zmiany.

To ważne. Po drugie, poddaje się standaryzacji pobór i badanie próbek. Czyli nie będzie już takiej sytuacji, że ktoś jest przestępcą lub nie jest przestępcą, w zależności od tego, czy próbka jest pobierana i badana przez Policję, czy przez ARiMR, a tak bywało w przeszłości.

To wszystko są dobre zmiany.

Dziękuję bardzo. Zapraszam pana posła Jarosława Sachajkę. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Kukiz’15 - Demokracja Bezpośrednia mam zaszczyt przedstawić stanowisko co do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jest on uzupełnieniem ustawy, która została przyjęta w 2017 r. i która pozwoliła na to, aby polscy pacjenci mogli kupować konopie medyczne w aptekach. Właściwie od lat słyszymy tutaj o tym, że wiele ugrupowań politycznych walczyło o to, żeby polscy pacjenci mogli korzystać z konopi medycznych, z terapii na podstawie konopi medycznych.

Ustawa została przyjęta, jednakże z naszego projektu w ubiegłej kadencji wycięto cały fragment związany z uprawą konopi w Polsce. W tej kadencji złożyliśmy projekt delikatnie różniący się od tego, który był w ubiegłej kadencji, i jest zgoda na to, aby polskie instytuty, instytuty podległe ministrowi rolnictwa uprawiały konopie medyczne do celów farmaceutycznych.

Druga bardzo ważna deklaracja jest taka, że te konopie będą w dużo lepszej cenie niż są obecnie, bo obecnie ta cena dla wielu pacjentów jest zaporowa.

Konopie medyczne powinny być uprawiane pod ścisłym nadzorem państwa. Za chwileczkę będziemy rozmawiali o konopiach siewnych i tam rolnicy mają pełną swobodę. Tutaj pod nadzorem państwa instytuty podległe ministrowi rolnictwa już wkrótce zaczną uprawiać konopie medyczne. Dziękuję. Pan poseł Andrzej Rozenek, koło Polska Partia Socjalistyczna. Bardzo proszę. Wysoka Izbo!

Przecież to jest niepoważne. To jest zwykła roślina. To jest roślina, którą nasze babcie, nasi dziadkowie hodowali, uprawiali w swoich ogródkach. Nikomu to nie przeszkadzało. Od konopi indyjskich, od marihuany nikt na świecie nie umarł. Nie ma takiego przypadku. Od alkoholu, oczywiście, ludzie umierają, od tytoniu ludzie umierają. Od konopi nikt nie umarł, a wy zakazujecie tej rośliny. Dyskutujemy nad tym, że będzie można w określonych warunkach uprawiać te konopie po to, żeby je sprzedawać w aptekach pod nadzorem lekarzy. Okej, dobrze, ludzie potrzebują tego lekarstwa. Główny inspektor farmacji będzie wydawał zezwolenie, a potem to zezwolenie będzie jeszcze podlegało opinii komendy wojewódzkiej Policji. Ludzie, co tu się dzieje? Policja będzie pilnowała uprawy krzaczków.

Poprzednia ustawa doprowadziła do tego, że dwie firmy, i to zagraniczne, mogą sprzedawać konopie w polskich aptekach. Wiecie, co to jest? Korupcja w biały dzień. Po prostu. Co to ma być w ogóle? Czym to się różni? Większość stanów w Stanach Zjednoczonych już zalegalizowała marihuanę. Nasi południowi sąsiedzi Czesi zalegalizowali marihuanę. Podpowiem: zrobił to rząd centroprawicowy, chadecki. Nie tych naukowców od słupków poparcia, tylko tych od marihuany, od konopi, od uzależnień. Trzeba to zalegalizować, bo nie legalizując, doprowadzacie do rozwoju mafii. No niestety. To jest malutki kroczek, oczywiście w dobrym kierunku, ale mikrokroczek, a my potrzebujemy dużych kroków. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, o godz. 12.10 przejdziemy do głosowania.

Wznawiam obrady. Obecnie przystąpimy, proszę państwa, do stwierdzenia kworum. W związku z tym bardzo proszę wszystkich państwa posłów o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu potwierdzenia udziału w posiedzeniu.

To są ministrowie, którzy są posłami.

Stwierdzam kworum. Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który poddam pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku oznaczać będzie, że Sejm, zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu, skierował ten projekt ustawy do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w celu rozpatrzenia. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 1989, zechce nacisnąć

Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował ten projekt ustawy do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w celu rozpatrzenia. Na podstawie art. 73 ust. 2 regulaminu Sejmu wyznaczam termin przedstawienia sprawozdania komisji umożliwiający rozpatrzenie go na bieżącym posiedzeniu Sejmu.

Przechodzimy do zadawania pytań.

Bardzo proszę. Jest pan poseł?

Panie Ministrze!

Co autorzy mieli na myśli, jeżeli chodzi o środki techniczne, które uniemożliwiają wejście osób nieuprawnionych? Dziękuję. Bardzo proszę, pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Chciałbym zapytać wnioskodawców o wyliczenie rentowności upraw, na które nakładacie państwo jednak dość drastyczne wymogi. Chciałbym wiedzieć, jaki zakładacie szacunkowy koszt nadzoru fizycznego, administracyjnego oraz elektronicznego w przeliczeniu na 1 kg zbiorów. Pytam o to w trosce o osoby, o których traktuje ten dokument. Czy po spełnieniu wszystkich wymogów koszt finalny produktu nie będzie na tyle wysoki, że mimo dopuszczalnych upraw i legalnej produkcji w kraju osoby chore lub ich rodziny będą nadal zmuszone do nielegalnego importu z zagranicy ze względu na ceny, które, jak się obawiam, mogą być strasznie wysokie? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Joanna Fabisiak, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze!

Bardzo proszę, pani poseł Beata Maciejewska, Lewica.

Dlaczego nie wprowadził pan zmian, które proponował Parlamentarny Zespół ds. Legalizacji Marihuany? Dlaczego nie wprowadził pan możliwości refundacji leków chociażby dla dzieci z padaczką lekooporną czy osób z glejakiem mózgu? Dlaczego nie wprowadził pan możliwości produkowania marihuany medycznej pod obostrzeniami przez przedsiębiorców w Polsce, którzy mogliby na tym zarabiać? Dlaczego nie wprowadził pan możliwości szkoleń dla medyków, żeby wiedzieli, na czym polegają dobroczynne skutki używania marihuany medycznej? Dziękuję. Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Czy jest pan poseł? Pan poseł Aleksander Miszalski, Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo! Wiemy, że konopie to rośliny o ogromnym potencjale medycznym, które znajdują zastosowanie tam, gdzie inne leki nie dają rady, np. nowotwory, padaczka lekooporna czy bóle chroniczne. Dziś sprowadza się ją z Izraela, z Kanady, z Hiszpanii, co niestety znacznie zwiększa jej koszty i ogranicza jej dostępność. Polscy rolnicy nie są mniej uczciwi niż ci z Kanady, z Izraela i mogliby też uczciwie uprawiać konopie w Polsce. Proponujecie jednak, by zajmowały się tym tylko instytuty badawcze, stąd moje pytanie: Dlaczego? Jak długo potrwa proces ich uzyskiwania? Z jakimi dużymi kosztami będzie wiązało się objęcie tych upraw monitoringiem? Jak to wpłynie na koszt wytworzenia tych leków przy tych obostrzeniach? Czy będzie możliwy również eksport i co z refundacjami? Dziękuję bardzo.

Pani Marszałek! Pani Minister! Panie Ministrze!

Tylko tutaj mamy instytut rolniczy, który będzie produkował surowiec farmaceutyczny, i Główny Inspektorat Farmaceutyczny, który dopuszcza surowiec farmaceutyczny do sprzedaży w aptekach. I moje pytanie do pana ministra: Czy już nawiązano ten kontakt, relację, czy główny inspektor farmaceutyczny powiedział, jakie wymagania będą musiały być spełnione przez ten surowiec farmaceutyczny, który będzie produkował instytut rolniczy, aby w ciągu kilku miesięcy pierwsze partie konopi medycznych były w aptekach? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica. Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! Przedmiotem ustawy jest zezwolenie na prowadzenie uprawy i zbioru konopi innych niż włókniste przez państwowy instytut badawczy, co w efekcie ma doprowadzić m.in. do obniżenia ceny marihuany medycznej w aptekach. Czy uprawa tych konopi w Polsce przez instytut badawczy rzeczywiście doprowadzi przy tych uwarunkowaniach formalnoprawnych, które są zawarte w ustawie, jeśli chodzi o uprawy i wszystkie kwestie nadzorcze, do obniżki cen marihuany medycznej w aptekach?

Dziękuję.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Występuję z podobną tezą jak socjaliści, co jest rzeczą zdumiewającą.

Rząd by tego nie przepuścił. Ponieważ każda ustawa powinna być opatrzona klauzulą, ile na tym stracimy, to chciałbym wiedzieć, ile budżet państwa polskiego straci na odrzuceniu tej ustawy. Mam nadzieję, że wnioskodawcy uzupełnią ten projekt tą niesłychanie ważną liczbą, bo chcielibyśmy wiedzieć, ile stracimy na odrzuceniu tej ustawy. Dziękuję za uwagę. Bardzo proszę, pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! To dobry krok.

Ile będą kosztowały nadzór i monitorowanie? Chciałam zapytać, w jakiej wysokości te przychody wyszacowaliście i o ile tańsze będą leki, jeżeli państwo nie będziecie przyjmowali refundacji. Chodzi o to, że dzisiaj marihuana medyczna sprowadzana jest z Kanady i z innych państw, a jeżeli będziemy mieć swoją, to o ile tańsze będą leki? Pan poseł Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Nawet jeśli coś państwo robicie w dobrym kierunku, to właśnie w tak beznadziejny sposób, że później znowu trzeba będzie po was sprzątać. Widzę, że niestety państwo z prawej strony poczuwają się do roli stróżów monopolu, jaki producenci alkoholu wywalczyli sobie na rynku substancji psychoaktywnych, i strzeżecie zazdrośnie przywileju trucia Polaków za pomocą jednej, wybranej substancji, którą właśnie jest alkohol i którą można w zasadzie ładować w klienta bez ograniczeń. Z kolei strzeżecie tego nie bezinteresownie, bo w alkoholu większość ceny to przecież podatki, to zrzutka na wasz rząd, więc właściwie to kto alkoholu nie pije, jak mówił poeta, ten jest wywrotowcem i świadomie uszczuplającym dochody państwa bezideowcem. Jeśli w imię pilnowania wpływów ze sprzedaży swojego ulubionego narkotyku ograniczacie możliwości produkcji leków, ustanawiając znowu jakiś idiotyczny monopol, to jesteście po prostu cynicznymi hipokrytami. Dziękuję bardzo. Pan poseł Artur Dziambor, Konfederacja. Ta ustawa jest oczywiście ustawą techniczną i takim mikrokroczkiem, co już tutaj dzisiaj było wspomniane, a więc nie mam co do niej wątpliwości i środowisko partii KORWiN na pewno poprze tę ustawę. Szanowni Państwo! Ale za każdym razem, gdy ten temat wchodzi do dyskusji publicznej, jedna rzecz mnie bardzo mocno męczy. Ta rzecz to hipokryzja. Otóż żyjemy w świecie, w którym każdy, kto chce, ma dostęp do kogoś, kto jest w stanie załatwić jakimiś krokami, jakimiś ścieżkami marihuanę, czy to medyczną, czy to rekreacyjną, to nie ma żadnego znaczenia.

Powinniście robić gigantyczne kroki i nauczyć się na tym zarabiać.

Panie Ministrze! Są rejestry producentów, są wskazane w ustawie instytucje, które wyrażają zgodę na produkcję, a potem okazuje się, że państwo cały czas mówicie o jednej firmie. Pan poseł Sachajko nie ukrywa, że chodzi o instytut roślin włóknistych z Poznania.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pana ministra.

Dlaczego państwo nie chcieliście się zgodzić na poprawkę, którą zgłosiłyśmy z posłanką Zawiszą na posiedzeniu Komisji Zdrowia? Wydaje mi się że polscy pacjenci mają prawo wiedzieć, dlaczego oni, osoby, które chorują na padaczkę lekooporną, pacjenci onkologiczni, którzy mierzą się z olbrzymim cierpieniem, są pozbawieni wsparcia w postaci refundacji ze strony państwa. Jeżeli pan minister nie odpowie dzisiaj na sali, bardzo proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję, pani poseł. Bardzo proszę, pani poseł Dorota Niedziela, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! W czerwcu zeszłego roku starałam się kupić marihuanę medyczną. Powiem państwu, jak wygląda ta droga przez mękę. Żaden lekarz w przychodni nie chce wypisać recepty.

Dlaczego to nie jest refundowane? I następne pytanie, bardzo ważne. Panie pośle Sachajko, to będzie pusta ustawa. Wie pan dlaczego?

czyli podstawowa rzecz, którą musi dysponować każdy instytut, który będzie ją produkował. Tylko jeden Instytut Farmaceutyczny w Warszawie. Jeśli tego nie mają, nigdy nie będą produkować surowca. Muszą być monitorowane ilości substancji, użycie pestycydów i wiele innych rzeczy. Badania użycia pestycydów wykonuje się w Niemczech, bo w Polsce żadne laboratorium tego nie robi.

Dziękuję bardzo, pani poseł.

Mam przyjaciela, który ma syna z porażeniem mózgowym, dziecko, które choruje również na padaczkę lekooporną, czyli taką, która nie reaguje na standardowe leki koncernów farmaceutycznych. To dziecko ma kilkanaście bolesnych ataków epilepsji dziennie. I mnóstwo cierpienia, bo najpierw w ogóle tego nie wolno było stosować, później niby można było, ale ciężko było znaleźć lekarza, bo nie ma procedur medycznych, a jak już znalazł się lekarz, to później był wielokrotnie problem z dostaniem tego, bo nie wolno u nas hodować. To jest skandal, to jest ogrom cierpienia, który wynika z tego, że ubzduraliście sobie jako politycy, że macie prawo mówić, co człowiek może jeść, palić, jakie leki może przyjmować. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Andrzej Rozenek, PPS. Pani Marszałek! Niedzieli się zwracam - nie będzie potrzebna żadna refundacja, jeżeli pozwolimy ludziom po prostu uprawiać krzaczki w domu. Nie byłoby tego problemu. Rzeczywiście cena jest zaporowa, ale to wynika z monopolu. Główny Inspektorat Farmaceutyczny będzie wydawał zezwolenia instytutom. Chciałbym o te instytuty zapytać, panie ministrze.

Ludzie, co wy robicie? Pozwólcie wszystkim Polakom uprawiać to, co chcą. Jeżeli nie chcą, to niech jej nie uprawiają, prosta sprawa. To jest niepoważne. Dziękuję bardzo. Pan poseł Piotr Borys, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo!

Ostatnie pytanie, pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Bardzo uprzejmie dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Drugie pytanie dotyczy konkretnych przypadków i osób, które chcą czy będą chciały korzystać.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia pana ministra Macieja Miłkowskiego o odpowiedź na pytania. Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo!

My takiej informacji od instytutu nie otrzymaliśmy.

Widzimy, że jest to możliwe wyłącznie w ramach programu lekowego, ponieważ tam dokładnie można dookreślić wskazania refundacyjne, komu ten lek najbardziej pomaga i w jakim dokładnie wskazaniu medycznym. I uważamy, że jest to zasadne, w szczególności po wejściu w życie tej ustawy. Po zarejestrowaniu surowca i po przygotowaniu produktu leczniczego z tego surowca na pewno będziemy starali się wzmocnić, przyspieszyć to, jeśli nie będzie wcześniej takiego wniosku. Rozmawiałem z kilkoma firmami, które mają rozeznanie na rynku produkcji tych leków, z firmami, które produkują w Polsce i które na dzień dzisiejszy mają rozeznanie już na rynku światowym w zakresie tego surowca i są zainteresowane również zakupieniem z produkcji polskiej, o czym mówiliśmy, instytutu nadzorowanego przez ministra rolnictwa. Tak jak państwo mówią, na dzień dzisiejszy jest to jeden instytut, ale instytutów nadzorowanych przez ministra rolnictwa jest więcej.

Jeśli chodzi o pytania pana posła Korwin-Mikkego, ile straci budżet, to tak jak już mówiłem, uważamy, że to jest dobry produkt, dobra działalność właśnie dla instytutów naukowo-badawczych i to jest ewidentnie produkcja, która może przynieść istotne dochody tym instytutom. Instytuty pokrywają swoje koszty z przychodów, w związku z tym uważamy, że to bardzo dobry kierunek, żeby te instytuty mogły mieć znacząco wyższą rentowność przeznaczoną na rozwój swojej działalności podstawowej, działalności badawczo-rozwojowej. Pytanie, dlaczego to mają być instytuty nadzorowane przez ministra rolnictwa.

I tutaj nie planujemy, tak jak państwo posłowie, żeby wychodzić z organizacji, żeby móc realizować wszystko, co nam się podoba.

Bardzo proszę, sprawozdawca komisji pan poseł Jarosław Sachajko. Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Dziękuję serdecznie wszystkim za tę debatę. Było kilka pytań merytorycznych np. o to, jaka jest rentowność upraw. Ja oczywiście w trakcie procedowania pytałem panią minister Gembicką o tę rentowność. Instytut zadeklarował, i mam nadzieję, że pani minister tego dopilnuje, aby gram był nie droższy niż 30 zł, czyli to i tak jest dwukrotnie taniej niż w tej chwili za sprowadzany. Ale niestety mieliśmy tutaj bardzo emocjonalne, wprost pełne hipokryzji wystąpienie pani poseł Maciejewskiej, która powiedziała, że jest to beznadziejna ustawa i zapytała, dlaczego się nie wprowadzi wielkiego poluzowania. Chciałbym wszystkim państwu nas oglądającym powiedzieć, że to właśnie Lewica miała wiele lat, żeby to zrobić i tego nie zrobiła.

Czy coś z tego zrobiła?

Tylko tak walczyli, że było coraz gorzej. Przyszła prawica, pojawił się Kukiz’15 i mamy ustawę, ustawę bardzo dobrą, tak jak powiedziałem, która za chwilę doprowadzi do tego, że będziemy mieć polskie konopie w aptekach, tanie konopie. Pani poseł tutaj mówiła o tym, że jest przeciwko pacjentom.

Cytuję. Pani poseł mówi: Dlaczego nie ma możliwości refundacji? Pan minister - jakby pani poseł pozostała na posiedzeniu komisji - powiedział, że będzie refundacja, ale leków, które później powstaną. I wszystkich chciałem poinformować, że zgłasza się kilka firm, polskich firm farmaceutycznych, które chcą pozyskać ten surowiec z instytutu, który ma bardzo duże doświadczenie w uprawie, i chcą produkować leki, które później będą refundowane.

Ja pani poseł chciałem powiedzieć, że lekarze wiedzą, co z tym robić, lekarze są wyszkoleni i o tym też była mowa w komisji, trzeba było tylko pozostać i posłuchać, a nie tutaj rozdzierać szaty. A więc jeżeli państwo mają takiego swojego lekarza rodzinnego, a każdy lekarz rodzinny może wypisać receptę na konopie medyczne, to trzeba zmienić lekarza. A instytut będzie miał zezwolenie. Te dwie instytucje się dogadają i będzie to w dostępnej cenie. Pan poseł Korwin pytał, ile stracimy jako ludzie, jeżeli ta ustawa nie będzie wprowadzona.

Tu chodzi o to, że ludzie potrzebują leku, a nie, tak jak mówi to słynne hasło, sadzić, palić, zalegalizować.

I dzięki temu jesteśmy na pierwszym miejscu pod względem spożycia alkoholu.

Bardzo proszę. Ad vocem tego, co powiedział pan poseł Sachajko, który żali się tutaj z mównicy, że ktoś krytykuje jego kadłubkowy projekt - nie odpowiedział w zasadzie na żadne z moich pytań i wydaje się, że nie ma zielonego pojęcia o tym. jaka jest dzisiaj sytuacja pacjentów i jaka jest dzisiaj rzeczywiście wiedza medyków na temat marihuany medycznej.

Ta ustawa, którą dzisiaj proponuje związany z PiS-em poseł Sachajko, który mógł znacznie więcej wynegocjować, nie wprowadza. Bardzo proszę, pan poseł Sachajko i zamykamy. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Ja nie chcę się osobiście odnosić do tego, co pani poseł powiedziała, ale ona obraża polskich lekarzy. Moja żona jest lekarzem i panią zapewniam, że ona wie, jak wypisywać, i wie, jak stosować. To, o czym pani mówi, to jest.

Kończymy. Są tysiące lekarzy, szanowni państwo, którzy wypisują. I powiedziałem to z tej mównicy. Jeżeli jest jakikolwiek lekarz, który nie chce państwu wypisać we wskazaniach medycznych konopi medycznych, to trzeba zmienić lekarza. Kupuje się to na czarnym rynku, bo właśnie ci szarlatani mówią, że mają taniej, że ich jest lepsza. Lepsza to jest właśnie ta kupiona w aptece, o której wiemy, co w niej jest, bo ta kupiona na czarnym rynku jest hodowana w różnych warunkach, jest o niewiadomym składzie, a bardzo często są tam dodawane inne środki psychotropowe. Obrażanie posłów, którzy przygotowali tę ustawę, mówienie, że ona jest kadłubkowa. Szanowni państwo, czas pokaże. Czas pokaże, jak Lewica we wszystkim się myli, próbując dyskredytować wszystkich innych. Ostatnia rzecz, o której mówiła pani poseł. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druki nr 1611 i 1977) Proszę pana posła Jarosława Sachajkę o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie komisji rolnictwa w sprawie druku nr 1611, czyli poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. W posiedzeniu z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczyła pani sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka. W trakcie posiedzenia zgłoszono 15 poprawek. Poprawka 1. wprowadza zmiany w celu uwzględnienia możliwości przetwarzania maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych z upraw własnych we własnym zakresie. Poprawki 12. i 13. nadają właściwemu dyrektorowi oddziału KOWR uprawnienia do przeprowadzania kontroli upraw oraz zbiorów maku lub konopi włóknistych, ponadto nadają uprawnienia do wydania nakazu zniszczenia uprawy lub plonów maku lub konopi włóknistych. Poprawka 14. doprecyzowuje, w jakich okolicznościach stosowane są przepisy karne w związku z naruszeniem ustawy.

Komisja w głosowaniu przyjęła wniosek o uchwalenie przez Sejm projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 34 głosami, przy jednym głosie przeciw i jednym głosie wstrzymującym się. Bardzo dziękuję, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Bardzo proszę, pierwszy głos zabierze pan poseł Krzysztof Szulowski, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa autorstwa, podobnie jak w przypadku poprzedniej ustawy, posłów Kukiz’15 i Prawa i Sprawiedliwości, druk nr 1611. Projekt ustawy dotyczy uprawy konopi włóknistych i maku. Ma na celu wsparcie tych upraw przy jednoczesnym, co dla nas oczywiste, uwzględnieniu nadrzędnego celu, jakim jest przeciwdziałanie narkomanii. Dotychczasowe rozwiązania wpływały ograniczająco na powierzchnię uprawy i możliwości rozwoju krajowej biogospodarki. Mówiąc o ograniczeniach, należy mieć na względzie chociażby to, że każdy producent oraz skupujący mak lub konopie składa corocznie wniosek, wraz z całą dokumentacją, do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast lub marszałków województw o wydanie decyzji upoważniającej do uprawy lub skupu maku lub konopi włóknistych. A jeszcze włączony do tego jest sejmik województwa odpowiedzialny za określenie powierzchni upraw maku i konopi. Zaproponowane rozwiązania, które ułatwią podmiotom prowadzenie działalności w zakresie uprawy oraz skupu maku lub konopi włóknistych, to: szybka rejestracja i prowadzenie zbioru danych (rejestr) w jednym miejscu; brak obowiązku corocznego gromadzenia i składania dokumentacji przez podmiot; brak obowiązku uzyskiwania corocznego zezwolenia; brak ograniczenia powierzchniowego, regionalnego i czasowego w wydawanym zezwoleniu w zakresie uprawy i skupu; rozszerzenie przeznaczenia i celów, na jakie może być wykorzystywany mak czy konopie włókniste. Te cele to cele energetyczne, weterynaryjne, paszowe, związane z materiałami kompozytowymi, rekultywacja i remediacja gruntów, cele pszczelarskie i nawozowe - tu jako naturalne środki ochrony roślin. Proponuje się również, aby mak i konopie włókniste mogły być uprawiane także na potrzeby własne, na potrzeby naukowo-badawcze oraz z przeznaczeniem do hodowli nowych odmian maku i konopi włóknistych.

Ma dotyczyć to także monitorowania skupu oraz prowadzenia rejestru podmiotów, które uprawiają mak lub konopie włókniste. Ten rejestr będzie prowadzony przez dyrektora oddziału terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres podmiotu. Oczywiście bardzo istotne jest to, że projekt ustawy zabezpiecza środki w celu przeciwdziałania narkomanii: rejestr podmiotów skupujących prowadzony przez KOWR dotyczy tylko tych pierwszych podmiotów skupujących mak lub konopie włókniste (to ułatwi kontrole prowadzone przez KOWR lub policję), wnioski o wpis do rejestru będą zawierać precyzyjne informacje, takie jak: dane wnioskodawcy, określenie podmiotów, z którymi zostały zawarte umowy na dostarczanie maku lub konopi włóknistych, albo oświadczenie o wykorzystaniu lub przetwarzaniu tych roślin we własnym zakresie na potrzeby lub cele określone w ustawie, w przypadku uprawy maku - oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą, informacje o odmianie maku lub konopi, planowanej powierzchni i lokalizacji uprawy. Wprowadza się przepis obligujący KOWR do przeprowadzania kontroli producentów i skupujących mak lub konopie włókniste, kontroli informacji zawartych we wnioskach oraz kontroli upraw maku i konopi włóknistych. Przed faktycznym rozpoczęciem uprawy opinię dotyczącą sposobu jej zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych będzie sporządzać policja, a zezwolenie będzie wydawać główny inspektor farmaceutyczny. Przewidziano również system kar, m.in. za przekazanie nieprawdziwych informacji we wniosku o wpis do rejestru, nieprzekazanie informacji o zmianie danych w stosunku do tych zawartych we wniosku. W przypadku uprawy maku lub konopi włóknistych bez wpisu do rejestru KOWR wydaje decyzję o zniszczeniu uprawy, w określonych sytuacjach powiadamia policję. Uważamy proponowany projekt za dobry, stwarzający perspektywę rozwoju biogospodarki w oparciu o zwiększoną podaż krajowego surowca konopi włóknistych i maku, a jednocześnie, tak jak powiedziałem, bezpieczny. Dlatego klub Prawa i Sprawiedliwości wyraża poparcie dla projektu. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pani poseł Anna Wojciechowska, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko klubu Koalicji Obywatelskiej dotyczące przedmiotowej ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Ustawa ma na celu wsparcie rozwoju upraw maku i konopi włóknistych przy jednoczesnym uwzględnieniu przeciwdziałania narkomanii.

To m.in. szybka rejestracja, rejestr wszystkich danych w jednym miejscu, brak ograniczenia powierzchniowego; tylko w przypadku uprawy na potrzeby własne jest ograniczenie do 10 a rocznie. Monitorowanie, rejestr i kontrolowanie upraw zostają przypisane Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Obecnie zajmują się tym urzędy marszałkowskie i gminy.

W sposób właściwy zabezpiecza się uprawy przed niepożądanymi odbiorcami.

Koszt obsługi tego przedsięwzięcia to 964 tys. rocznie - ale powstanie 12 nowych etatów - oraz 100 tys. rocznie na obsługę informatyczną. Klub Koalicji Obywatelskiej poprze ten projekt ustawy. Bardzo proszę, pani poseł Beata Maciejewska, Lewica. Wysoka Izbo! Konopie w Polsce służą do kryminalizowania ludzi.

Druga rzecz to ogromne obostrzenia, które dotychczas obowiązywały: konieczność rejestrowania się i corocznego otrzymywania zgód. Parlamentarny Zespół ds. Legalizacji Marihuany opracował, podobnie jak poseł Sachajko, projekt, który ma ułatwiać rolnikom uprawę konopi włóknistych. Przypomnę państwu, że w grudniu ub.r. powstała Polska Izba Konopi, zrzeszająca ponad 100 producentów konopi, założona z inicjatywy stowarzyszenia Wolne Konopie.

Szkoda, że nie dotyczy to także marihuany medycznej.

Chodzi o to, żeby rolnicy podobnie jak pacjenci mogli korzystać z dóbr konopi, czy to konopi włóknistych, czy to konopi innych niż włókniste. Jako Lewica będziemy składać poprawki do tego projektu dotyczące drobnych rzeczy, drobnych spraw: konieczności podłączania faktur, tego, w jaki sposób mają być prowadzone kontrole, dlatego że uznajemy, że ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii powinna być w jak najmniejszym stopniu stosowana wobec upraw konopi włóknistych.

Jako Lewica poprzemy ten projekt ustawy. W tym momencie składam na ręce pani marszałek nasze poprawki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Projekt dotyczy wsparcia rozwoju upraw maku i konopi włóknistych przy jednoczesnym uwzględnieniu nadrzędnego celu, jakim jest przeciwdziałanie narkomanii. W projekcie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zaproponowano rozwiązania, które ułatwią podmiotom prowadzenie działalności w zakresie uprawy oraz skupu maku lub konopi włóknistych przez: szybką rejestrację i prowadzenie zbioru danych w jednym miejscu, brak obowiązku corocznego gromadzenia i składania dokumentacji przez podmiot, brak obowiązku uzyskiwania corocznego zezwolenia, brak ograniczenia powierzchniowego, regionalnego i czasowego w wydawanym zezwoleniu w zakresie uprawy i skupu, rozszerzenie przeznaczenia i celów, do jakich może być wykorzystany mak czy konopie włókniste. Proponowana nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii będzie zawierała również dwie definicje, dotyczące producenta maku i producenta konopi włóknistych, określające podmioty prowadzące działalność w tym zakresie. Proponuje się również rozszerzyć cele, dla których mają być prowadzone uprawy maku i konopi włóknistych, m.in. o cele energetyczne, weterynaryjne, paszowe, dotyczące materiałów kompozytowych, rekultywacji i remediacji gruntów, pszczelarskie, nawozowe - jako naturalnych środków ochrony roślin. Dodatkowo mak i konopie włókniste będą mogły być uprawiane także na potrzeby własne, potrzeby naukowo-badawcze oraz z przeznaczeniem do hodowli nowych odmian maku i konopi włóknistych. Procedowana ustawa przenosi obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z samorządów właściwych ze względu na miejsce położenia uprawy na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Jednocześnie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uwzględnia wprowadzenie rejestru podmiotów, które uprawiają mak lub konopie włókniste. Proponuje się, aby rejestr ten był prowadzony przez dyrektora oddziału terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres podmiotu. Chciałbym zwrócić uwagę na przepisy, które ograniczają rolę samorządów w kreowaniu ich lokalnej gospodarki. Oczywiście rozumiemy fakt, że wprowadzenie rejestru ma duży wpływ na dążenie do przeciwdziałania narkomanii oraz ułatwienie kontroli upraw w takim stopniu, aby stwierdzić, czy uprawiana roślina jest legalna, a produkt roślinny uzyskany z tej uprawy jest bezpieczny. Właśnie takie obawy dotyczące omawianego projektu ustawy wystosowała naczelna rada pielęgniarek i położonych, która obawia się, że nowelizacja spowoduje łatwiejszy dostęp do marihuany, zwiększenie spożycia, wystąpienie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych oraz bezwzględne zwiększenie nakładów ze środków publicznych na leczenie i rehabilitację osób uzależnionych oraz dodatkowe obciążenia podmiotów leczniczych. Jednocześnie popieramy stanowisko samorządu wielkopolskiego, który stwierdził, że pojawienie się konieczności wprowadzenia nowego rozwiązania w postaci rejestru skupiającego wszystkich uczestników rynku w zakresie uprawy i skupu maku i konopi przy obecnym stopniu wykorzystania rozwiązań informatycznych jest problemem, który można rozwiązać w prosty sposób - przez utworzenie platformy wymiany informacji, w której uczestniczyć mogą zarówno samorządy, jak i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Trzeba jednak przyznać, że jeśli chodzi o główną materię, ten projekt ustawy ma dobre założenia i może w wymierny sposób rozwinąć polskie rolnictwo. Dowodem niech będzie fakt, że Krajowa Rada Izb Rolniczych w trakcie opiniowania tego projektu złożyła zaledwie jedną poprawkę, kosmetyczną, polegającą na dodaniu kilku słów do brzmienia ust. 2 w art. 45 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W oczywisty sposób zyska na tym rolnictwo poprzez zwiększenie możliwości uprawy zarówno konopi, jak i maku. W tym wypadku największy zysk będą mieli konsumenci dzięki zwiększeniu podaży na konopie i mak. Co za tym idzie, nastąpi spadek cen produktów wykonywanych z tychże roślin. Na końcu zyska również państwo, które pobierać będzie opłaty za wpis do rejestru, a także zyska na innych daninach w postaci podatków. Klub parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe poprze tę ustawę.

I bardzo proszę, pan poseł Michał

Wysoka Izbo! Jako Konfederacja popieramy ułatwienie prowadzenia plantacji konopi i maku przy jednoczesnej kontroli mającej na celu przeciwdziałanie narkomanii. Jednocześnie popieramy ułatwienie, wsparcie dla osób produkujących choćby konopie włókniste, gdyż mają one szerokie zastosowanie w przemyśle i mogą realnie przyczynić się do poprawienia sytuacji budżetowej naszego kraju. Jak wiemy, ten rząd bardzo lubi nowe podatki, więc nie dziwię się, że to wprowadza. Jesteśmy zwolennikami wspierania krajowych producentów, ułatwiania zakładania własnych hodowli i przedsiębiorstw oraz uniezależniania się od rynków zagranicznych, bo wiemy, że polskie rolnictwo ma z tym problem już od lat, nie tylko w tej jednej branży. Wykorzystywanie konopi w celach medycznych jest i bezpieczne, i skuteczne w leczeniu wielu dolegliwości, więc w interesie chorych jest to, aby dostęp do leków stworzonych z tych substancji był jak najszerszy, aby było to jak najskuteczniejsze, właśnie dla Polaków. Podsumowując, powiem, że wsparcie upraw konopi i maku z zastrzeżeniem, że będą to wyroby medyczne i przemysłowe, jest jak najbardziej do zaakceptowania. Proszę, pan poseł Artur Dziambor, Konfederacja.

W poprzednim wystąpieniu troszkę wspomniałem o tym, jak mógłby wyglądać cały rynek konopi i upraw tych konopi, ale jestem zadowolony, że chociaż jakieś małe kroki są podejmowane, i myślę, że zadowolona z tego będzie również druga strona sceny politycznej, która, myślę, od zawsze do tego nawoływała. Szanowni Państwo!

Do skorzystania z tego rynku zachęcamy, zachęcamy jako wolnorynkowcy, jako ludzie, którzy uważają, że rynek powinien być wolny, że jeżeli ktoś chce coś kupić, to powinien móc to kupić, a ktoś inny powinien to wyprodukować dla tego kogoś, kto chce kupić. Zacznijmy od tego, które jest tutaj. Bardzo dobrze, ale mam nadzieję, że na tym dyskusja się nie skończy. My to poprzemy i mamy nadzieję, że państwo będziecie bardziej chętni do dyskusji o rozszerzaniu tej listy w przyszłości, a my z kolei zapewniamy, że postaramy się zrobić wszystko, żeby obciążenia podatkowe w odniesieniu do wspomnianego przeze mnie przed chwilą wolnego handlu były jak najniższe dla przedsiębiorcy i dla klienta. Bardzo proszę, pani poseł Joanna Mucha, Polska 2050. Pani Marszałek!

Najważniejsze, co trzeba powiedzieć o tym projekcie, to to, że Polska troszeczkę dzięki temu projektowi normalnieje. Normalnieje z punktu widzenia tych, którzy uprawiają mak i konopie włókniste.

Normalnieje wreszcie z punktu widzenia urzędów państwowych, które będą mogły zajmować się tym, co bardzo potrzebne, a nie tym, co było zupełnie bezsensowne, bo ten projekt ustawy daje szansę na to, żeby szybko rejestrować te uprawy, żeby prowadzić w jednym miejscu rejestr tych upraw. To do tej pory nie było praktykowane, a to na pewno jest potrzebne.

I to jest, wydaje mi się, bardzo istotne w tej ustawie. Mniejsze koszty po stronie państwa, jednocześnie poprawa skuteczności systemu nadzoru nad tymi uprawami. Oczywiście jest to niewielki krok do przodu, ale jednak krok do przodu. Z tego powodu będziemy oczywiście popierać tę ustawę.

Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Kukiz’15 - Demokracja Bezpośrednia mam zaszczyt przedstawić stanowisko koła w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. W poprzedniej kadencji mieliśmy również podobny projekt. Ustawa odpowiada na wszystkie problemy, jakie rolnicy zgłaszali. Przepraszam, nie na wszystkie, bo jeszcze mam poprawki, jeszcze jest jedna rzecz do poprawy.

Dobrze, że w tym kierunku idziemy.

Niech państwo sprawdzą projekt ustawy. Projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, gdzie właśnie z rolników zrobiono przestępców, został wprowadzony w 2005 r. właśnie przez Lewicę. I to jest ta hipokryzja, że w tej chwili Lewica rozdziera szaty, że krzywda się dzieje, a sama tę krzywdę zrobiła. Dlatego jeszcze raz dziękuję pani minister oraz wszystkim posłom, którzy uczciwie, bez emocji pracowali nad poprawą tego wszystkiego, co przez lata - powtórzę: od czasów Lewicy - zepsuto.

Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zgłosić się do zadania pytania? Jeżeli nie, zamykam listę. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Rafał Adamczyk, Lewica. Pani Minister! W uzasadnieniu ustawy czytamy: Zakłada się, że projektowane zmiany mogą przyczynić się do poprawy sytuacji budżetu państwa w związku ze zwiększeniem wpływów podatkowych związanych z rozwojem biogospodarki w oparciu o zwiększoną podaż krajowego surowca konopi włóknistych i maku, uwzględniając także dodatkowy wydatek na stworzenie i utrzymanie systemu monitorowania upraw przez KOWR i oszczędności związane z przeniesieniem zadań w tym zakresie z administracji samorządowej. Bardzo bym prosił o informację, w jakiej wysokości będą to wpływy. Czy macie państwo to oszacowane? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Wysoka Izbo! Mając na względzie dobro oraz bezpieczeństwo osób prowadzących działalność w obrębie produkcji konopi, chciałbym zapytać, co należy rozumieć pod pojęciem ˝pomieszczenie˝ oraz ˝środek transportu zabezpieczony przed kradzieżą produktu˝ Od osoby prowadzącej działalność wymagane jest wydanie takiego oświadczenia, więc ona ponosi za to odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność karną. Jaki organ i na jakiej podstawie może w Polsce wydawać decyzje o tym, czy pomieszczenie lub pojazdy we właściwy sposób zabezpieczają produkty przed kradzieżą? Czy Policja, na wniosek plantatora konopi, wystawi mu takie zaświadczenie? Jeśli nie Policja, to poproszę o wskazanie właściwej instytucji, która takie zaświadczenie będzie wystawiała. Uprzejmie proszę o odpowiedź na piśmie. Pani poseł Joanna Fabisiak, Koalicja Obywatelska.

Pani Minister! Przez całe wieki Polska była producentem maku. Nasi sąsiedzi kupowali go, eksportowaliśmy go, kupowali od nas. To niedobry kierunek i chyba niemądry. Produkujemy mak, bo chcielibyśmy kupować go właśnie w polskich sklepach. Zastanawiam się także, czy to rzeczywiście jest zasadne, aby Policja wydawała zgodę, Policja kontrolowała. Toć Policja ma całkiem inne zadania, wydaje mi się, że dużo ważniejsze. Czy naprawdę należy ich na pola makowe kierować? Uważam, że nie. Bardzo słuszny jest kierunek ustawy, aby wreszcie zająć się normalną produkcją, normalnych roślin, które są do Polski jak gdyby przypisane. Natomiast sama droga. Czy istotnie jest ona drogą rozwoju tej formy rolnictwa, czy raczej dalszego ograniczenia, choć może nie ma już penalizacji? Dziękuję bardzo. Pan poseł Jarosław Rzepa, Koalicja Polska. Wysoka Izbo! Pani Minister!

To jest wielkie pytanie, panie ministrze. Ten, który to zapisał - jaką miał intencję, jeśli chodzi o dopuszczenie tego do uprawy na powierzchni 100 a? Panie pośle, wiem, że pan zmienił miejsce siedzenia i teraz ta centralizacja panu się też podoba. Ale myślę, że żaden marszałek nigdy nie pozwolił sobie na to, żeby ograniczyć jakąkolwiek powierzchnię ze względu na wnioskowanie przez poszczególnych producentów, za pośrednictwem gmin, jeśli chodzi o uprawę maku czy konopi. Myślę, że ten pomysł na zmianę jest niedobry. Uważam, że powinniśmy zostać przy tym systemie, który był, czyli wójtowie, marszałkowie województwa. Pani poseł Marta Wcisło. Pani poseł Anna Wojciechowska, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo!

Czy nie jest to sztuczne i nieuzasadnione rozbudowanie kadr KOWR-u? Dziękuję bardzo.

Panie Człowieku Wolności Kaczyński! Wysoka Izbo! Ułatwienia w produkcji konopi włóknistych to krok w dobrą stronę, więc proponuję, abyśmy poszli za ciosem i odmrozili także projekt o marihuanie rekreacyjnej. Według naukowców marihuana w mniejszym stopniu uzależnia niż alkohol czy nikotyna.

Wskażcie choć jeden racjonalny argument, dlaczego nie zalegalizować marihuany. Bo argumenty za są na wyciągnięcie ręki. Koniec dilowania wśród młodzieży, przemycania ton tej substancji przez granicę, ograniczenie działań mafii narkotykowej. Państwo może monitorować, ile osób bierze marihuanę. Policjanci mogą zająć się ważniejszymi sprawami, podatnik nie płaci za odsiadkę palaczy i sądy nie sądzą ich. W USA - 200 tys. nowych miejsc pracy (Dzwonek), w Polsce - niech to będzie nawet 20, przydałoby się. Na koniec petarda - ostatnie zdanie, pani marszałek - przy objęciu marihuany akcyzą i stawką VAT, jak przy artykułach tytoniowych, to dodatkowe nawet 9 mld zł do budżetu. Dziękuję, pani poseł. Pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. W procedowanej ustawie należy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Uprawa konopi i maku w naszym kraju jest obecnie pod kontrolą.

Nowe rozwiązania znoszą te wymogi. Aby móc uprawiać konopie czy mak, trzeba będzie jedynie zgłosić wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ustawa jest dużym ułatwieniem dla producentów rolnych. Jak do zawartego w tytule przeciwdziałania narkomanii ma się to, że jednocześnie planuje się dodanie przepisu, który pozwoli na zwiększenie zawartości substancji halucynogennej w suszu? Bardzo proszę, pan poseł Jarosław Sachajko, Kukiz’15.

Wysoka Izbo!

Nie jest powiedziane, że tylko ten instytut będzie to uprawiał.

Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Pani Minister! Wysoka Izbo! Dosyć rygorystyczne są przepisy, jeżeli chodzi o jednostki, które mogą podjąć tę działalność.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski. Szanowna Pani Minister!

Jakie będą koszty dla budżetu państwa związane z wprowadzeniem dodatkowych zadań dla KOWR?

Jeśli tak, to jakie są w tej sprawie przywidywania? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jan Duda, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Przeniesienie kontroli i rejestracji upraw konopi i maku na poziom oddziałów KOWR jest bardzo dobrym rozwiązaniem.

Czy KOWR jest przygotowany? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo!

To nie jest prawda. To się odnosi do całości.

Uprawa konopi włóknistych na potrzeby własne może być realizowana na cele włókiennicze, energetyczne, spożywcze, weterynaryjne, paszowe itd., które określone są w ustawie. My wprowadzamy taką możliwość. Co pozwoli nam też na kontrolę rynku. Ale jednocześnie nie wprowadza się też ograniczenia powierzchni upraw z przeznaczeniem na inne potrzeby czy cele. Jeżeli chodzi o kwestię samorządów, tutaj stoimy na stanowisku, że jednak te dotychczasowe wymogi dotyczące właśnie opinii urzędów marszałkowskich to jest po prostu niepotrzebne utrudnienie, to dodatkowe formalności. Nie chcemy, żeby była taka sytuacja, że to mogłoby opóźniać rolnikom uzyskanie wpisu.

Tak jak powiedział pan poseł Sachajko, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadzoruje 12 instytutów.

Z tych informacji uzyskanych z instytutu wiemy, że jest on w stanie wypełnić to zapotrzebowanie. Jesteśmy w stałym kontakcie roboczym także z GIF-em.

Jeżeli chodzi o koszty obsługi nowego mechanizmu, to ok. 864 tys. rocznie będzie przeznaczone na etaty, na osoby, które będą odpowiedzialne za te kwestie, oraz ok. 100 tys. rocznie na koszty prowadzenia obsługi systemu informatycznego, a jednorazowy koszt budowy systemu informatycznego wyniesie ok. 440 tys. zł. Bardzo dziękuję. I bardzo proszę sprawozdawcę komisji pana posła Jarosława Sachajkę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję ponownie za te pytania, które były dużo bardziej merytoryczne niż poprzednio. Ogólnie można by było powiedzieć, odpowiadając na dużą część pytań, że po prostu w tej chwili tą ustawą likwidujemy te absurdalne zapisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które powstały za rządów lewicy. To trzeba przypominać: lewica spowodowała to, że z rolników można było robić producentów narkotyków. Pan Szopiński pytał właśnie o pomieszczenia i pojazdy, pytał, kto będzie wydawał zaświadczenia.

To w ustawie jest napisane, tylko w drugą stronę, dlatego może pan poseł tego nie zrozumiał. No właśnie nie. Właśnie o to chodzi, że teraz policja i różne inne instytucje nie będą ścigały rolników, tylko zajmą się ściganiem przestępców. Pan poseł Jarosław Rzepa mówił o tym, że im bliżej rolnika, czyli marszałek i wójt, tym lepiej. No, panie pośle, proszę zapytać o to rolników, bo właśnie ten marszałek i ten wójt bardzo często wydawali zgody po czasie, gdy minął czas, kiedy rolnik mógł to zasiać. Bo właśnie była taka inercja tych urzędów, że one traktowały rolników, przepraszam, per noga: tak, kiedyś się mu to wyda. Teraz będzie to centralnie dla całej Polski i będzie zwykła rejestracja, a nie pozwolenia. Wiem, że wielu polityków jest przyzwyczajonych do tego, że rolnik czy obywatel musi chodzić na kolanach do urzędu i o wszystko prosić. Tu nie ma o co prosić. Tu trzeba tylko poinformować, a nie prosić, tak jak do tej pory bywało. No, to zależy od urzędników gminy i urzędników urzędu marszałkowskiego. Te etaty mogą być zagospodarowane dużo lepiej niż w tej chwili, nie tak żeby wydawać puste kwitki pozwalające na uprawę rośliny takiej, która jest podobna do tytoniu, do marchewki, do pszenicy. Ci urzędnicy mogą się skupić na zupełnie innej pracy, tak żeby Polacy nie czekali tygodniami na zgody i na różne inne dokumenty z urzędów gmin. No właśnie gminy zyskają, bo jeżeli gmina ma mieć zysk z tego, że za każdy papierek będzie brała od obywateli pieniądze, że będzie nakazywała o wszystko pytać i za to brać pieniądze, jeżeli tak byśmy patrzyli, to rzeczywiście gminy stracą, tylko gminy nie są od tego, żeby grabić swoich obywateli, tylko są od tego, żeby im ułatwiać życie. I my tą ustawą ułatwiamy życie rolnikom i Polakom. A jednocześnie dzięki temu, że będzie większa produkcja, że będzie przetwórstwo lokalne, gminy zyskają, zyskają właśnie na tym, czyli nie będą. Dużo gmin w tej chwili mówi o tym, że są biedne, bo są tylko rolnicze. No tak, dlatego tutaj pozwalamy zarabiać nie tylko na wytwarzaniu produktów podstawowych, ale dajemy rolnikom również możliwość przetwarzania i sprzedaży, czego do tej pory nie było.

Bardzo proszę, 1 minuta.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister!

Być może, że te dwa projekty bardzo bliskie w jakiś sposób nałożyły się, że to było w pierwszym, ale w moim odczuciu, i bardzo proszę o wyjaśnienie tej kwestii, czy Policja będzie interweniowała wtedy, kiedy będą nieprawidłowości, ale w całej procedurze dopuszczania do produkcji nie będzie miała udziału i potrzeby zajmowania się tą sprawą. Jeszcze pan poseł chce sprostować. Tak? Pani Minister! Pani Poseł! Dziękuję za to doprecyzowanie. Przy konopiach siewnych Policja nie będzie miała żadnego udziału. Powtórzę, konopie siewne to jest taka sama roślina jak tytoń, pszenica czy buraki, więc tutaj Policja nie bierze żadnego udziału. Proszę zauważyć, że tam jest tylko opinia Policji, która nie jest wiążąca. Jeszcze jedna rzecz w tym projekcie jest zapisana - i tu Policja nie widziała problemu - żeby w taki sposób było to zapisane, że Policja będzie miała tylko 30 dni na wydanie tej opinii, czyli nie będziemy czekać nie wiadomo ile.

Czyli idziemy naprawdę do przodu z tymi dwoma projektami, tak żeby gospodarka się rozwijała, żeby pacjenci mieli dostęp do konopi i żeby rolnicy mogli zarabiać na konopiach siewnych. Dziękuję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1515 i 1845) Bardzo proszę pana posła Janusza Kowalskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Mam ogromny zaszczyt i honor przedstawić sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z druku nr 1515. Jest to, szanowni państwo, tym bardziej dla mnie honor i zaszczyt, że jako pełnomocnik rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa inicjowałem i byłem koordynatorem przygotowania tego projektu ustawy, który rzeczywiście w sposób merytoryczny został przez komisję i podkomisję rozpatrzony. W tym momencie przypomnę, jak te prace w ramach komisji i podkomisji wyglądały. 1 października Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu i projekt ustawy, projekt tej największej od 20 lat reformy Kodeksu spółek handlowych, został skierowany do rozpatrzenia w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. 14 października Komisja Nadzwyczajna również odrzuciła wniosek o odrzucenie projektu i skierowała go do prac w podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego kierowanej przez pana posła Grzegorza Lorka. Na kilku posiedzeniach podkomisji w dniach 8, 9, 23 listopada oraz 7 grudnia szczegółowo omówiliśmy przedłożony projekt. Projekt, który jest projektem rządowym, ale sytuacja z tym projektem jest nadzwyczajna, bo został on przygotowany przez zespół kilkudziesięciu ekspertów, przez stronę społeczną. 15 grudnia Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach przyjęła projekt w brzmieniu przedkładanym Wysokiej Izbie.

Tym bardziej że w pracach podkomisji i komisji uczestniczyli członkowie Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego utworzonej w Ministerstwie Aktywów Państwowych, znakomici profesorowie, znakomici prawnicy, jest to dla mnie wielki honor, aby najważniejszych autorów tej kodyfikacji, którzy również brali udział w toku dyskusji, w tym miejscu, w Sejmie Rzeczypospolitej, wymienić. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Aktywów Państwowych, to szefem Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, największej od 20 lat reformy, był i jest pan premier Jacek Sasin, ja miałem zaszczyt być, i jestem nadal, wiceprzewodniczącym tej komisji. Na poziomie ministerstwa prace koordynowało dwoje dyrektorów, dr Filip Ostrowski, obecny na sali, i pani dyrektor Izabela Wojtyczka.

Szczególnie chcę podziękować i podkreślić rolę pana prof. Andrzeja Szumańskiego, współautora Kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 r. W pracach nad tym projektem, ale również w pracach podkomisji i komisji brali udział m.in. dr Radosław Kwaśnicki, prof. Piotr Pinior, prof. Mirosław Pawełczyk, dr Rafał Kos, mec. Jan Ginko, pani prof. Dominika Wajda, pan Mateusz Berger, pan Jakub Modrzejewski, pan prof. Piotr Niczyporuk, mec. Radosław Potrzeszcz, mec. Przemysław Ciszak.

W tym miejscu chcę podkreślić osobiste zaangażowanie pana ministra Zbigniewa Ziobry, który koordynował przyjęcie tego projektu na poziomie rządowym razem z panem premierem Jackiem Sasinem, oraz rolę pana dyrektora Artura Grajewskiego z Ministerstwa Sprawiedliwości, sędziego Piotra Perczyńskiego, a także bardzo ważną rolę pana wiceministra Marka Niedużaka, byłego wiceministra rozwoju i prezesa Prokuratorii Generalnej (Dzwonek) pana Mariusza Haładyja oraz Luizy Modzelewskiej. Jeżeli mogę szybciutko wymienić najważniejsze zmiany w toku.

Jeżeli chodzi o drugą grupę poprawek, dotyczyła ona regulacji grup spółek.

Oczywiście musi posiadać, ale unikamy ryzyka uznania czynności z art. 58 za nieważną. Jeżeli chodzi o czwartą zmianę, dotyczyła ona tego, że wszystkie dokumenty, które są wydawane wspólnikowi, wydawane są w formie zgodnej z jego żądaniem. Piąta zmiana dotyczyła kwestii zawierania umów o zarządzanie i przekazywanie zysku spółki.

Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Bardzo proszę. Szanowni Państwo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec przygotowanej przez ponad 60 ekspertów w Ministerstwie Aktywów Państwowych przy współpracy z innymi ministerstwami reformy Kodeksu spółek handlowych.

Z punktu widzenia Kodeksu spółek handlowych bardzo ważne jest wprowadzenie prawa grup spółek po raz pierwszy - art. 7, który nie wypełniał swojej roli, zostaje zniesiony. Polska wzorem innych państw, takich jak Niemcy, Słowenia, Czechy czy Portugalia, będzie miała bardzo nowoczesne przepisy prawa handlowego w obszarze korporacyjnym, w obszarze dotyczącym zarządzania grupami spółek. Przyjęliśmy również założenia dotyczące fundamentalnej reformy funkcjonowania rady nadzorczej. Rady nadzorcze, szanowni państwo, w rozumieniu projektu reformy k.s.h. staną się nie tylko organem kontrolnym, ale przede wszystkim partnerem w spółce, przez co zostanie wyeliminowanych bardzo wiele patologii.

Ta kwestia musiała być w sposób precyzyjny uregulowana.

Niby rzecz oczywista, ale jednak orzeczenia niektórych sądów sprawiały ogromne ryzyko dla wielu przedsiębiorców.

Wysłanych było kilkaset zaproszeń do udziału w konsultacjach społecznych, i do kancelarii prawniczych, i na wszystkie uniwersytety. Ten projekt jest projektem zbiorowym kilkudziesięciu prawników. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za udział w tych pracach. Jeżeli chodzi o Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, to pozwolę sobie, pani marszałek, złożyć kilka poprawek.

Bardzo proszę, pani poseł Barbara Dolniak, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Tak chwaliliście Polski Ład i co? Totalny bubel. Wymaga poprawek, zmian. Przedsiębiorcy z każdej strony mówią, że trzeba go zawiesić. I mamy kolejny bubel prawny: projekt dotyczący Kodeksu spółek handlowych. Jego koncepcja jest sprzeczna z praktyką obrotu gospodarczego, co zagraża bezpieczeństwu tego obrotu. 75% tego projektu wymagało poprawek merytorycznych czy legislacyjnych, czy też merytoryczno-legislacyjnych.

Uwagi zgłaszane przez kluby opozycyjne, jak i podmioty zewnętrzne, np. Krajową Radę Radców Prawnych czy Konfederację Lewiatan, nie zostały uwzględnione. Brak było odpowiedzi na zadawane pytania, a konsultacje przed wniesieniem projektu trwały zaledwie czterdzieści parę dni, i to latem. Nie przeprowadzono również żadnej analizy, a przynajmniej nie przedstawiono jej treści, mimo że zwracaliśmy się o przedstawienie takiej analizy. Proces tworzenia prawa nie może być eksperymentem. Prawo spółek musi się zmieniać, ale nie w oderwaniu od gospodarki i jej zidentyfikowanych i udowodnionych potrzeb.

I tak np. Krajowa Rada Radców Prawnych podnosi, że w zakresie regulacji prawa grup spółek projekt należy ocenić jednoznacznie negatywnie. Negatywną opinię tego projektu wyraziły również Naczelna Rada Adwokacka czy Krajowa Rada Komornicza. Projekt nie zyskał również poparcia Konfederacji Lewiatan. Jak skrajnie niedobry jest to projekt, wynika chociażby z opinii Sądu Najwyższego, który wskazał: Można mieć poważne obawy, że ewentualne wejście w życie projektowanych przepisów nie uporządkuje należycie prawa koncernowego, a może sprzyjać powstaniu jeszcze większej liczby wątpliwości, zróżnicowaniu sytuacji prawnej rozmaitych faktycznie istniejących grup spółek, a przez to godzić też w stabilność i bezpieczeństwo obrotu prawnego. Czy można sobie wyobrazić gorszą opinię? Chyba nie. Wiele zastrzeżeń przedstawiło również Biuro Analiz Sejmowych. W ocenie znawców prawa handlowego, którzy zajmują się tym prawem zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, takich jak prof. Tomasz Siemiątkowski, prof. Michał Romanowski i prof. Andrzej Kidyba, projekt nie nadaje się do procedowania ani stosowania w praktyce. Wady projektu są tak fundamentalne, że dyskwalifikują go w całości.

Tyle było chwalenia, tyle wygłaszania pozytywnych opinii, a gdy projekt wszedł w życie, okazał się totalnym bublem. Uratujmy przynajmniej w tej części polskich przedsiębiorców i uchrońmy ich przed tak złym projektem ustawy. uwzględniając zarówno wnioski przedsiębiorców, praktykę, jak i orzecznictwo, które wykształciło się przez wiele lat. Inaczej będziemy mieli kolejny przykład bubla prawnego, który natychmiast trzeba będzie zmienić. Takie tworzenie prawa nie służy przedsiębiorczości, wręcz tę przedsiębiorczość zabija. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Dariusz Wieczorek, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rzeczywiście usłyszeliśmy tutaj od posła sprawozdawcy, inicjatora tego przedsięwzięcia, dużo ciepłych słów o tym, jak ten projekt ustawy był procedowany.

Jedno z drugim raczej nie ma nic wspólnego. Myślę, że analizując ten projekt ustawy, co do jednej rzeczy możemy być przekonani: rzeczywiście potrzeba rozwiązań, które będą jasne, klarowne i czytelne, jeżeli chodzi o możliwość tworzenia holdingów i grup kapitałowych. Ale niestety ten projekt tego problemu nie rozwiązuje, a w naszej ocenie, w ocenie klubu Lewicy, jeszcze wprowadza dużo niejasnych zapisów, które później w jakichś procesach mogą być rozstrzygane przez sądy. I wcale nie upraszcza to tworzenia tych holdingów, nie upraszcza to funkcjonowania grup i spółek zależnych, a wręcz w naszej ocenie to utrudnia. Zastanawialiśmy się, skąd wprowadzanie tego typu zmian nagle w Kodeksie spółek handlowych. I niestety mamy nieodparte wrażenie, że właściwie chodzi tutaj o jeden zapis, który został, mówiąc krótko, ładnie obudowany wieloma różnymi innymi artykułami. A ten zapis brzmi mniej więcej tak, że: członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny. Czyli, mówiąc krótko, dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją taką, że za te wszystkie błędne decyzje w tych wszystkich spółkach, w których Skarb Państwa ma udziały, za te środki finansowe wydatkowane bez sensu, już nie chcę mówić o tych różnych instytucjach, dzisiaj nikt na podstawie tego zapisu nie będzie ponosił odpowiedzialności, bo znajdziecie zawsze jakąś opinię, że trzeba było Ostrołękę budować, znajdziecie opinię, że trzeba było drukować karty do głosowania, znajdziecie opinię odnoszącą się do szeregu innych waszych przedsięwzięć, na które wydaliście setki milionów złotych, i w tym momencie te zarządy nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności. I myślę, że o to głównie w tej ustawie chodzi. Natomiast ustawa oczywiście wprowadza różne inne zapisy i, jeszcze raz chcę podkreślić, wcale nie ułatwia tworzenia holdingów, natomiast wprowadza bardzo niejasne zapisy, chociażby w kwestii dotyczącej spółek dominujących i poleceń wiążących. Do końca w tej ustawie nie jest określone, jeżeli chodzi o spółkę dominującą, który organ może wydawać polecenia - rada nadzorcza, zarząd, nie wiadomo. Jeżeli chodzi o te polecenia wiążące, to rodzi się pytanie, jak one mają być wydawane - ustnie, pisemnie, uchwałami, więc tutaj może doprowadzać to do bardzo dużego bałaganu. Rzecz kolejna to oczywiście kwestie dotyczące możliwości zmian umów spółek zależnych czy tych spółek, które są w grupie, przez spółkę dominującą. To jest kwestia również tych wszystkich odmów wykonania tych poleceń, kwestia rad nadzorczych, bo tutaj wprowadzamy zapis dotyczący tego, że rady nadzorcze będą mogły na koszt spółki wynajmować własnych audytorów. Znowu może być naturalny konflikt między radą nadzorczą a zarządem, czy rada działa w interesie spółki. Do tego są zapisy mówiące o tym, że w radzie nadzorczej nie musi być 100% członków, żeby jakiś nowy punkt wprowadzić, również mamy sposób głosowania wprowadzany bezwzględną większością głosów, czyli generalnie tych głosów wstrzymujących się tutaj nie uznaje. Tak że na tym etapie niestety jest to projekt, który nie może być poparty, bo on nie rozwiązuje tych problemów, o których pan poseł Kowalski mówił. Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Paszyk, Koalicja Polska. Bardzo dziękuję. Panie i Panowie Posłowie! Panie Pośle Wnioskodawco! W biznesie wśród przedsiębiorców bardzo dużą popularnością cieszy się takie powiedzenie wyrażające oczekiwanie od władzy publicznej, aby ona nie przeszkadzała lub aby jak najmniej przeszkadzała. Wówczas ta działalność będzie możliwa do prowadzenia w sposób nieskrępowany i efektywny. Ta ustawa niestety trochę wbrew temu oczekiwaniu wyrażonemu i powtarzanemu bardzo często przez przedstawicieli biznesu niestety przeczy i to jest jej największy problem. Niestety zgadzając się z tymi krytycznymi spostrzeżeniami, które zostały przez przedmówców wyrażone, trzeba powiedzieć, że to nie jest taki projekt, który byłby oczekiwany. Najbardziej chyba miażdżąca, ale też konstruktywna, merytoryczna krytyka tego projektu została złożona przez pana prof. Michała Romanowskiego, który bardzo dobitnie prezentuje też dorobek i praktykę, którą w spółkach dotychczas przygotowano, opracowano, ale też obala niestety ten mit, który pan poseł wnioskodawca próbował zbudować, jakoby właśnie tych rozwiązań oczekiwano. Oczekiwano czegoś znacznie bardziej ambitnego, na miarę czasów i potrzeb. Tu też zgadzam się z tymi opiniami, które zostały wyrażone, że niestety nie odbierając dobrych chęci, szczerych intencji, które być może przyświecały przy tworzeniu projektu, nad którym procedujemy, trzeba powiedzieć, że jest to trochę znowuż próba uszczęśliwiania Polaków na siłę.

Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Krzysztof Bosak, Konfederacja.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Dobrze, że debatujemy nad nowelizacją prawa gospodarczego. Dziwi sytuacja, że w czasach tak szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej wszyscy tutaj chwalimy to, że pierwszy raz od 20 lat nowelizujemy Kodeks spółek handlowych. Wydaje mi się, że powinniśmy nad takimi przepisami pochylać się częściej. Jeżeli coś nie domaga - tutaj mój przedmówca mówił, iż zmiany powinny iść dalej, powinny dotykać większej liczby kwestii - to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten dialog był bardziej ożywiony i żeby Sejm częściej zajmował się tym prawem, aczkolwiek przede wszystkim mając na względzie stabilizację reguł działania biznesu w Polsce i to, żeby te przepisy były proste, przewidywalne i żeby nie wprowadzać zmianami niepotrzebnego zamieszania. Jeżeli chodzi o przedłożoną nowelizację, to wypowiadałem się już na poprzednich posiedzeniach Sejmu w tej sprawie. Te przepisy można podzielić na dwie grupy. Po pierwsze, są przepisy ułatwiające zarządzanie grupą spółek poprzez spółkę dominującą w związku z realizacją wspólnej strategii gospodarczej grupy. Trudno takiej zmiany nie pochwalić, bowiem rzeczywiście we współczesnym życiu gospodarczym często działa się nie poprzez pojedynczy podmiot, ale właśnie poprzez bardziej złożone grupy kapitałowe. Druga grupa przepisów to przepisy zapewniające ochronę wierzycieli spółek zależnych i ich wspólników lub ich akcjonariuszy, a także członków organów spółki zależnej i spółki dominującej.

Mamy do czynienia z przepisami, które chwaliłem - w zasadzie chyba mogę tak uczciwie powiedzieć - podczas swojego poprzedniego wystąpienia w tej sprawie, a więc ze wzmocnieniem rady nadzorczej.

Rada będzie mogła badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji jej stanu majątkowego, żądać od zarządu, prokurentów przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących sytuacji spółki. Mamy też związane z nadużyciami przepisy, które mają utrudnić osobom skazanym pełnienie jakichkolwiek funkcji, a więc zakaz sprawowania funkcji w zarządzie, w radach nadzorczych, w komisji rewizyjnej, bycia prokurentem czy likwidatorem spółki przez osoby skazane za bierne i czynne łapownictwo, płatną protekcję oraz nadużywanie uprawnień funkcjonariusza publicznego. Na pochwałę zasługuje (Dzwonek) w mojej ocenie także wprowadzenie zasady biznesowej oceny sytuacji, która ma zabezpieczyć osoby pozostające w organach spółek przed bezzasadnym posądzaniem o działanie na szkodę spółek. Znamy wiele takich spraw, gdy osoby podejmujące ryzyko biznesowe były później poddawane różnego rodzaju postępowaniom czy po prostu skazywane za działanie na szkodę spółek, a była to normalna działalność gospodarcza. To krok w kierunku normalności i przybliżenia przepisów do współczesnych realiów życia gospodarczego. Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Bardzo uprzejmie dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050 w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw po przedstawieniu sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Prace nad przedłożonym przez rząd projektem trwały rzeczywiście długo. Niemniej jednak niestety czas prac nie przełożył się na zasadniczą zmianę w przypadku tego projektu ustawy.

Gdyby przyjęto te wszystkie uwagi, być może projekt zasługiwałby dzisiaj na inną ocenę. Niestety zmuszeni jesteśmy wystawić ocenę negatywną, która w naszym przypadku będzie oznaczała wniosek o odrzucenie projektu ustawy w drugim czytaniu.

W żaden sposób nie sprzyja to czytelności nadzoru, nie sprzyja to jakości sprawowanego nadzoru. W związku z tym, że w czasie 3 minut nie ma możliwości przedstawienia kompleksowej oceny, pozostanie wypowiedziane to, co już powiedziałem, a na ręce pani marszałek składam wniosek o odrzucenie tego projektu ustawy. Dziękuję, panie pośle. Szanowni Państwo! Przechodzimy do pytań. Wyznaczam czas - 1 minuta. Pierwsze pytanie zadaje pan poseł Rafał Adamczyk, klub Lewica. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dostrzegł w świetle projektowanych przepisów ryzyko polegające na tym, że członkowie organów krajowego podmiotu nadzorowanego nie będą ponosić odpowiedzialności za wykonanie wiążącego polecenia otrzymanego od akcjonariusza większościowego, a narzędzia służące egzekwowaniu odpowiedzialności takiego akcjonariusza przez organ nadzoru są ograniczone. Bardzo bym prosił o pisemne odniesienie się do tych uwag Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę. W polskim ustawodawstwie przyjęło się, że pomimo wspólnych zasad funkcjonowania jednoosobowe spółki prawa handlowego traktowane są gorzej niż pozostałe. Ta ustawa niestety wpisuje się w ten trend, dlatego mam pytanie. Dlaczego w przypadku grupy spółek spółka zależna z kapitałem zgromadzonym w rękach jednego udziałowca może domagać się naprawienia szkody wyrządzonej w wyniku decyzji spółki dominującej wyłącznie w sytuacji, gdy szkoda ta doprowadzi do jej niewypłacalności, natomiast pozostałym spółkom przysługuje naprawa szkód w dużo szerszym zakresie? Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Bardzo proszę, panie pośle.

Wysoka Izbo! Prawo do własności jest fundamentalne, stanowi podstawę funkcjonowania społeczeństwa. Bez szacunku do prawa własności nie jest możliwe kształtowanie odpowiedzialności za dobro wspólne. Ano dlatego, że ten projekt przewiduje możliwość przymusowego wykupu udziałów lub akcji: 25% - w spółkach zamkniętych, 5% - w spółkach publicznych. Instytucja squeeze out jest oczywiście obecna dzisiaj w K.s.h., ale dotyczy mikroskopijnych akcjonariuszy. Specjaliści określają ich jako plankton albo ziarna piasku na pustyni, ale 1/4 akcjonariatu, a chociażby nawet 5% udziałowców to nie jest plankton, to nie są ziarnka piasku, to jest grupa, której przysługują bardzo silne uprawnienia korporacyjne. Dziękuję. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym zadać pytanie przedstawicielom wnioskodawców, panu posłowi. Dotyczy ono kosztów związanych z możliwością zatrudniania przez rady nadzorcze w ramach prowadzonej działalności audytorów i innych osób, które mają pomóc radzie nadzorczej wykonywać czynności nadzorcze.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Pani poseł Iwona Maria Kozłowska, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! To, że jest to zły projekt, powiedziała już pani poseł Barbara Dolniak, natomiast chciałabym odnieść się do przepisu art. 18 ust. 2, który rozszerza wachlarz przestępstw pozbawiających możliwości pełnienia funkcji członka zarządu spółki. Przedsiębiorcy, z którymi konsultowałam te zmiany, wskazywali wyraźnie na przypadki, kiedy osoby skazane za oszustwa, przywłaszczenia, niezgłoszenie upadłości spółki we właściwym czasie nadal, bez konsekwencji, piastują swe funkcje w zarządach.

Jak pokazuje praktyka, dotychczasowe działania sądu są nieskuteczne, a skazany przestępca nadal jest członkiem zarządu. W opracowaniu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dr Tomasz Czułowski wyraźnie o tym mówi. Bardzo proszę o zadanie pytania. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Procedowana ustawa obfituje w wiele negatywnych rozwiązań. Można odnieść wrażenie, że autorzy projektu pokazują, że nie rozumieją fundamentu prawa spółek. Czy można źle zarządzać własną spółką, a winą obarczać zarząd innej spółki? Już niedługo, po wejściu w życie planowanej nowelizacji ustawy takie sytuacje mogą stać się codziennością. Ponadto w ustawie planuje się wprowadzić nadrzędność interesu grupy spółek nad własnym interesem spółki zależnej. To według was są dobre zmiany? Jaką rolę w spółce zależnej będzie odgrywał zarząd, który będzie pozbawiony częściowo, a może i całkowicie, wpływu na prowadzenie spółki? Pani poseł Barbara Dolniak, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! W trakcie prac w komisji czy podkomisji zadawaliśmy szereg pytań. Czy interes spółki zależnej jest oderwany od interesu spółki matki? Co w przypadku, gdy spółka matka ma 100% udziału w spółce zależnej? Kto będzie rozstrzygał, jaki jest interes spółki zależnej? Czy spółka matka ma też odrębny interes? Kto go definiuje? Czy jeżeli grupa spółek nie zdecyduje się utworzyć grupy, to oznacza to, że nie ma grupy spółek i nie może być realizowana strategia grupy? Te i wiele innych pytań pozostało bez odpowiedzi. Bez odpowiedzi pozostał też nasz wniosek o przedstawienie analizy tego projektu. Skoro nie przedstawiliście jej państwo do tej pory, to oznacza tyle, że tej analizy w ogóle nie wykonaliście. Dziękuję. Proszę bardzo. Wysoka Izbo!

Dlaczego chcecie wprowadzać zmiany w tak ważnym obszarze spółek handlowych, nie konsultując tego w ogóle z przedstawicielami tychże właśnie spółek? Nie uwzględniliście praktycznie żadnych poprawek zgłoszonych przez organizacje zrzeszające podmioty, których ta ustawa dotyczy. Znowu wsadzacie kij w dobrze funkcjonujące tryby polskiej gospodarki. Chcecie to wszystko popsuć. Wprowadzacie np. odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej, jeżeli szkoda ta powstała w następstwie wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia spółki dominującej oraz jeżeli egzekucja przeciwko spółce zależnej należącej do grupy spółek okaże się bezskuteczna. Przełóżmy to na język polityki. To może spróbujmy to przełożyć tak: wprowadzimy odpowiedzialność partii dominującej (Dzwonek) za szkody wyrządzone przez koalicjanta. Rachunek wystawiony za szkody wyrządzone przez pana Ziobrę, pana Kowalskiego i innych spółkodawców pójdzie w miliardy. Chcecie zmian? Rozmawiajcie o nich. Nie chcecie rozmawiać? Odejdźcie z polityki. Pan poseł Dariusz Stefaniuk, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze! Chciałem zadać pytanie, bo opozycja cały czas podważa ten projekt, jakoby nie było konsultacji społecznych, mój przedmówca również do tego nawiązywał, chciałbym zapytać posła wnioskodawcę oraz pana ministra o konsultacje społeczne, jak one wyglądały, jak się odbywały, jak były szerokie.

Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Istotą spółki prawa handlowego jest to, że odpowiada jedynie przed prawem i odpowiada przed właścicielem, ale przed właścicielem odpowiada w sposób ograniczony. Właściciel może zmienić zarząd, może zmienić radę nadzorczą, ale nie może wtrącać się w bieżące zarządzanie spółki, bo musi być czytelna odpowiedzialność. Taka sytuacja niczego nie uzdrowi, tylko skomplikuje wszystko, co jest możliwe w zarządzaniu. Może o to chodzi. Załóżmy, że są nadużycia i są błędne decyzje. Kto może stwierdzić, że niższa instancja wykonała polecenie i nie jest winna temu, że jest ono źle wydane albo nie w odpowiedni sposób? I wreszcie kompetencje ludzi, którzy to robią. Dzisiaj niestety jest niekompetencja. Dziękuję. Pan poseł Grzegorz Lorek, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie! Ten wątek odpowiedzialności opozycji też by był ciekawy, być może kiedyś będziemy go rozważać.

Czy ciężar nie został przechylony w inną stronę? Pytanie jest bardzo proste: Czy rada nadzorcza nie uzyskuje nadmiaru kompetencji w stosunku do zarządu?

Też bym prosił o wyjaśnienie w tym zakresie. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Są oczywiście dwa modele prowadzenia działalności gospodarczej: albo polskie prawo będzie jasne i czytelne dla przedsiębiorców, albo będzie nieczytelne. I teraz pytanie: Czy w Polsce potrzebne jest prawo grup spółek? Czy takie grupy spółek jak Grupa RMF, Grupa Żywiec, Axel Springer, nawet Grupa Agora, nie mówiąc oczywiście o Grupie PKN Orlen czy grupie PGE, potrzebują nowoczesnego prawa gospodarczego prywatnego w obszarze grup spółek? Otóż tak. Powiem więcej. Przywoływany przez opozycję, przez Platformę Obywatelską pan prof. Michał Romanowski o tym właśnie pisał w marcu 2008 r., o tym, jak archaiczny jest art. 7 Kodeksu spółek handlowych i że trzeba stworzyć grupy spółek. Dzisiaj się oczywiście z tego wycofał, ponieważ jego kancelaria zarabia na tzw. kodeksie grup kapitałowych i łupi albo łupiła przedsiębiorców, uznając, że niepotrzebne jest prawo, tylko wystarczą jego usługi.

A wy chcecie powiedzieć temu ˝nie˝ Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę. Wysoka Izbo!

Wysoka Izbo! Gdyby poszukać definicji totalniactwa, to ta definicja znalazłaby odzwierciedlenie w zachowaniu polityków Platformy Obywatelskiej w kontekście pracy nad tą ustawą. Przejąłem tę ustawę po panu ministrze Januszu Kowalskim, któremu bardzo serdecznie chciałbym podziękować za stworzenie tak profesjonalnego zespołu, który opracował ten projekt. W momencie kiedy dołączyłem do prac legislacyjnych nad tą ustawą, byłem świadkiem czegoś niespotykanego: krytyka w 100%. Państwo przychodziliście na pierwsze posiedzenie komisji nadzwyczajnej, później na pierwsze posiedzenie podkomisji, a następnie bojkotowaliście całkowicie prace. Co za tym idzie, nie zgłosiliście żadnych poprawek merytorycznych do tego projektu.

Została powołana specjalna komisja w Ministerstwie Aktywów Państwowych przez wspomnianego już premiera Jacka Sasina i przez pana ministra Janusza Kowalskiego. Na początku zadajmy sobie pytanie, dlaczego ta ustawa jest potrzebna. 62% ankietowanych wypowiedziało się pozytywnie o normatywnym uregulowaniu prawa grup spółek. Natomiast w odniesieniu do wzmocnienia kompetencji rad nadzorczych pozytywne stanowisko wyraziło 55% ankietowanych, a jedynie 38% - negatywne.

Również chcę podziękować panu dyrektorowi dr. Filipowi Ostrowskiemu. Udział w tym brali również członkowie organów oraz dyrektorzy spółek dużych, WIG20, i osoby, które miały reprezentować mniejszych przedsiębiorców, takie jak zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorców czy członek władz Lewiatana, również osoby znajdujące się w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa, w spółkach prywatnych. Tak że ten projekt został skonsultowany z szerokim gronem eksperckim. Państwo tutaj oczywiście mówicie, że ustawa jest niechlujna, że jest niepotrzebna. Po co ta ustawa, skoro mamy orzecznictwo? Jeśli pomieszamy wątki, pomieszamy systemy prawne i zapomnimy, że w Polsce jednak obowiązuje system prawa stanowionego, a nie system prawa precedensowego czy zwyczajowego, to może tak. A nawet gdyby przyjąć, że jest prawo zwyczajowe, precedensowe, to kto to widział, żeby traktować orzeczenia referendarzy jako wyznacznik tego, jak mają funkcjonować grupy spółek? Te przepisy, które przygotowało Ministerstwo Aktywów Państwowych, są więc niezwykle ważne. Jeden dotyczył właśnie definicji grup spółek, która została w ramach prac parlamentarnych zmodyfikowana. A drugi zarzut dotyczył wykluczenia spółek publicznych. Sugerowałbym politykom Platformy Obywatelskiej, aby się zdecydowali, czy są za tym, aby te regulacje jeszcze szerzej szły, jeszcze większy zakres spółek obejmowały, czy jednak węższy.

Od tego jest praca parlamentarna i to pokazuje otwartość Ministerstwa Aktywów Państwowych na to, aby ten projekt udoskonalać. My naprawdę byliśmy otwarci na to. Przypomnę: ani jednej poprawki nie złożyliście w ramach prac parlamentarnych. Rozwiązanie, które funkcjonuje, to jest kalka rozwiązania niemieckiego. Tutaj próbuje się dopisywać, dodawać jakąś interpretację polityczną do rozwiązań, które wspierają przedsiębiorców, dają im narzędzia, aby mogli podejmować, tak jak to w biznesie, czasami ryzykowne decyzje. Muszą mieć świadomość, że jeśli nie popełnią przestępstwa, to nie spotka ich odpowiedzialność karna.

Dziękuję, panie ministrze. Pani poseł Barbara Dolniak w trybie sprostowania. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Gdyby pan rzetelnie przysłuchiwał się dyskusji na posiedzeniach komisji i podkomisji, to doskonale by pan wiedział, że rzeczywistość była zupełnie inna: brak odpowiedzi na pytania, skracanie czasu wypowiedzi. Nawet zaproszonym gościom limitowano czas, mimo że pracowaliśmy nad trudnym projektem. Wskazywaliśmy na istotne niedociągnięcia tego projektu. Nikt nie brał tego pod uwagę. Mało tego, nie brano pod uwagę również przedstawicieli instytucji, którzy uczestniczyli w posiedzeniach komisji czy podkomisji. To wszystko pokazuje, że państwo przedstawiacie rzeczywistość w zupełnie innym świetle. Jakby tego było mało, dołączyliście państwo do poprawek - mówimy o Kodeksie spółek handlowych, proszę państwa -mnóstwo poprawek dotyczących innych ustaw (Dzwonek), np. ustaw o Krajowym Zasobie Nieruchomości, o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, o utworzeniu polskiej agencji rozwoju, o działach administracji rządowej. Jeśli chodzi o przebieg prac parlamentarnych, to najlepszym podsumowaniem będzie państwa zachowanie. Zbojkotowaliście posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej w momencie, kiedy pan minister Kowalski i inni członkowie przypomnieli, że prof. Romanowski, który teraz tak gorliwie krytykuje z wami ten projekt, sam był członkiem komisji do spraw nadzoru właścicielskiego. Gdy pokazaliśmy dowód, to wywołało to reakcję alergiczną i zamknęło wam usta. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Bardzo serdecznie dziękuję za tak profesjonalne podsumowanie ze strony pana ministra Jana Kanthaka. Serdecznie mu dziękuję za dokończenie prac nad tą reformą.

Dzisiaj na tej sali obniżyła pani poziom emocji. Jestem przekonany, że pan Dariusz Wieczorek chciałby głosować za tym projektem, ale z politycznych powodów nie może. Jego kolega, pan mecenas Szejna, naprawdę bardzo wspierał nas w czasie posiedzenia podkomisji i w czasie prac komisji. Bardzo merytoryczne było pytanie pana posła Suchonia.

Przerywa wiele niepotrzebnych procesów, które w tej chwili toczą się w Polsce. Chcę jasno powiedzieć, że po tej dyskusji - to jest moja ocena - mam nieodparte wrażenie, że jedyną osobą z opozycji, która przeczytała, za co bardzo serdecznie dziękuję, projekt ustawy, który dotyczy największej od 20 lat reformy Kodeksu spółek handlowych, jest pan poseł Krzysztof Bosak. Na tym właśnie polega praca nad prawem gospodarczym prywatnym, że odpowiadamy konkretnie na konkretne pytania. Pan wiceminister Jan Kanthak wskazał, że Platforma nie zgłosiła ani jednej poprawki, nawet najmniejszej, nawet przecinka.

Łatwo krytykować, ale warto zgłosić propozycje. To naprawdę nie była kwestia polityczna. Powiem tylko jedno.

Co do pana posła Dyducha, z wielką sympatią. Nie ukrywam, że będąc członkiem rady nadzorczej spółki KGHM, jednego z największych polskich koncernów, doszedłem do wniosku i wymyśliłem, że ta reforma jest potrzebna właśnie po to, żeby takie spółki jak Polska Miedź, KGHM, Grupa Orlen, Grupa Żywiec - jak wszystkie polskie firmy, które funkcjonują jako zgrupowania spółek, mogły prowadzić ekspansję gospodarczą, realizując własną wspólną strategię w ramach grupy spółek. Te przepisy prawa holdingowego są tak bardzo potrzebne, dlatego że - tak jak powiedziałem - 440 tys. firm na to czeka.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy wnioski o odrzucenie oraz poprawki, na podstawie art. 95 ust. 2 regulaminu Sejmu kieruję ten projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach celem przedstawienia sprawozdania. Komisja Kultury i Środków Przekazu przedłożyła sprawozdanie o poselskim projekcie uchwały w związku z setną rocznicą urodzin Tadeusza Gajcego, druk nr 1995. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Marszałek Sejmu proponuje, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk nr 1913) Uprzejmie proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Ryszarda Bartosika o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Bardzo proszę, panie ministrze.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Przedkładany projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawiera szereg zmian w obowiązujących przepisach, które z jednej strony mają na celu usprawnienie działania tej agencji, z drugiej - złagodzenie warunków udzielania pomocy w spłacie wierzytelności agencji. W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie możliwości umorzenia wierzytelności z tytułu Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa na wniosek osoby, która była stroną umowy o kredyt udzielony z tegoż funduszu, bądź jej następcy. Chodzi o osobę, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz nie posiada innej nieruchomości niż ta, w której zamieszkuje. W projekcie ustawy proponuje się także wprowadzenie możliwości umarzania wierzytelności, jeżeli wyłączną wierzytelnością jest wierzytelność z tytułu odsetek na wniosek osoby, która była stroną umowy o kredyt udzielony ze środków funduszu, bądź jej następcy prawnego. Dłużnikami z tytułu funduszu są przede wszystkim rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne na początku lat 90. Oznacza to, że obecnie dochodzenie tych roszczeń następuje od osób będących w wieku emerytalnym i oznacza windykację lub egzekucję roszczeń agencji z przysługujących im świadczeń emerytalno-rentowych, z rolniczego ubezpieczenia społecznego rolników. Należy również podkreślić, że zadłużenie z tytułu należności głównej wynosi ok. 1/4 całkowitego zadłużenia z tytułu funduszu. Pozostała część zadłużenia to zadłużenie z tytułu odsetek oraz zadłużenie z tytułu kosztów dochodzenia roszczeń przez agencję. Jednocześnie każdego roku narastające zadłużenie z tytułu odsetek jest wyższe niż odsetki spłacone. Poziom zadłużenia odsetkowego obsługiwanego przez spłatę nie osiąga nawet poziomu 50% narastającego zadłużenia z wyżej wymienionego tytułu. W przedkładanym projekcie proponuje się także uregulowanie umorzenia należności z programu przedakcesyjnego SAPARD. Obecnie należności w ramach programu SAPARD zarejestrowane są w księgach rachunkowych agencji i są należnościami obciążającymi wyłącznie budżet krajowy. W księgach rachunkowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozostają czynne 33 sprawy windykacyjne z otwartym saldem należności. W projekcie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przewiduje się również wprowadzenie przepisów umożliwiających wstrzymanie naliczania odsetek w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii od wierzytelności agencji, których spłata została odroczona lub rozłożona na raty, analogicznie do tego, jak to ma miejsce w przypadku środków ze wspólnej polityki rolnej. Mając na względzie, że nadzór nad instytucją zarządzającą PROW sprawuje minister rolnictwa i rozwoju wsi, zaproponowano, aby nadzór nad agencją na podstawie ustawy sprawował wyłącznie minister, natomiast minister finansów, podobnie jak w przypadku innych agencji, będzie sprawował nadzór nad agencją na podstawie przepisów o finansach publicznych czy na podstawie przepisów o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W przedkładanym projekcie przewiduje się również możliwość utworzenia przez agencję spółki z o.o., której celem będzie realizacja zadań polegających na zapewnieniu rozwoju systemów i rozwiązań teleinformatycznych służących do realizacji zadań agencji, w szczególności m.in. przez budowę, rozbudowę systemów lub rozwiązań teleinformatycznych. Jednocześnie w celu usprawnienia współpracy między instytucjami i organizacjami publicznymi oraz zapewnienia sprawnej obsługi rolników i innych podmiotów, na rzecz których realizowane są zadania publiczne w zakresie działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne lub rybołówstwo, spółka będzie mogła realizować również takie zadania (Dzwonek) na rzecz podmiotów innych niż agencja. Wnoszę o przyjęcie proponowanej przez rząd ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawi Wysokiej Izbie pan poseł Maciej Górski. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie!

I tutaj pan minister nie zdążył chyba tego wspomnieć, że to jest na wyraźną prośbę agencji, ponieważ doradca jest często wyznaczany, zatrudniany do konkretnego zadania, nie ma sensu z nim nawiązywać umowy o pracę, powołanie wydaje się znacznie szybszą i łatwiejszą formą i w przypadku zawarcia, i w przypadku rozwiązania.

Również ważną zmianą jest zmiana piąta, bo pozwala na zawieranie umów bez naboru stażystom, którzy odbyli staż w agencji restrukturyzacji, o ile są to umowy na zastępstwo lub nie krótsze niż 6 miesięcy, i to też wynika ze zmieniającego się rynku pracy. I tutaj mogę dodać, że jako były pracownik agencji spotkałem się z takimi sytuacjami, że przychodziły osoby z naborów i to utrudniało bieżące funkcjonowanie agencji, bo pozyskanie stażysty, który już zna specyfikę pracy, ma uprawnienia, ma zdane egzaminy, ma odpowiednie wdrożenie w dany proces to jest wartość dodana, to jest jakieś pół roku spokojnie.

I to też jest na prośbę ministra finansów. Zmiana siódma jest tutaj najbardziej wzbudzającą emocje, o czym wspomniał pan minister, umożliwi ona wzorem innych agencji wykonawczych powołanie przez agencję spółki do zadań IT. Spółka ta będzie w 100% podległa agencji, będzie pracować, jak czytamy w uzasadnieniu, na przekazanym, powierzonym w ramach umowy sprzęcie przez agencję, będzie też składać się z tych pracowników. Powołanie tej spółki zapewni zatrzymanie wysoko wykwalifikowanych pracowników do modernizacji tych systemów, do tworzenia i obsługi aplikacji niezbędnych do funkcjonowania nowoczesnego agencji. Co więcej, spółka ta będzie mogła wykonywać różne zadania powierzone przez właściwego ministra na podstawie umowy i będzie też miała zapewnione wtedy finansowanie tego ministerstwa. A więc myślę, że tutaj takie instytucje jak KRUS, KOWR czy ośrodki doradztwa rolniczego z czasem zaczną korzystać z usług tej spółki. Skończył się czas, a nie skończyłem. Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie popierał tę ustawę i zagłosuje za jej przyjęciem. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pani poseł.

Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej przedstawić projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej ustawą o agencji. Sam projekt tej ustawy jest bardzo duży.

Samo wyjaśnienie zajmuje 42 strony tego projektu ustawy. Są też propozycje np. oddłużania agencji, jeżeli chodzi o wierzytelności, jakieś takie historyczne, z bardzo dawnych lat, gdzie są problemy ze znalezieniem dłużników, część z nich jest już w wieku emerytalnym i spłata tych długów rzeczywiście przekracza ich możliwości. Część artykułów dotyczy rozszerzenia katalogu przesłanek, w oparciu o które mogą być umarzane wierzytelności agencji. Niektóre są.

Niektóre proponują, żeby pomoc udzielana podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie podstawowej produkcji rolnej została uznana za pomoc de minimis w rolnictwie. Część jest taka, że. Proponowana jest zmiana mająca na celu wykreślenie przepisów, zgodnie z którymi umorzenie wierzytelności agencji, której kwota przekracza 40 tys. zł, nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Jest również przepis, który proponuje wprowadzenie wyłączenia obowiązku przeprowadzenia naboru na zasadach określonych w tej ustawie. W przypadku zatrudnienia pracowników na czas określony chodzi o zastępstwo pracownika, który ma usprawiedliwione nieobecności.

Docelowe zatrudnienie w tej spółce jest planowane dla ok. 300 osób. 100-procentową własnością tej spółki byłaby agencja.

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi udzieli agencji dotacji celowej na pokrycie wkładu pieniężnego wnoszonego do spółki. Nadwyżka środków finansowych ustalona na koniec roku będzie odprowadzana do budżetu państwa. Model finansowania spółki w początkowych latach działalności w większości ma być w formie dotacji z budżetu państwa. Przewiduje się również, że minister właściwy do spraw rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych lub rybołówstwa może powierzyć spółce realizację zadań spółki na rzecz jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych. Oczywiście zamówienia w trybie z wolnej ręki z pominięciem Prawa zamówień publicznych, a więc praca (Dzwonek) podana.

Spółka będzie mogła nieodpłatnie uzyskiwać dane ze zbiorów danych, w tym zbioru danych osobowych, prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne.

Dziękuję. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Pan minister pokaże, czym chce się zajmować.

Pan minister nie zajmuje się tym, żeby pomagać rolnikom, walczyć z klęskami, wspierać polską wieś, tylko tak naprawdę tworzy kolejną spółeczkę dla swoich kolesi, przyjaciół Prawa i Sprawiedliwości. Jak się wczytać w to uzasadnienie, o którym tak szeroko mówiła pani poseł, to tam tak naprawdę widać takie modelowe, metodyczne podejście do tego, jak uwłaszczyć się na majątku państwa, w tym przypadku - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. A nie działa system informatyczny. Ten system informatyczny faktycznie w tej agencji nie najlepiej działa, ludzie za mało zarabiają, są kłótnie między tymi ludźmi itd. W normalnej firmie szef by to zdiagnozował, zobaczył, co się dzieje, próbował coś wdrożyć, monitorował i naprawiał. Otóż w państwie Prawa i Sprawiedliwości robi się coś zupełnie innego: tworzy się spółkę, która wyciągnie, wyssie z tej agencji 109 osób. One jak za dotknięciem magicznej, czarodziejskiej różdżki wszystko naprawią i wszystko będzie normalnie funkcjonowało, nie będzie więcej problemów z obsługą rolników, jeśli chodzi o cały ten system IT. Spółka to rady nadzorcze, spółka to szefostwo, a jak szefostwo to przecież gadżety, biuro, samochody, dodatkowe uposażenie.

Po cóż to jest, drodzy państwo?

Jeden aspekt, który przychodzi mi do głowy, to jest to, że państwo bardzo często posługujecie się czymś takim jak tajemnica spółki, tajemnica handlowa. Przecież wielokrotnie to powtarzaliście. Kończąc, pani marszałek, chciałem tylko powiedzieć, że klub Lewicy ocenia ten projekt negatywnie. Przynajmniej nie ma wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu. Pan poseł Stefan Krajewski w imieniu klubu Koalicja Polska. Bardzo proszę o zabranie głosu. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - PSL, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, druk nr 1913. Wysoka Izbo! W 2016 r., kiedy prezes Daniel Obajtek opowiadał o wielu nieprawidłowościach w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kiedy mówił, co trzeba naprawić, co trzeba zmienić, rozpoczęła się wielka naprawa. Przecież pamiętamy, jak prezes Obajtek z ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem otwierali Departament Informatyki w Lublinie, który miał być rozwiązaniem tych wszystkich bolączek, naprawieniem tego, co nie działa. Po prostu trzeba powoływać spółkę, bo ten departament nie spełnił swojej roli. Jak się weźmie pod uwagę siatkę płac.

To nie jest dobre z punktu widzenia tej zmiany, bo dzisiaj rolników interesuje to, żeby programy były realizowane sprawnie, żeby były wydatkowane pieniądze. Jeśli nie wprowadzi się dobrych zmian, takich, które naprawdę zreformują tę instytucję, to niestety będzie problem z wydatkowaniem pieniędzy, z rozliczeniem, z pracą. Drugi problem: pracownicy. Dzisiaj okazuje się, że nie ma ich kim zastąpić. Dobrze, że stażysta może przyjść do instytucji, pouczyć się, zobaczyć, jak to wszystko wygląda.

To trzeba zmienić.

Trzeba spłaszczyć siatkę płac, wynagrodzeń, bo główny specjalista może zarabiać od 3900 zł do 8900 zł, co jest niesprawiedliwe, bo na tych samych stanowiskach pracują ludzie, którzy zarabiają dwukrotnie więcej. To trzeba oczywiście naprawić i zmienić.

Będziemy się przyglądać i oczywiście proponować swoje poprawki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. I pan poseł Mirosław Suchoń w imieniu koła Polska 2050. Bardzo proszę, panie pośle. Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050 wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szanowni Państwo!

To nic innego jak przejęcie nadzoru nad bardzo lukratywnym tortem. Wychodzi na to, że ostatnie, powiedziałbym, spory w rządzie pomiędzy ministrem rolnictwa a ministrem finansów zakończyły się w tym zakresie zwycięstwem ministra rolnictwa.

Oceniamy, że to są zmiany idące w dobrym kierunku, chociaż pewnie wiążą się one po części z możliwością zatrudnienia politycznych nominatów, niemniej jednak dzisiaj widać wyraźnie, że rąk do pracy w agencji brakuje i ułatwienia w tym zakresie są potrzebne.

Natomiast art. 1 pkt 7 dotyczy możliwości powołania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez agencję i tutaj jak w soczewce widać wszystkie problemy i patologie władzy, które dzisiaj tę władzę obecnie rządzących cechują. Po pierwsze, agencja to kolejna spółka, która ma przejąć zadania, których nie potrafi zrealizować, jak wynika z uzasadnienia. Po drugie, kwestia wynagrodzeń.

To wypływa wprost z tego projektu. Będziemy się przyglądać, jak ten projekt się zmieni.

Przykro mi. Demokracja. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Jakie mamy gwarancje, że spółka zależna będzie spełniać zadania dotyczące ciągłości dostawy usług np. dla rolników, którzy będą korzystać z systemów informatycznych ARiMR-u? Jak będzie wyglądać serwis, obsługa reklamacji i jak to wpłynie na jakość obsługi właśnie rolników? I czy to będzie po stronie spółki, czy to będzie po stronie bezpośrednio ARiMR-u? Jak będą wyglądać kryteria zatrudnienia w porównaniu z tym, co jest dzisiaj? Ci nowi programiści, analitycy, kierownicy projektów, dyrektorzy, członkowie zarządu - przecież to są już nowe stanowiska. Chociaż rozumiem i akceptuję w pełni fakt, że powinni być traktowani właśnie rynkowo, skoro są specjalistami.

Czy to nie będzie też dokapitalizowanie właśnie tej spółki poprzez np. zawyżanie wycen analitycznych i wykonawczych? Bo to się będzie wiązać z niegospodarnością. To są ryzyka, z którymi będą państwo się musieli zmierzyć i wezmą państwo za to odpowiedzialność. I przy okazji też pozwolę sobie zwrócić uwagę na to, że dzisiaj zajmujemy się nową spółką córką, a są inne i ważniejsze jeszcze problemy w rolnictwie, jak właśnie ASF, jak to, że ci, którzy dzisiaj hodują trzodę, są w strefach i mają problem ze sprzedażą do skupów, jak to, że dzisiaj nasi hodowcy drobiu są atakowani chociażby na polu medialnym.

Dokument był pełen manipulacji, niedomówień czy materiałów właśnie nie z Polski. Na to nie ma naszej zgody.

Przechodzimy do pytań. Zamykam listę osób chcących zadać pytanie. Panie Ministrze! Sugerując się tymi wypowiedziami, szczególnie pana posła z Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak również pana posła Suchonia, chciałbym zapytać pana ministra o skalę wypłat płatności bezpośrednich. Ile zostało wypłaconych zaliczek? Ile zaliczek było wypłaconych za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego?

Chodzi o to, że gdy Prawo i Sprawiedliwość wzięło odpowiedzialność za Polskę, to na biurku pana ministra rolnictwa leżało pismo pana prezesa ARiMR-u, nie będę wymieniał nazwiska, że system w ogóle nie działa (Dzwonek) i nie ma przygotowanego systemu. Czy to jest prawda, że wtedy Agencja w ogóle nie była przygotowana do wypłaty dopłat? Pani poseł Iwona Maria Kozłowska, Koalicja Obywatelska. Uprzejmie proszę o zadanie pytania. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Art. 1 pkt 7 projektu ustawy przewiduje możliwość utworzenia przez agencję spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu świadczenia na rzecz ARiMR usług informatycznych. W uzasadnieniu możemy przeczytać, że państwo PiS nie jest w stanie zapewnić pracownikom odpowiednich płac, że szybko rosnące płace powodują, że ARiMR przestaje być atrakcyjnym pracodawcą. Tak, uzasadnienie w tej części jasno wskazuje, w jakim znaleźliśmy się w tej chwili miejscu. Doprowadziliście państwo do tego, że tworzycie spółkę, aby lepiej płacić pracownikom. Ten projekt, to nie tylko obraz dyskryminowania pracowników poprzez różnicowanie wynagrodzeń, ale przede wszystkim jest to obraz klęski szczytnie zapowiadanych wizji państwa dobrobytu pod kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości jako kraju dbającego w równym stopniu o wszystkich obywateli. Przez ostatnie 7 lat miało być lepiej, bogato, a Polacy mieli masowo wracać do Polski. Panie Ministrze! Pan poseł Rafał Adamczyk, klub Lewicy. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązań ułatwiających zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, skrócenia procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Interesuje mnie rok 2022, a szczególnie to, czy planują państwo jakieś zmiany na stanowiskach kierowniczych. Jeśli tak, to jakie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Ministrze! Szanowni Państwo!

Niestety, szanowni państwo, w ubiegłym roku w województwie zachodniopomorskim susza wystąpiła, natomiast aplikacja uniemożliwiła generowanie protokołów. Zresztą nawet pracownicy IUNG-u wysłani, żeby zobaczyć, czy faktycznie ta susza była, stwierdzili ją. Natomiast ta wspaniała aplikacja, którą przygotowali wspaniali informatycy, stwierdziła, że suszy w Polsce, w tym w województwie zachodniopomorskim, nie było. Ja w imieniu tych zachodniopomorskich rolników proszę pana ministra o to, żeby jednak pochylił się pan nad ich problemem, bo 4 lata - 3 lata susza, rok nawalne deszcze (Dzwonek) - to jest naprawdę ogromny problem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Czas - 1 minuta. Uprzejmie dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Trzy pytania. Po pierwsze, ten projekt i uzasadnienie dowodzą, że pracowników IT w agencji systemowo wynagradza się poniżej kwalifikacji. W mojej ocenie nosi to znamiona dyskryminacji. Czy ministerstwo w tej sprawie podjęło jakiekolwiek działania, żeby zmienić tę chorą sytuację, kiedy ludzi wynagradza się poniżej ich kwalifikacji? Po drugie, kiedyś, w dwa tysiące... już nie pamiętam którym, ale ok. 10 lat temu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego zamieniły system przygotowany przez ITS na system przygotowany przez PWPW, czyli wytwórnię państwową. To wiązało się z dziesięciokrotną podwyżką. 10 razy tyle dzisiaj WORD-y płacą za system teleinformatyczny. Czy daje pan gwarancję, że nie będzie dokładnie tak samo w tym przypadku? Dlaczego nie wykorzystano spółki Aplikacje Krytyczne, która została założona przez Ministerstwo Finansów (Dzwonek) i dysponuje odpowiednim zapleczem? Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Wrzuca się tam punkt, w którym mówi się o osobach starszych, które rzeczywiście mają problem z zapłaceniem swojego zadłużenia sprzed wielu, wielu lat. Dlaczego dopiero teraz się za to wzięto? Powstanie rada nadzorcza, zarząd, znowu będą osoby wynagrodzone. Niepokoi też dostęp spółki do zbiorów danych osobowych prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne. Istnieje w chwili obecnej centralna agencja rządowa z prężnym ośrodkiem informatycznym, który realizuje duże projekty, prowadzi rejestry (Dzwonek) i posiada już kadry. Ilu doradców prezesa jest zatrudnionych na dzień dzisiejszy w agencji?

Bardzo proszę. Znaczna część projektu poświęcona jest możliwościom i zasadom tworzenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spółek teleinformatycznych finansowanych ze środków agencji. Rząd wprost przyznaje, że powoływanie spółek IT przez agencję ma na celu obejście przepisów regulujących wysokość płacy w tejże agencji. Panie premierze, ja wiem, że dzięki Polskiemu Ładowi mają obowiązywać w naszym kraju dwa, a nawet trzy systemy podatkowe i każdy będzie mógł pewnie sobie wybierać, jak je mieszać pomiędzy sobą. Natomiast czy właściwym jest, aby ten sam rząd ustalał jakieś przepisy jedną ustawą, jak w tej ustawie, a w drugiej wskazywał, co należy zrobić, aby te przepisy obejść? Może w spółkach IT zasiądą całe kadry kierownicze agencji i w ten sposób będą mogły sobie ustalać wynagrodzenie na zupełnie innym poziomie niż dzisiaj. Do dyspozycji pozostają też rady nadzorcze w tych spółkach IT, które już wiemy, jak będą obsadzone.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Miesiąc temu zadawałem panu pytanie odnośnie do ASF-u, wypłaty wyrównań, pożyczek. Udzielił mi pan odpowiedzi, że pożyczki są udzielane płynnie, 2559 rolników otrzyma 130 mln zł w trybie bardzo pilnym. A dzisiaj ci rolnicy przychodzą do mnie do biura i pytają: Panie pośle, jak to się ma do tego? Chciałbym panu ministrowi powiedzieć jedną rzecz, że we Francji rolnicy mają takie same problemy finansowe jak polscy rolnicy.

Chciałbym, żeby państwo polskie też tak działało i żeby ta agencja, o której mówimy, wypłaciła rolnikom z Nowego Miasta (Dzwonek), Iławy, Działdowa, Żuromina odszkodowania z tytułu ASF.

Wysoka Izbo! Co zrobić, gdy dla swoich brakuje miejsca w agencjach i spółkach? Zlikwidować konkursy na stanowiska i zastąpić je dumnie brzmiącym powołaniem - właśnie do tego zmierza ta ustawa. W projekcie ustawy proponujecie zmiany w zakresie zasad zatrudniania w agencji. Proponujecie rezygnację z otwartych i przejrzystych naborów i jeszcze w szerszym zakresie aniżeli przewidują to ustawy o służbie cywilnej i ustawa o pracownikach samorządowych. Stwarza to oczywiście niebezpieczny precedens. Czytając projekt, mam wrażenie, że niektórym marzą się masowe czystki i wyrzucenie z dnia na dzień na bruk wieloletnich i zasłużonych pracowników i zastępowanie ich partyjnymi działaczami. Czy wam nie jest już dosyć? A może na skrzynce mailowej pana Dworczyka już jest prowadzony nabór na te stanowiska? Po co chcecie powoływać kolejną spółkę IT? Przecież wcześniej utworzyliście tzw. Departament Informatyki. A może jakiś znajomy znajomego chce otworzyć firmę informatyczną (Dzwonek) i chce współpracować z nowo powołaną spółką? Bardzo proszę o zadanie pytania. Wysoki Sejmie! Budzi nasze obawy nie sam fakt wydzielenia działalności IT w agencji, ale to, że to potwierdza, iż płace w agencji są na bardzo niskim poziomie. Pracownicy podstawowi w biurach powiatowych agencji, znaczna część z nich, ma wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej. Pytanie: Kiedy to się zmieni i jakie w tym roku przewiduje się podwyżki płac dla pracowników? Po drugie, chciałbym zapytać, korzystając z obecności pana ministra, o to, na jakim etapie jest w Komisji Europejskiej wniosek polskiego rządu dotyczący możliwości udzielenia dopłaty do nawozów. Jutro w całej Polsce wyjadą rolnicy swoimi ciągnikami i będą protestować przeciwko drożyźnie i kosztom funkcjonowania, m.in. w naszym województwie w Skalmierzycach (Dzwonek), również na drodze krajowej nr 25. Wobec powyższego to jest bardzo istotne. Dziękuję bardzo. Pan poseł Konrad Frysztak, Koalicja Obywatelska. Nie ma. Pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Uprzejmie proszę, pani poseł. Wysoka Izbo! Procedowana ustawa zakładająca m.in. poszerzenie katalogu stanowisk o doradcę prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to nic innego jak kolejny skok na stanowiska. Czyżby ktoś z otoczenia władzy pilnie potrzebował pracy? Zamiast tworzyć posady pod kogoś, może ministerstwo przyjrzy się temu, jaka panuje nierówność wynagradzania pracowników w agencji. Pracownicy mówią wprost, że nie liczą się wiedza i umiejętności, lecz jest tak, że kto ma układy polityczne, ten awansuje i dobrze zarabia.

Niestety. Pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Na pytania postawione przez panie i panów posłów odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Ryszard Bartosik. Zapraszam, panie ministrze.

Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Pytań padło wiele. W wielu pytaniach były zawarte treści, na które po prostu nie będę odpowiadał, bo państwo już wszystko wiedzą przed uchwaleniem ustawy, jak to będzie funkcjonowało. Bardzo długa lista zarzutów. Chcę powiedzieć, że padało tu sformułowanie: państwo PiS. Chciałbym powiedzieć, że nasze państwo to jest Rzeczpospolita Polska. Dobrze by było, abyście państwo posłowie znali nazwę i państwo, w którym funkcjonujecie, w którym zostaliście wybrani na reprezentanta narodu. Prosiłbym, aby się do tego w odpowiedni sposób odnosić, bo takie sformułowania po prostu nie powinny padać z tej mównicy. Szanowni Państwo! Ta ustawa przede wszystkim ma służyć rolnikom, poprawie obsługi rolników. Wiemy, że przed nami jest realizacja nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, wdrażanie planu strategicznego, dlatego też potrzebujemy wysoko specjalistycznych działań IT, wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Ta spółka będzie mogła obsługiwać również inne instytucje działające w rolnictwie, będzie mogła na wyższym poziomie świadczyć wysoko wyspecjalizowane usługi na rzecz przede wszystkim agencji w zakresie budowy, rozbudowy i unowocześniania istniejących systemów informatycznych. Szanowni Państwo!

Do tego dojdą te, o których mówiłem, czyli nowa perspektywa finansowa, plan strategiczny i inne działania. W związku z tym ta spółka jest nam niezbędna. Szanowni Państwo!

Właśnie tak, panie pośle. Ktoś tu pytał, czy zaliczki były wcześniej płacone. To za naszych rządów zaczęliśmy płacić zaliczki, a w takiej wysokości to w ostatnim czasie agencja to realizuje i te wypłaty są prowadzone bardzo sprawnie.

3/4 środków jest już w tej chwili wypłacone. Chcę powiedzieć, że wszystkie kwestie związane z wynagradzaniem są ściśle związane z budżetem państwa. W związku z tym wynagrodzenia i podwyżki będą realizowane.

Będziemy nadal pracować w komisji rolnictwa nad tą ustawą. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, poprawki czy propozycje Wysokiej Izby, państwa posłów. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Zamykam dyskusję. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy w bloku głosowań. W związku z tym, że legislatorzy pracują jeszcze nad poprawkami, a jest nam to potrzebne do przejścia do kolejnego punktu porządku dziennego, zarządzam 15 minut przerwy.

Wznawiam obrady. Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, druk nr 1997. W związku z tym, na podstawie art. 74 regulaminu Sejmu, marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Marszałek Sejmu proponuje, aby w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciw. Wobec? Zawsze mam tolerancję. W związku z tym uzgodniliśmy, że dla kół - 4 minuty. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (druki nr 1990 i 1997) Uprzejmie proszę pana posła Grzegorza Matusiaka o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, druk nr 1990. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 73 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierowała w dniu 7 lutego 2022 r. powyższy projekt ustawy do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych do pierwszego czytania. Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2022 r. wnosi: Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 4-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, druk nr 1990. Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych przeprowadziła w dniu dzisiejszym pierwsze czytanie projektu i rekomenduje jego przyjęcie.

Jednocześnie wydaje się, że bardzo pilna jest notyfikacja tzw. nowych wytycznych Komisji Europejskiej. Nowe zasady, znajdujące się w tych nowych wytycznych, wymagają ustawy. Stąd to pilne procedowanie nad dzisiejszą ustawą. Jeżeli wprowadzimy te zmiany i ich notyfikację, to tak naprawdę będzie to pomagało w uruchomieniu dodatkowych środków finansowych.

Może to też być produkcja energii odnawialnej oraz zmniejszenie zużycia energii.

Dlatego Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera przyjęcie tej ustawy. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Sławomir Neumann w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! To, że pani marszałek Witek i większość sejmowa traktują Sejm z dużą lekkością, nie oznacza, że wszyscy musimy się na to godzić. Bo proponujecie nam państwo na procedowanie nad tym projektem właściwie 24 godziny. Nad projektem, który wpłynął jako projekt pilny, rządowy, czyli do szybkiej ścieżki. Ale 24 godziny nad projektem, który ma 45 mld wagi, bo tyle pieniędzy przez kilka najbliższych lat ma być przeznaczonych na pomoc, to trochę mało. Tego nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak mało czasu. A jak wyglądał harmonogram prac?

W grudniu te wytyczne zostały ostatecznie opublikowane. Cały ubiegły rok rząd miał czas, żeby przygotować ten projekt.

To nie są, proszę państwa, dobre zasady legislacji i myślę, że powinniście wyciągnąć jakieś wnioski z tego bubla, który nazywacie Polskim Ładem, bo on pokazuje mnóstwo niedociągnięć.

Kiedy ustawę matkę, czyli tę ustawę podstawową, przyjęto w 2019 r., cena uprawnień wynosiła 24 euro za certyfikat. Dzisiaj to jest ponad 90 euro, prawie 100, i jeszcze pewnie może rosnąć. Tak wysokie ceny energii bardzo mocno odbijają się na branży energochłonnej.

Bo to nie dotyczy tylko huty, ale też zwykłej piekarni czy innej małej firmy. To są już efekty tych 6 lat zaniedbań i 6 lat błędnych decyzji, które państwo podejmowali. To są też skutki ponoszonych przez spółki energetyczne kosztów niezwiązanych z certyfikatami, a tak absurdalnych jak finansowanie różnego rodzaju fundacji, w tym Fundacji Narodowej.

To są też koszty, które spółki ponoszą, i one też wchodzą w cenę energii, np. na ostatnio zauważoną kłamliwą propagandę na bilbordach, która mówi o tym, że jakoby 60% kosztów energii to koszty związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, a wszyscy doskonale wiemy, że to jest absolutna nieprawda, bo opłaty związane z certyfikatami to jest ok. 23-24% kosztów tej energii. Reszta to koszty i różnego rodzaju obciążenia spółek, które generują m.in. taką głupią, kłamliwą, nieprawdziwą kampanią. Korzystając z tego, że dzisiaj mówimy o cenie energii, o kosztach, chcę z tej mównicy zapowiedzieć, że zwrócę się z pismem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z wprowadzeniem klientów w błąd przez spółki energetyczne, w związku z możliwym oszustwem związanym z ponoszeniem nieuzasadnionych kosztów i wpisywaniem tych kosztów z pozycji monopolistycznej, w jakiej są dzisiaj spółki w stosunku do klienta, w rachunki płacone przez klientów. My za te wszystkie rzeczy płacimy. Natomiast ta ustawa oczywiście jest potrzebna, bo pomoże chociaż części firm. 200 firm, które będą mogły korzystać z tej ustawy, przynajmniej ma szansę na to, że koszty energii będą dla nich niższe. Przypomnę, że w debacie w 2019 r. wiele osób wspominało na tej sali historię huty w Krakowie, która już wtedy ledwo dawała radę z tak wysokimi kosztami energii.

To jest pytanie otwarte. Ta ustawa, to wsparcie jest (Dzwonek) konieczne, potrzebne. Czy nie jest za małe? Mam olbrzymie wątpliwości, że jest za małe. Pan poseł Maciej Konieczny w imieniu klubu Lewica. Bardzo proszę. Przyznam, że ten tryb procedowania naprawdę jest wymagający, bo ta duża ustawa, o dużym poziomie skomplikowania pojawiła się wczoraj. Siłą rzeczy trudno było bardzo precyzyjnie rozmawiać o tym projekcie, a teraz już jesteśmy na sali plenarnej. Ale takie są warunki. W skrócie chodzi o przeznaczanie 25% wpływów pochodzących z handlu uprawnieniami do emisji w ramach systemu ETS na wsparcie tych sektorów przemysłu, które podwyżki cen energii dotykają najbardziej. Rekompensaty mają na celu utrzymanie konkurencyjności europejskiej produkcji przy jednoczesnym realizowaniu ambitnych celów klimatycznych. Chodzi o to, żeby ta produkcja nie uciekła poza granice Unii Europejskiej. Procedowana ustawa wdraża nowe wytyczne Komisji i radykalnie zwiększa skalę środków przeznaczonych na te rekompensaty. To wynika wprost z rosnących cen uprawnień. Mówimy o kwocie niebagatelnej, bo w ciągu 10 lat będzie to prawie 50 mld. Założenia są jak najbardziej słuszne, chociaż nie mam wątpliwości, że nie zabraknie podczas tej debaty głosów odsądzających od czci i wiary Unię Europejską, europejską biurokrację i obciążających Unię winą za wszystkie grzechy świata ze szczególnym uwzględnieniem rosnących cen i spadającego poparcia PiS. Ale może tym bardziej warto wykorzystać okazję, aby powiedzieć parę słów o tym, po co nam w ogóle te mechanizmy i te ambitne cele klimatyczne. Mamy kryzys klimatyczny, grozi nam globalna katastrofa. Przyczyną jest emisja gazów cieplarnianych. Jeżeli chcemy uniknąć najgorszego i przekazać kolejnym pokoleniom planetę zdatną do życia, to nasza gospodarka musi się radykalnie zmienić. Zdaję sobie sprawę z tego, że na tym etapie zgubiłem już część sali, która uparcie odmawia zaakceptowania wiedzy naukowej. Ale cóż, spróbujmy zgubić kogoś jeszcze, bo musimy być świadomi. To globalny kapitalizm, prymat zysku ponad wszystko doprowadziły nas na skraje katastrofy.

Nie podejmą takiej decyzji z oczywistych względów: bo natychmiast zostaliby zwolnieni. Taki mamy system. Zyski natychmiast lądują na kontach nielicznych, a przyszłe i obecne koszty cedowane są na nas wszystkich, a w największym stopniu, co wydaje się wyjątkowo niesprawiedliwe, na tych, którzy dopiero wkraczają w dorosłe życie albo dopiero wkroczą w nie w przyszłości. Dlatego potrzebujemy regulacji. Potrzebne są mechanizmy, które skłonią przedsiębiorstwa do zmiany i przekierują naszą cywilizację na zielone tory. Jako że nie są to rzeczy, które da się załatwić na poziomie jednego kraju, to w naszym wypadku mówimy głównie o regulacjach europejskich. Unia Europejska zdecydowała się na system handlu uprawnieniami do emisji, po to żeby opłacało się raczej mniej emitować dwutlenku węgla niż więcej. Sam nie jestem wielkim fanem tego rozwiązania. Rynkowy, a nawet spekulacyjny charakter ETS-u naraża przedsiębiorstwa nie tylko na dotkliwe, ale i nieprzewidywalne koszty. Zapewne można sobie wyobrazić bardziej funkcjonalny i bardziej przewidywalny system opodatkowania emisji. Z pewnością trzeba skończyć ze spekulacyjnym charakterem ETS-u, ale też nie można wylewać dziecka z kąpielą, nie można zapominać, że to wszystko jest po coś. Jedno jest pewne: ambitne cele klimatyczne wiążą się z kosztami i obawa o konkurencyjność europejskiej gospodarki jest w tym kontekście jak najbardziej uzasadniona. Dlatego ta ustawa jest potrzebna i dlatego te rekompensaty mają sens. Dlatego także inne mechanizmy, jak np. cło węglowe na wejściu do Unii Europejskiej, tak żeby wyrównać te szanse, są dobrym rozwiązaniem. Warto również zwrócić uwagę, że wśród wymogów stawianych przedsiębiorstwom ubiegającym się o rekompensaty są te dotyczące standardów energooszczędności. To jest kolejny impuls rozwojowy, który musi się zwrócić w przyszłości, bo kryzys klimatyczny jest faktem, a nowa zielona rewolucja przemysłowa jest koniecznością. Zresztą dzisiaj już płacimy cenę za to, że naszego systemu energetycznego nie zmienialiśmy przez ostatnie 10-20 lat. Jeżeli dzisiaj nie będziemy świadomie podejmować wysiłku na rzecz zmiany, to będziemy coraz bardziej w tyle, te koszty będą spadały na nas w coraz większym stopniu.

Ale też nie da się ukryć, że startowaliśmy z dużo niższego poziomu i że jako Polska jesteśmy w dużo trudniejszej sytuacji niż nasi zachodnioeuropejscy partnerzy. Ale nie da się uniknąć wrażenia, że dla obecnie rządzących Unia Europejska (Dzwonek) już nie jest przestrzenią walki o polskie interesy, a jedynie wymówką dla nierobienia niczego. Dziękuję bardzo. Pan poseł Władysław Teofil Bartoszewski w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - PSL, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Jest rzeczą zabawną, że dotyczy on dyrektywy nr 87 z 2003 r., przeciwko której cała prawa strona tego Sejmu protestuje, mimo że ostatnie zmiany do tej ustawy w 2018 r. podpisał nie kto inny, jak pan premier Mateusz Morawiecki.

I co myśmy zrobili przez ostatnie lata?

W 2016 r. większość parlamentarna, czyli Zjednoczona Prawica, zabiła ustawę o wiatrakach na lądzie, czyli 10H. 2 mln Polaków czeka na podłączenia do paneli słonecznych, a daliśmy przyzwolenie na 86 tys. Biomasa została wykreślona z programu zmiany energetycznej.

A ile będzie kosztowała z wiatraków na morzu? Dwa razy tyle.

Do tego, ponieważ nie inwestujemy w sieci niskiego napięcia.

Mimo wszystko jest to mały krok w dobrym kierunku i klub Koalicji Polskiej poprze ten projekt z nadzieją, że rząd się zreflektuje i zacznie zwracać uwagę również na odnawialne źródła energii. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Mirosław Suchoń w imieniu koła Polska 2050. Uprzejmie dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050 w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. To jest oczywiście ważny projekt i nie mamy co do tego żadnych wątpliwości, ale też niezrozumiała w związku z tym jest postawa rządu, który w zasadzie od września czekał, żeby przedstawić ten projekt ustawy Wysokiej Izbie. Dzisiaj mamy to przeprocedować w jeden dzień, ale tak naprawdę pokazuje to stosunek rządu generalnie do transformacji energetycznej, do zmian klimatycznych, do OZE i wszystkich tych aspektów, które są dzisiaj wyzwaniem dziejowym, wyzwaniem, któremu jeżeli podołamy, to przyszłe pokolenia będą miały szansę tutaj mieszkać, będą miały szansę normalnie żyć, a jeżeli nie podołamy, to zniszczymy planetę. I powiem tak: niestety te działania rządu nie sprzyjają ochronie tej planety na takim poziomie, jakiego dzisiaj wszyscy wymagamy. Oczywiście kwestia wsparcia firm energochłonnych, przemysłów energochłonnych jest poza jakąkolwiek dyskusją. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, co by było, gdyby dzisiaj te firmy narażone na wysokie koszty energii, na cały system finansowy, który istnieje, zostały pozbawione tej pomocy.

W związku z tym to wsparcie jest konieczne, ale też przez ostatnie lata nikt za bardzo tym się nie interesował. Trzeba przypomnieć, że firmy, zamiast być motywowane do tego, aby myślały o przyszłości, myślały o tej zmianie energetycznej, myślały o zmianie paradygmatów, były zachęcane raczej do tego, żeby tym się nie przejmować, nie brać tego pod uwagę w kosztorysach, nie brać tego pod uwagę w planach inwestycyjnych. I oczywiście z każdym krokiem, z każdym rokiem, kiedy odsuwa się takie zmiany, one stają się coraz bardziej kosztowne. Dzisiaj rosnące ceny energii powodują, że boli to każdego. Te rekompensaty, choć są potrzebne, oczywiście nie wyczerpują tego obszaru pomocy, który jest potrzebny. Dzisiaj powinniśmy jako państwo dać jasny sygnał, jasny impuls dla wszystkich tych przemysłów, że nadszedł czas na racjonalne, męskie decyzje, które spowodują, że do 2050 r. firmy te będą w stanie osiągnąć neutralność energetyczną, neutralność klimatyczną. Dzisiaj po stronie rządu nie widzimy tej determinacji, która skutkowałaby podejmowaniem przez gospodarkę odpowiednich działań, która skutkowałaby zapobieganiu tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, czyli niewprowadzane w odpowiednim momencie zmiany skutkują wyższymi cenami energii, skutkują wyższymi obciążeniami dla obywateli. Dzisiaj potrzebujemy tej zmiany paradygmatów. Potrzebujemy także takiego impulsu dla innowacyjności. Już o tym mówiłem podczas posiedzenia komisji.

To jest niezwykle ważne, żebyśmy dzisiaj nie tylko poprzestawali na wsparciu, ale także dali impuls do myślenia o przyszłości. I druga rzecz: podnosimy nakłady z 50% do 55%, uważając, że to jest ten docelowy kierunek. Bardzo proszę o przyjęcie tych poprawek. Dziękuję. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przemysł energochłonny w Polsce to 1,5 mln zatrudnionych osób wraz z kooperantami, to setki miliardów dochodu tworzonego w Polsce, to prawie 90 mld podatków, które w sumie kumuluje ten przemysł, które przynosi do polskiego budżetu. To jest olbrzymia, fundamentalna część polskiej gospodarki. Ta fundamentalna część polskiej gospodarki jest dzisiaj rozjeżdżana walcem przez unijną politykę klimatyczno-energetyczną i trzeba to sobie jasno powiedzieć.

Szanowni Państwo! To jest jeden z ostatnich dzwonków alarmowych, to jest jeden z ostatnich momentów, żeby zawrócić z tej błędnej drogi. Ten dyktat brukselski przychodzi i mamy to wykonywać, mamy niszczyć naszą gospodarkę i mamy na gwałt się dostosowywać. Koszty są nieporównywalnie wyższe niż zyski płynące ze wszystkich funduszy unijnych, ze wszystkich planów zadłużenia zwanych planami odbudowy. Zróbmy wreszcie rachunek zysków i strat. Chodzi o to, żeby Polska była i pozostawała jedynie podrzędną montownią w europejskim obiegu gospodarczym. Chodzi o to, żeby realizować utopię zielonych ładów, a raczej kolejnych nieładów w perspektywie najbliższych lat i dekad. Powiedzmy też sobie jasno, że rozwiązania, które forsuje dzisiaj Bruksela, będą prowadziły do tego, że europejskie gospodarki, w tym zwłaszcza gospodarka polska, nie będą konkurencyjne na świecie, będą traciły na konkurencyjności.

Nadajmy polskiej gospodarce nowy dynamizm.

Policzmy pieniądze, panie pośle. No to właśnie policzmy. Dziękuję bardzo, panie pośle. Przechodzimy do pytań. Wyznaczam czas na zadanie pytania - 1 minuta. Pytanie pierwsze zada.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Pani Minister!

Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Kolejne pytanie zada pan poseł Jan Szopiński, Lewica.

Wysoka Izbo! W dokumencie tym widać oczywiście fachową rękę twórców Polskiego Ładu. Tak jak i poprzednio pod ustawą podpisał się pan premier Mateusz Morawiecki, który pewnie tak jak w przypadku Polskiego Ładu powie za kilka dni, że chciał dobrze, ale dokładnie nie wiedział, co tam było napisane.

Tymczasem w treści ustawy w art. 33 widnieją nowe limity dopłat na lata 2022-2031. Kwota na rok 2021 pozostała bez zmian, na poziomie ustalonym w roku 2019, więc na długo przed skokową zmianą cen nośników energii. Należy w związku z tym spodziewać się, że projekt ten ma charakter w tej części chyba jednak propagandowy i za kilka miesięcy (Dzwonek), gdy przedsiębiorstwa otrzymają odmowy dopłat, do dymisji poda się minister odpowiedzialny za przygotowanie tego projektu. Pani poseł Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska. Nie ma pani poseł. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Bardzo bym prosił, żeby ministerstwo było uprzejme wyjaśnić, czy planuje jakieś zachęty bądź też inne działania, które by stanowiły impuls dla przemysłów energochłonnych do przygotowania zmiany technologicznej, zmiany w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej, i bardzo bym prosił o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo, panie pośle.

Zapraszam, panie pośle. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Kolejny raz mówimy o rekompensatach.

Wszystko to wynika z nieróbstwa rządu Prawa i Sprawiedliwości. źródeł energii, żeby przygotować grunt pod te firmy, które dzisiaj mają rzeczywiście problemy, żeby mogły sięgnąć po energetykę odnawialną. Panie ministrze, pytam pana w imieniu tych małych, średnich, mikro przedsiębiorców, jaką dla nich macie dzisiaj ofertę. Te zakłady pracy dziś się zamykają, podnoszą ceny. Co rząd chce dać tym firmom? Kolejne pytanie. Panie ministrze, czy rząd w jakiś sposób koordynuje i sprawdza, monitoruje (Dzwonek) podmioty, które otrzymują dofinasowanie, ceny tych towarów, które wypuszczają te firmy na rynek?

Bardzo proszę, panie pośle. Panie Ministrze! Przemysł energochłonny to w większości przemysł przeróbki rud metali, a więc rudy żelaza, dalej produkcja stali, ale też miedzi, aluminium i w mniejszych ilościach innych metali. Wszyscy wiemy, jak jest to ważne w gospodarce i budownictwie, w tym w energetyce. Przesył energii elektrycznej, ale także przesył paliw i gazu to są tory kolejowe, linie energetyczne.

Dlatego cieszy dzisiejsza ustawa. Ale jaka jest dalsza droga, aby zapobiec ucieczce tego przemysłu z Unii? Czy ministerstwo planuje poza rekompensatami wsparcie dla zmniejszenia zużycia energii, zmniejszenia emisji czy też stosowanie własnej energetyki odnawialnej? Czy są prowadzone w Polsce badania, jak zmniejszyć zużycie energii? To ważne, dlatego że zmniejszenie emisji (Dzwonek) miało miejsce już w przemyśle samochodowym i tutaj zmniejszenie emisji znacznie się udało. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, panie pośle. Jeżeli chcemy taniej energii elektrycznej i taniego ciepła, i konkurencyjnej polskiej gospodarki, to ten patologiczny unijny system handlu emisjami trzeba po prostu zlikwidować. Polska powinna wyjść z unijnej polityki klimatycznej, bo to jest jedna wielka drożyzna.

My naprawdę chcemy się od rosyjskiego gazu uwolnić. Unia Europejska dzisiaj jest przez Władimira Putina szantażowana. Naprawdę proszę nie brnąć w narrację Waldemara Pawlaka i bronić sprawy przegranej. Polska powinna wykorzystywać swoje własne zasoby, dlatego ja bronię polskiego węgla, a pan, jak widać, niestety broni rosyjskiego gazu. Przypominam, że jesteśmy w punkcie: pytania. Pan poseł Grzegorz Matusiak, Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł, ale ja pani nie pytałam. Proszę tak naprawdę wziąć głęboki oddech. Bardzo proszę. Szanowni państwo, słuchając tutaj wypowiedzi opozycji, można zadać pierwsze takie klasyczne pytanie... jestem za, a nawet przeciw.

To nie wypada, żebyście dzisiaj państwo krytykowali coś, czego jesteście winni, bo dzisiaj wina leży po stronie Tuska, pani Kopacz. To właśnie wy zrealizowaliście plany Unii Europejskiej w stosunku do naszych sektorów, a szczególnie energochłonnych. Panie ministrze, jest takie pytanie, czy były przeprowadzane konsultacje z przedsiębiorstwami na temat właśnie dzisiejszej ustawy i czy ta ustawa ze względu na tempo, które nadajemy, jest bardzo konieczna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Sławomir Neumann, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo!

A potem mówicie, że chronicie Polskę przed rosyjskim gazem, który też kupujecie, a za chwilę chcecie kupować go przez Baltic Pipe, bo tam będzie dostarczany rosyjski gaz. A więc trochę pokory. Natomiast sprawa jest poważna, bo cena energii tylko w 23% wynika z certyfikatów i ich cen. Pozostaje 75% i jest do was pytanie: Czy wy się zastanawiacie, jak przeprowadzić transformację, żeby wszystkim firmom żyło się lepiej i były tańsze rachunki za gaz, za prąd? Dziękuję bardzo, ale pytanie było na koniec. Oddaję hołd. Pani poseł Gabriela Lenartowicz, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie!

Pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska.

I tam nie ma nic o pomocy dla polskiego górnictwa.

W innych krajach podwyżki cen nośników energii i gazu to ok. 50% w tej sytuacji, jaką mamy, a u nas dla piekarza 1000%. On ma 1000% podwyżki, a inne kraje potrafiły dać wsparcie dla przedsiębiorców (Oklaski), dać taką samą taryfę jak dla ludności. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W ubiegłym roku Polska na sprzedaży praw do emisji dwutlenku węgla zarobiła ponad 25 mld zł. Ze wszystkich europejskich krajów to jest najwięcej. Co najmniej połowa tych pieniędzy powinna zostać przeznaczona na cele związane z poprawą klimatu, ale zamiast tego wpompowaliście te środki do budżetu, a od dawna przez was zapowiadany Fundusz Transformacji Energetyki wciąż nie istnieje. Panie Ministrze! Kiedy wreszcie weźmiecie się do pracy, kiedy wreszcie doczekamy się otworzenia tego funduszu? Czy potrafi pan podać konkretną datę?

Gdy zamiast tego po raz kolejny będziecie te pieniądze przejadać w spółkach, wyrzucać w błoto, na TVP, na CPK, na bezsensowny mur na granicy, pomyślcie o swoich dzieciach, wnukach i ich dzieciach. To ich przeszłość dzisiaj przejadacie. Ale czy warto? Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! Oto balonik propagandowy firm energetycznych. Żaróweczka, którą każdy otrzymuje - tu jest tylko 6% kosztów własnych, a 94%, łącznie z tym czerwonym, winne jest państwo, bo nakłada podatki. Winna jest Unia Europejska i polityka klimatyczna. My, dobrzy ludzie z Enei i innych, to tylko 6%. Obywatele, którzy mają taryfę G, właśnie dostają takie pozdrowienia.

Wysoki Sejmie!

Chciałbym się odnieść do bardziej ogólnych kwestii, ściśle związanych z tym projektem i nie tyle może zarzutów, co pewnych wątpliwości związanych przede wszystkim z tym, dlaczego m.in. on był w takim tempie procedowany.

Komisja Europejska rzeczywiście. Jeśli chodzi o same wytyczne, to one zostały przedstawione w 2020 r.

Bez tego, bez informacji, które tam zostały zawarte i upublicznione, czyli wskaźników, nie byliśmy w stanie w ogóle obliczyć poziomu rekompensat. Jeśli chodzi o sam poziom rekompensat, to chciałbym uspokoić tych, którzy wskazywali ewentualnie na głosy, które wskazywały na to, że on mógłby być niedostateczny.

Wszystkie wnioski powinny zostać rozpatrzone pozytywnie.

Limit wynosi 4 mld i prawie 200 mln, dokładnie 189 mln zł.

To jest bardzo duży zakres produkcji.

Chodzi o świadomość tego, że konkurencja wymaga nowych technologii. Było bardzo duże oczekiwanie ze strony branży właśnie na to, żeby tego typu pomocna dłoń ze strony państwa została wyciągnięta i żeby te rekompensaty wreszcie zafunkcjonowały. Oczywiście, to nie jest wszystko.

Pracujemy nad tarczą osłonową, jeśli chodzi o te kwestie, chociaż one oczywiście w większości nie będą się tutaj mieścić. Ministerstwo Rozwoju i Technologii w tej chwili takie prace prowadzi.

Dotychczas w Unii Europejskiej, z tego co się orientuję, jedynie Włochy wdrożyły ten środek. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Ogłaszam przerwę do godz. 17.45.

obrady.

W związku z tym, na podstawie art. 74 regulaminu Sejmu, marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Marszałek Sejmu proponuje, aby w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o pilnym rządowym projekcie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (druki nr 1989 i 1996) Proszę pana posła Radosława Fogla o przedstawienie sprawozdania komisji. Dziękuję uprzejmie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W związku ze skierowaniem pilnego rządowego projektu ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii komisja rozpatrzyła ten projekt ustawy. Zaproponowano poprawki, z których część komisja zaopiniowała pozytywnie. Po posiedzeniu w dniu 8 lutego komisja wnosi, by Wysoki Sejm raczył uchwalić załączony projekt ustawy. Bardzo dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Jako pierwszy pan poseł Radosław Fogiel w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję serdecznie raz jeszcze, panie marszałku. W pełni podtrzymuję wszystko to, co mówiłem w moim porannym wystąpieniu, podczas pierwszego czytania.

Rozwiązanie jest zgodne z wymogami i potrzebami sytuacji.

Brzmienie jest w treści poprawki.

Ponieważ w ustawie - Prawo telekomunikacyjne nie było definicji dekodera telewizyjnego, było potrzebne właściwe odwołanie do takiej definicji, która jest w niniejszej ustawie.

Dziękuję serdecznie. Proszę o zabranie głosu pana posła Grzegorza Napieralskiego, Koalicja Obywatelska.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Podobnie jak pan poseł przede mną powiem, że podtrzymuję to wszystko, co mówiłem dzisiaj rano, jeżeli chodzi o nasze stanowisko w tej sprawie. Ale dlaczego tak późno i dlaczego tak na szybko i tak pilnie, panie pośle, panie ministrze?

Druga kwestia to oczywiście przygotowanie tej ustawy. Mamy co do niej dużo zastrzeżeń ze względu na taką.

To pokazuje, że ktoś naprawdę pisał to bardzo szybko i nie zdążył tego dokładnie przemyśleć. Bardzo, bardzo mi przykro, że to tak niestety wygląda. A sprawa jest poważna, bo jeżeli nie przyjmiemy tych rozwiązań i ludzie nie wymienią dekoderów, to od czerwca czy lipca blisko 2 mln albo ponad 2 mln, bo tego dokładnie nie wiemy, gospodarstw domowych nie będzie mogło oglądać telewizji, nie będzie mogło oglądać swoich ulubionych programów edukacyjnych, informacyjnych czy też programów, które przynoszą im rozrywkę i radość.

To też padało dzisiaj na posiedzeniu komisji i w dyskusji, że jednak te osoby, które są niepełnosprawne, a potrzebują dodatkowej pomocy, nie zostały w tym projekcie uwzględnione, one nie zostały w ogóle potraktowane priorytetowo. One naprawdę mają już trudne życie, a jednak ta ustawa również dotyczy ich. A wiemy, że ta nowa technologia może być im również pomocna i może być dla nich bardzo dobra. Cały czas mówicie, że to osoby, które się zgłoszą i zadeklarują.

Będziemy o to prosić tak naprawdę. Chcielibyśmy tę umowę, która zostanie zawarta z operatorem, najpierw omówić na posiedzeniu komisji, zobaczyć, jak ona wygląda. Nie łamiemy tajemnicy państwowej, to są przecież publiczne pieniądze, więc taką propozycję też będziemy wnosić, panie ministrze, szanowni państwo, po to, aby to działało.

My składamy sześć poprawek. Te poprawki, panie ministrze, panie pośle, składamy. Te poprawki są tutaj. Pani poseł Małgorzata Prokop-Paczkowska, klub Lewicy. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ustawa jest procedowana w trybie pilnym, a więc rano - pierwsze czytanie, wyraziliśmy jako kluby opozycyjne swoje wątpliwości i pytania. Podczas posiedzenia komisji pan minister starał się na te pytania odpowiedzieć, starał się zniwelować nasze wątpliwości. Z pewnością nie wszystkie wątpliwości udało mu się odeprzeć. Krzysztof Gawkowski pytał np. o osoby niepełnosprawne, osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie te niewidome, niedowidzące, jak im pomóc w dostępie do telewizji cyfrowej.

Pan minister odpowiedział mi, że promocją zajmuje się Instytut Łączności i że będziemy mieli pełny wgląd w wydatki, w to, na co te pieniądze zostaną przeznaczone, w jaki sposób ta kampania informacyjna będzie przebiegała. Bo oczywiście bałam się i dalej się boję, że jakaś część z tych pieniędzy przeznaczonych na kampanię informacyjną trafi np. do TVP. Tak że, panie ministrze, nie wszystko nam pan wyjaśnił i rozjaśnił. Lewica poprze tę ustawę, aby pomóc tym rzeczywiście najbiedniejszym, którzy nie mają możliwości wydatkowania z własnych środków 100 zł na dekoder. Mamy nadzieję, że osoby dobrze sytuowane nie wystąpią o tę pomoc, która nie jest im potrzebna. Dziękuję. Pani poseł Urszula Nowogórska, Koalicja Polska, zdalnie. Dzień dobry, panie marszałku. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ponownie mam zaszczyt przedstawić stanowisko mojego klubu, klubu Koalicji Polskiej - PSL, Unii Europejskich Demokratów, Konserwatystów, Marka Biernackiego, w sprawie rządowego projektu ustawy zawartego w druku nr 1989 o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. W poprzednim wystąpieniu, panie marszałku, zadawałam wiele pytań dotyczących zabezpieczenia danych osobowych osób, które będą ubiegać się o dofinansowanie na zakup dekodera. Te pytania wynikały z głębokiej troski o konieczność zabezpieczenia danych wrażliwych Polaków, by uchronić ich przed oszustami, handlem bądź wyciekiem danych osobowych. Powiem szczerze, że dalej nurtują mnie te pytania w zakresie bezpieczeństwa. Te pytania pogłębiły się w zasadzie po posiedzeniu komisji cyfryzacji, ponieważ na tym posiedzeniu usłyszałam, iż dane osób będą zbierane nie w formularzach ministerstwa, tylko w formularzach, które zostaną stworzone przez operatorów dopuszczonych do programu. Dlatego zastanawiam się, w jakiej bazie danych będą gromadzone dane wrażliwe Polaków i jak one będą zabezpieczone. Szybkie procedowanie nad ustawą, mimo iż już od długiego czasu wiadomo o konieczności wprowadzenia zmian w standardach nadawania, może spowodować braki w dostępności do dekoderów lub gwałtowny skok cen tych urządzeń, co może utrudnić realizację założeń programu.

Z tą niepewnością będą borykały się osoby, które przystępują do programu i będą chciały skorzystać z dofinansowania. Panie Marszałku! Mam nadzieję, że wszystkie niejasności lub wątpliwości zostaną uszczegółowione w przepisach wykonawczych do projektu ustawy. Mam również nadzieję, że umowy zawierane między operatorami a ministerstwem będą jasne i rzetelne, szczególnie w zakresie przekazywania środków finansowych. Oczywiście jako klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej jesteśmy też w niezręcznej sytuacji, bo projekt procedowany jest szybko. Ale mimo to, panie marszałku, poprzemy ten projekt, dlatego że uważamy, że każde rozwiązanie systemowe, które wspiera Polaków, szczególnie seniorów np. w trudnej sytuacji materialnej, jest warte poparcia. Bardzo dziękuję. Teraz pan poseł Artur Dziambor, Konfederacja.

Szanowni Państwo! Ta ustawa - dość szybko napisana, o czym już było wspomniane, bo troszkę poprawek redakcyjnych trzeba było tam zrobić i możliwe, że jeszcze do tego jakoś będzie trzeba zajrzeć - jest o tyle ciekawa, że chociaż cały czas mamy hulającą inflację, to wy znowu chcecie rozdawać pieniądze. To po pierwsze. Po drugie, usłyszałem tutaj z sali, że jest to bardzo ważna sprawa, ponieważ jeżeli czegoś z tym nie zrobimy, to już za pół roku niektórzy nie będą mogli oglądać swoich ulubionych programów. Wiadomo, ten sprzęt się starzeje. Rząd powinien jakoś zadziałać, dać tym ludziom możliwość dostępu do wszystkich aplikacji, które mają ci, których z jakiegoś powodu stać było na zakupienie nowego sprzętu. Jest to oczywiście coś odlotowego, ale też przyzwyczailiście nas państwo do tego, że takie decyzje podejmujecie. Mamy sytuację, w której oczywiście tworzycie rynek dla tych dekoderów.

On nie ma w tym momencie żadnego zastosowania, szczególnie że dofinansowaliście Telewizję Polską 2 mld zł, po to żeby mogła rozkręcać tę propagandę wedle waszego, partyjnego uznania, bo przypomnę, że jeden z waszych partyjnych funkcjonariuszy z działu propagandy jest prezesem Telewizji Polskiej i ta telewizja w odpowiedni sposób się ustawia wobec władzy. Szanowni Państwo! Nie do końca rozumiem, dlaczego nagle ta ustawa się pojawiła i dlaczego chcecie to wprowadzić. Nie wiem, kogo chcecie tym zadowolić, chociaż jestem w stanie sobie wyobrazić, że może wam zależeć na tym, żeby znowu elektoratowi powiedzieć: proszę bardzo, my, Prawo i Sprawiedliwość, rozdajemy pieniądze.

Nie wiecie, gdzie jesteście. Pisząc tę ustawę. To jest jedna z najbardziej fascynujących rzeczy, ponieważ tu, w Sejmie, gdy pisze się ustawy, to trzeba podać koszty tych ustaw, a wy strzelacie. No już, trzeba to odrzucić.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W zasadzie posiedzenie komisji i prace, które prowadziliśmy w ciągu dzisiejszego dnia, nie wyjaśniły większości moich wątpliwości związanych z tym projektem. Oczywiście jestem przekonany, że to dofinansowanie jest potrzebne i prawdopodobnie, nawet na pewno będę zachęcał moje koleżanki i kolegów do tego, żeby poprzeć to rozwiązanie. Natomiast w dalszym ciągu jest tutaj wiele niewiadomych. Obawiam się, że tych niewiadomych nie rozwiążemy. Główna niewiadoma to kwestia notyfikacji europejskiej tego prawa, które przecież stanowi pomoc publiczną.

Nie będzie można kupić np. nowego telewizora, korzystając z rządowego dofinansowania. W tym kontekście po raz kolejny złożę poprawkę Koła Parlamentarnego Polska 2050, która rozszerza zakres urządzeń, które można współfinansować w oparciu o rządowe świadczenie, również o odbiorniki naziemnej telewizji cyfrowej. Pojawia się wiele kontrowersji, np. w jaki sposób chcą państwo sprawdzać prawdziwość oświadczeń dotyczących sytuacji materialnej, dlatego że jednym z elementów, które będą upoważniały osobę do otrzymania takiego świadczenia, będzie złożenie przez nią oświadczenia o tym, że ma trudną sytuację materialną, która nie pozwala jej zakupić takiego dekodera czy odbiornika we własnym zakresie. To oświadczenie oczywiście będzie składane pod groźbą postępowania karnego, tylko nie za bardzo wiadomo, co dalej, tzn. nie za bardzo wiadomo, co będzie w przypadku, gdy ktoś takie oświadczenie złoży, a ono nie będzie zgodne z prawdą. Reasumując, psują państwo rynek.

Koło Parlamentarne Polska 2050 składa poprawkę, która chociaż w jednym aspekcie odpowie na nadzieje ekspertów formułowane w korespondencji związanej z tą ustawą. Dziękuję bardzo. Jako pierwszy pan poseł Rafał Adamczyk z Lewicy. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Bardzo bym prosił o informację, na podstawie jakich danych i jakich źródeł pan ocenił, że 2 mln gospodarstw w Polsce będzie wymagało zakupu dekodera do odbioru co najmniej telewizji naziemnej. Dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ale jeżeli już mamy pomóc Polakom, to rzeczywiście tam, gdzie trzeba, pomagajmy. I taki powinien być finał tej wypowiedzi. Niestety trzeba Polakom też jasno powiedzieć, że skala informacji, którą przekażą tym, którzy mają im wypłacić te 100 zł, za chwilę może spowodować to, że ci wszyscy, którzy nie płacą abonamentu, zapłacą go, bo rząd nic nie daje za darmo.

W związku z tym mówimy A, ale może powiedzmy, panie ministrze, B.

Poproszę o odpowiedź na piśmie. Panie Człowieku Wolności Kaczyński! Wysoka Izbo! Poprę dofinansowanie w wysokości 100 zł na dekodery pod warunkiem, że oprócz dostosowania do odbioru telewizji naziemnej będą miały także funkcję odkłamywania telewizji rządowej. Jeśli zdekodują te steki kłamstw, manipulacji, nienawiści, które każdego dnia sączy w uszy Polek i Polaków TVPiS. Jak najbardziej, dofinansujmy takie dekodery, które sprawią, że PiS-owska szczujnia znów stanie się telewizją publiczną, z której można dowiedzieć się prawdy na temat afery Pegasusa, inwigilacji, szwindli na maseczkach, respiratorach, o wyborach kopertowych, niespotykanej wcześniej inflacji i setkach innych afer. Obawiam się jednak, że takie dekodery jeszcze nie istnieją. Przez chwilę miałem nadzieję, że pani nie ma na sali.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Beneficjenci tej ustawy będą mogli składać wnioski dotyczące wsparcia na zakup dekodera również za pośrednictwem placówek Poczty Polskiej. Nie odkryję chyba Ameryki, twierdząc, że wiele placówek pocztowych w naszym kraju już teraz nie radzi sobie z komfortową obsługą klientów.

W związku z tym, że - jak sami państwo zakładacie - ze wsparcia na zakup dekodera może skorzystać nawet 2 mln Polaków, w tym szczególnie osoby starsze, chciałbym zapytać, czy planujecie państwo przy tej okazji wprowadzenie dodatkowych rozwiązań w urzędach pocztowych, tak aby komfort dla klientów, a także dla pracowników poczty uległ znaczącej poprawie. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, klub Lewica. Szanowny Panie Ministrze!

Projekt tego nie przewiduje. Można by było np. to uczynić poprzez.

Czyli też byłoby bezgotówkowe rozwiązanie dla tych, którzy dokonali zakupu.

Dziękuję. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Mam wrażenie, że rząd nie wie, że na wynagrodzenie trzeba ciężko zapracować. Panie ministrze, kiedy rząd wykorzysta dane (Dzwonek), które zbierzecie, do tego, żeby ścigać ludzi za nieopłacony abonament telewizyjny?

Czy ci, którzy kupili, dostaną dopłatę do dekodera, czy będą inaczej traktowani niż ci, którzy czekają do ostatniej chwili? Druga sprawa.

Przyznajcie wreszcie, że jest to podatek, i przenieście to z poczty do urzędów skarbowych, bo poczta jest teraz.

Ale pociągnijmy to, ponieważ rzeczywiście jest tak, że wymyśliliście sobie, że będziecie dopłacać do dekoderów, a nie będziecie dopłacać do innego sprzętu. Dlaczego dekodery, dlaczego akurat to?

Panie pośle sprawozdawco, gdyby miał pan jakiś cynk, gdzie można zainwestować, żeby teraz szybko zarobić, ponieważ wprowadzacie taką ustawę, którą wymyśliliście pewnie wczoraj wieczorem, żeby ją dzisiaj wprowadzić, to chciałbym o tym wiedzieć, bo też lubię dobrze inwestować swoje pieniądze.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Chciałbym upomnieć się o grupę niepełnosprawnych, którzy mają problemy ze wzrokiem.

Możemy to zrobić i warto to zrobić. Dlatego, panie ministrze, proszę, żeby pan spróbował w taki sposób dokonać różnego rodzaju zmian i korekt w tym projekcje, żeby ta grupa takie wsparcie otrzymała. Jeżeli go zabraknie na poziomie legislacji sejmowej, a później senackiej i nie będzie takich poprawek, to w imieniu Lewicy zapowiadam, że będziemy dokładnie taki projekt chcieli przedłożyć, żeby właśnie tę grupę niepełnosprawnych wzrokowo wesprzeć. Pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Wysoka Izbo!

Grozi mu wtedy grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do 2 lat. Przecież taki przedsiębiorca odpowiada z art. 271 Kodeksu karnego za poświadczenie nieprawdy, bo poświadcza nieprawdę, że sprzedaje dekoder, sprzedając co innego.

Bardzo dziękuję. Pan poseł Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Panie Marszałku! Jeżeli ktoś w Sejmie, uchwalając prawo, w pierwszej kolejności myśli o tym, jak przy tej okazji zarobić, to sam sobie wystawia świadectwo.

Zainspirowało mnie ono i stąd moje pytanie do pana ministra, czy jest możliwe podjęcie w ministerstwie cyfryzacji prac badawczo-rozwojowych nad dekoderami osobistymi, bo jak widać, niektórzy koledzy parlamentarzyści potrzebowaliby takich, żeby odzyskać kontakt z rzeczywistością, podobnie jak ci, którzy nie zauważyli, że głosowaliśmy w tej Izbie za obniżką VAT-u kilka tygodni temu, że PIT został obniżony o 1 punkt procentowy, wprowadzony PIT-0 dla młodych do 26 lat. Pan poseł Grzegorz Napieralski, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wróćmy jeszcze do pytania o niepełnosprawnych.

Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz proszę o zabranie głosu sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pana Janusza Cieszyńskiego. Bardzo proszę, panie ministrze.

Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za pytania, dziękuję za te głosy w dyskusji. Pan poseł Napieralski pytał, czy uda się dotrzeć z tym przekazem. Tak jak mówiłem, jest planowana kampania i już teraz są prowadzone działania, które mają na celu uświadomienie, że ten stan, ta zmiana standardu nadchodzi. W momencie, w którym tylko wejdzie w życie ustawa, będziemy też mogli mówić o tych rozwiązaniach. Oczywiście zachęcam wszystkich państwa parlamentarzystów do tego, żeby wspólnie z nami informowali o tym, bo to jest, jak myślę, przekaz ponadpolityczny, ważny dla wielu wyborców. Także my tu oczywiście będziemy do państwa dyspozycji. Państwo wskazujecie, że nie zostały priorytetowo potraktowane potrzeby osób z niepełnosprawnościami. I tutaj miałem okazję zapoznać się z poprawką, którą państwo zgłosiliście. Tak jak wskazywałem, my jesteśmy skłonni w przypadku osób z niepełnosprawnościami nawet szerzej o tym wsparciu porozmawiać. Ja wiem, że czasu dzisiaj było niewiele, ale mamy jeszcze przed sobą pracę w Senacie. Tak jak mówię, w naszej ocenie warto o to zawalczyć, ponieważ to jest grupa ze szczególnymi potrzebami i tu jak zawsze rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie działał na rzecz tego, żeby potrzeby tej grupy były odpowiednio zaadresowane. O to też pytali inni państwo parlamentarzyści.

Tak jak już wskazywałem podczas posiedzenia komisji, mamy tutaj porozumienie pośród wszystkich operatorów telewizyjnych i oni za to nie wezmą ani złotówki, ponieważ to będzie emitowane jako ogłoszenie społeczne, zresztą to jest w interesie wszystkich nadawców, a nie tylko telewizji publicznej. Pani poseł Nowogórska pytała o kwestię związaną z danymi. Tutaj warto wyjaśnić jedną rzecz. Tym operatorem wyznaczonym nie będą te podmioty, które będą realizowały zakupy, tylko tym operatorem wyznaczonym będzie Poczta Polska. I tylko Poczta Polska będzie przetwarzała te dane, które obywatel oczywiście sam będzie widział, że je podaje. To będą proste dane teleadresowe. W naszej ocenie, a tutaj mamy ekspertów od bezpieczeństwa zarówno po stronie poczty, jak i po stronie kancelarii premiera, tutaj jakichkolwiek zagrożeń dla wycieków danych nie ma. W szczególności są wskazane też przeznaczenia, czyli te sposoby czy cele, na które będą przetwarzane te dane. I nie jest jednym z tych celów pobieranie opłat za abonament radiowo-telewizyjny, co niektórzy z państwa posłów w swoich wypowiedziach sugerowali. Pan poseł Dziambor nas co prawda opuścił, ale bardzo mnie dziwi, że jest taka krytyka tego projektu ze strony Konfederacji, dlatego że to jest, szanowni państwo, projekt po prostu 100-procentowo prowolnościowy. Państwo zarabia bardzo dużo pieniędzy na sprzedaży częstotliwości i w związku z tym, że ze względu na to tymi działaniami w pewnym sensie wywłaszcza Polaków z ich telewizorów, ponieważ z tych telewizorów w starych technologiach nie dałoby się już korzystać, oferuje uczciwą rekompensatę, nie za dużą, nie za małą, rynkową, tak, że każdy może tę szkodę, którą poniósł, sobie zrekompensować. To jest tak, jak w mojej ocenie powinno sprawne państwo funkcjonować. Pan poseł Gramatyka pytał o pomoc publiczną. Wielokrotnie już to wyjaśnialiśmy. Nie może o tym być mowy w tym przypadku, m.in. dlatego są te kryteria socjalne. Pan poseł Adamczyk pytał o szacunki, dlaczego 2270 tys. osób. Otóż, szanowny panie pośle, to jest szacunek, który został nam przedstawiony przez Krajowy Instytut Mediów na podstawie badań, które instytut przeprowadza. To jest jednostka powiązana z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Takie badania prowadzi. Lepszych informacji nie mamy i na tym się opieraliśmy. Pan poseł Szopiński pytał o kwestie związane z wynagrodzeniami pracowników Poczty Polskiej. To jest, szanowny panie pośle, decyzja zawsze po stronie Poczty Polskiej czy dowolnej innej spółki, która z nami współpracuje. Nie wchodzimy w to tak głęboko, natomiast to są dodatkowe środki, tak że bardzo często jest tak, że za dodatkowymi środkami, dodatkową pracą idzie też dodatkowe wynagrodzenie. Były też pytania o osoby, które już zdecydowały się na ten zakup. Tutaj warto wskazać, że mówimy o wsparciu, które ma charakter właśnie wsparcia socjalnego, czyli dotyczy osób, które nie były w stanie pozwolić sobie na taki wydatek. Dokonując takiego zakupu, niestety osoba, można powiedzieć, dowodzi, że tak w jej przypadku nie było.

Bardzo mi przykro, że skończył się czas, bo chciałem jeszcze powiedzieć coś o tych osobistych dekoderach, ale niestety nie zdążę. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm skierował ponownie ten projekt do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w związku z setną rocznicą urodzin Tadeusza Gajcego (druki nr 1988 i 1995) Proszę pana posła Mariusza Kałużnego o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowni Państwo!

Sama uchwała nie budziła żadnych kontrowersji wśród członków komisji. Treść uchwały została wypracowana na zasadzie kompromisu, przy uwzględnieniu wszystkich poprawek redakcyjnych i wszystkich najważniejszych poprawek wszystkich sił politycznych, które uznały, że warto, a nawet trzeba, w dniu dzisiejszym upamiętnić tego wspaniałego poetę, wielkiego Polaka. Propozycja ta została przyjęta jednogłośnie, przez aklamację, na posiedzeniu komisji kultury. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jako pierwszy pan poseł Mariusz Kałużny, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości i w imieniu własnym jako wnioskodawca chciałbym rekomendować państwu przyjęcie uchwały upamiętniającej Tadeusza Gajcego.

Tak, naród polski. Wspaniały poeta i wielki patriota. Działacz polskiego podziemia niepodległościowego. Przedstawiciel pokolenia Kolumbów, pokolenia, które życie poświęciło za ojczyznę. Brylant, którym pokryta jest korona Orła Białego. Pełnił funkcję redaktora naczelnego wydawanego w podziemiu miesięcznika literackiego ˝Sztuka i Naród˝, którego motto brzmiało: ˝Artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej˝ W czasach, kiedy tak ciężko o artystów, w czasach, w których coraz mniej atrakcyjne jest to, co narodowe, w których ciężko o narodową wyobraźnię, wspominamy wielkiego poetę, w którego twórczości przewodnim motywem była myśl o sensie ofiary w imię miłości do ludzi i ojczyzny, a kluczowymi kwestiami - oswajanie śmierci i wybór między nienawiścią a miłością, oczywiście na korzyść miłości. Tadeusz Gajcy był wreszcie żołnierzem Armii Krajowej. Na koniec napisał najtrudniejszy i najpiękniejszy wiersz: wiersz o poświęceniu życia dla ojczyzny, wiersz własnego życia, gdyż poświęcił własne życie za ojczyznę. Poległ wspólnie z przyjacielem poetą Zdzisławem Stroińskim w trakcie powstania warszawskiego w wysadzonej przez Niemców kamienicy. Dziś zawdzięczamy mu nie tylko piękną twórczość, ale również wolność naszej ojczyzny.

W 100. rocznicę jego urodzin pragnę w tej Izbie znowu odnieść się do wartości, które stanowią i rozwijają nasz naród. Są to kultura, wolność i miłość do ojczyzny.

Pani poseł Urszula Augustyn, Koalicja Obywatelska. 1 sierpnia 1993 r. na antenie Polskiego Radia Tadeusza Gajcego wspominała jego przyjaciółka Zofia Orszulska: ˝Był to chłopak wyjątkowego uroku. Niezbyt wysoki, świetnie zbudowany, bardzo ruchliwy i nawet wbrew tej swojej twórczości, która sięgała do katastrofizmu, tryskał humorem i wdziękiem˝ Czesław Miłosz o Gajcym mówił tak: ˝Wybuchowy, pełen radości życia, chciwy życia. Z tego powodu jego śmierć była tak dla mnie bolesna. I ze względu na obietnicę dużego talentu. Wtedy sądziłem nawet, że Gajcy ma większe możliwości niż Baczyński. Oczywiście trudno tu snuć przewidywania, kiedy ktoś umiera w tak młodym wieku˝ - tak wspominał po latach. Tadeusza Gajcego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego uważano za najwybitniejszych twórców pokolenia Kolumbów. Także Herbert, choć cenił wiersze Baczyńskiego, wolał poezję Gajcego: ˝Pisze językiem męskim, zdecydowanym, zaborczym, ale bezsilnym wobec potężnej zgrozy. Słowa jakby na krawędzi przepaści. Strofa równo odmierzona, kamienna˝ Tenże Zbigniew Herbert o materii wyobraźni organizującej u Gajcego treści uczuciowe mówił, że to materia z ognistego proroczego snu. Właśnie, marzenie spod znaku ognia - to jest chyba najbliższe temperamentowi Tadeusza Gajcego jako poety. Sam autor zresztą w swym testamencie poetyckim ˝Do potomnego˝ akt twórczy łączy z ciosaniem płomienia. Słowo poety jest zaś wysokie i ogniste. Z takich opinii przyjaciół i krytyków, z pozostawionych tekstów narysować można obraz niezwykłego poety: wrażliwego, przekraczającego granice wyobraźni i słów. Zdążył opublikować jedynie dwa tomiki wierszy, ale to te dwa tomiki zapewniły mu miejsce w historii literatury. Warto - należy, trzeba, to nasz obowiązek - wspomnieć także o tym, że to nie tylko poezja jest czymś, co plasuje go w naszych sercach i w historii. Od pierwszego dnia, od 1 sierpnia 1944 r. Tadeusz Gajcy pod pseudonimem Topór walczył w powstaniu warszawskim na Starym Mieście w drużynie szturmowo-wypadowej Chmury, czyli Zdzisława Stroińskiego. Zresztą obaj poeci zginęli w gruzach kamienicy, którą wysadzili Niemcy, więc zginęli w walce. Chcę zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz. W 2009 r. Muzeum Powstania Warszawskiego wydało płytę ˝Gajcy˝, na której utwory do tekstów poety wykonują współcześni muzycy: Maleo, Kazik, Dezerter czy Lech Janerka. Jest też płyta, na której wiersze Tadeusza Gajcego recytowane są przez Borysa Szyca z towarzyszeniem muzyki skomponowanej przez Adama Pierończyka. To są piękne świadectwa tego, jak poezja Gajcego, człowieka, który oddał życie w obronie ojczyzny, w walce za ojczyznę, poezja trudna i wrażliwa jest dziś ważna (Dzwonek), aktualna i do dziś rozważana.

Pani poseł Małgorzata Prokop-Paczkowska, Lewica. Wysoka Izbo! Kiedy podejmujemy decyzję o uchwałach rocznicowych, a szczególnie jeśli dotyczą one artystów, chciałoby się, aby przechodziły bez kontrowersji. W tym przypadku właściwie tak było. Ale pewne pytania trzeba zadać. Tadeusz Gajcy to wybitny poeta czasu wojny, żołnierz AK, który zginął w powstaniu warszawskim, ale też członek Konfederacji Narodu, organizacji konspiracyjnej o charakterze polityczno-wojskowym utworzonej w środowisku działaczy ONR-Falanga, czyli polskich faszystów. Na szczęście w swojej pracy redakcyjnej Gajcy odciął się od tej faszystowskiej, antysemickiej ideologii. Konfederacja Narodowa liczyła na zwycięskie zakończenie wojny i budowę imperium słowiańskiego z dominującą rolą Polski w granicach sprzed pierwszego rozbioru. Gajcy oddał życie za ojczyznę, ale czy musiał, czy powinien? I tu trzeba zadać pytanie, czy decyzja dowódców o wybuchu powstania skazująca niechybnie młodych ludzi na śmierć była decyzją słuszną. Bo syn polskiego imperium do powstania szedł wyposażony w jeden granat. Jego przyjaciel Zdzisław Stroiński, inny poeta dysponował pistoletem bez pocisków. W swoim ostatnim wierszu, który stworzył podczas powstania napisał: ˝Wszyscy święci, hej do stołu! W niebie uczta: polskie flaczki,/ Wprost z rynsztoków Kilińskiego! Salcesonów misa pełna/ Świeże chrupkie. Do godów, święci, do godów,/ Przegryźcie/ Chrystusem Narodów! Ten ostatni wiersz zapisał na papierowej torbie, widząc skutki masakry mieszkańców Warszawy. Jacek Cieślak na łamach ˝Rzeczpospolitej˝ napisał: ˝Trudno się dziwić, że Gajcy swym szyderczym wierszem postawił krzyżyk na mesjanizmie swojego środowiska, które dziś znów odżywa˝ Lewica poprze uchwałę upamiętniającą poetę Gajcego. Bardzo proszę, pan poseł Jarosław Rzepa, Koalicja Polska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mało jest poetów, których życie stało się symbolem losu całego pokolenia. Niewątpliwie należy do nich Tadeusz Gajcy, jeden z najważniejszych przedstawicieli rocznika 1920. Nazwano ich Kolumbami, bo odkryli nieznany wcześniej kontynent terroru, cierpienia, strachu i śmierci. Wybitnie utalentowany poetycko, redaktor podziemnego czasopisma ˝Sztuka i Naród˝, przekonany o swojej wyjątkowości, żył jak jego rówieśnicy - intensywnie, szybko i twórczo, czując nadchodzącą śmierć. Opublikował dwa szczupłe tomiki poetyckie, które przeszły do historii literatury. Do dziś zwracają uwagę oryginalną fantastyką, którą przeszywa lęk, dziecięcą wrażliwością utkaną z obrazów apokaliptycznej grozy, wreszcie poczuciem absurdu chwili dziejowej, obserwowanej z niedowierzaniem - jak rodzaj przerażającej groteski. Po blisko 80 latach od śmierci Gajcego muszą nas nurtować pytania: Kim był ten młodziutki poeta i dramaturg? Co wiązało go z ultraprawicowym środowiskiem ˝Sztuki i Narodu? Czym wzbudził niechęć Czesława Miłosza, co diametralnie zmieniło się po latach? Pod czyim nazwiskiem ukrywa się w powieści ˝Kolumbowie.

W pierścieniu śmierci˝ prześwietla tragiczne życie poety, sięgając do wspomnień rodziny oraz znajomych, ale przede wszystkim dogłębnie analizując jego twórczość.

Dziękuję wnioskodawcy za jego przygotowanie.

Wysoka Izbo! Pokolenie, które wchodziło w swoją dorosłość w latach II wojny światowej, było być może najlepszym pokoleniem, jakiego doczekała się nasza ojczyzna w swojej ponadtysiącletniej historii. A wśród tych najlepszych synów i córek naszego narodu jednym z najwybitniejszych artystów był właśnie on - Gajcy. Był to człowiek, który zapisał się w polskiej literaturze, w polskiej poezji, w polskiej historii, w polskiej pamięci jako postać wybitna, nietuzinkowa, jako niesamowity potencjał, mimo że zginął, mając 22 lata. I nie tylko on przecież ze środowiska sztuki i narodu, można choćby wymienić Trzebińskiego czy innych. Tak, z tego środowiska sztuki i narodu, które było niejako artystycznym, kulturalnym ramieniem Konfederacji Narodu, które w ciemnych latach okupacji niemieckiej i sowieckiej, w ciemnych latach terroru brunatnego i czerwonego doskonale rozumiało, że trzeba budzić ducha Polaków, że nie można zohydzać pamięci, tożsamości narodowej, że sztuka nie jest po to, żeby gorszyć, prowokować, szokować, że sztuka jest po to, żeby inspirować, żeby nieść natchnienie, żeby dawać nadzieję, żeby nieść dobro. Jakże to znamienne i jakże aktualne w dzisiejszym świecie. Jakże aktualne w dzisiejszym świecie postmodernizmu, brzydoty i zniekształcenia sztuki w happening, prowokację, w obrazoburstwo. Jakże charakterystyczne, że nawet przy okazji tej uchwały ze strony Lewicy musieliśmy usłyszeć atak. Atak na co? Na Gajcego? Na dwudziestodwulatka, który oddał życie za Polskę? Nie. Atak na to, co on reprezentował sobą: tożsamość narodową, dążenie do tego, żeby Polska była państwem wielkim, żeby naród był narodem wielkim, o wielkich aspiracjach, a nie zagrzebanym w swoje słabości, w swoje uwikłania. I wreszcie ten atak idzie z prostego powodu - ponieważ tak jak Konfederacja Narodu, tak jak Narodowe Siły Zbrojne, Narodowa Organizacja Wojskowa, będąca fundamentem po scaleniu Armii Krajowej, te środowiska wiedziały, że w latach 40. Polska (Dzwonek) ma dwóch wrogów: pierwszego - brunatnego, niemieckiego okupanta i drugiego, który szedł ze wschodu - czerwonego, totalitaryzm komunistyczny, który przyniósł również ze sobą tych, którzy dzisiaj siedzą po tej stronie sali, ich spadkobierców. Dziękuję. Dziękuję. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. A nie, przepraszam. Przepraszam bardzo. Jeszcze są pytania. Pan poseł Jan Szopiński z Lewicy chce o coś spytać.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie ma życiorysów białych i czarnych. Dzisiaj uchwałą Sejmu czcimy 100. rocznicę urodzin Tadeusza Gajcego, który oddał swoje życie za ojczyznę i był wyjątkowym poetą, który zginął na powstańczej reducie. 100. rocznica jego urodzin to doskonały czas, aby w programach szkolnych przypomnieć jego twórczość, nieco już zapomnianą. W związku z tym mam apel do ministerstwa edukacji, aby dzisiejsza uchwała Sejmu nie skończyła tylko jako uchwała Sejmu, aby rzeczywiście w programach szkolnych powróciła twórczość Tadeusza Gajcego nieco szerzej niż dotychczas. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Oczywiście myślę, że są tacy ludzie, zdarzenia i rzeczy, które łączą. Wydaje się, że Gajcy jest taką osobą. Jego poezja, jego patriotyzm to są rzeczy, które łączą, które można rozpatrywać w sposób pozytywny, pokazując drogę, którą młodzi ludzie mogą podążać.

Dziękuję bardzo. Pani poseł Paulina Matysiak, klub Lewicy. Wysoka Izbo! Sejm ma zamiar upamiętnić w 100. rocznicę Tadeusza Gajcego, poetę, studenta polonistyki na tajnych kompletach, przedstawiciela pokolenia Kolumbów i młodego patriotę, który zginął w wieku 22 lat, biorąc czynny udział w powstaniu warszawskim jako żołnierz Armii Krajowej. Tadeusz Gajcy, mimo że związany ze środowiskiem narodowców, nie był zaślepiony skrajną ideologią, lecz bardziej skłonny do pojednania z pisarzami o innych poglądach. Patriotyzm w jego twórczości jest szczery i głęboko przeżywany. W jego wierszach odnajdziemy apokaliptyczną wizję i rzeczywistość ukazaną za pomocą bogatej symboliki. Łączył ze sobą rzeczywistość ze światem snu, oswajał śmierć i dokonywał wyboru między miłością a nienawiścią. W jego poezji wybrzmiewa głos młodych ludzi, którym okrucieństwo wojny odebrało szansę na wejście w dorosłość. Niech to będzie dzisiaj dla nas, polityków, swego rodzaju memento. Pani poseł Hanna Gill-Piątek, Polska 2050. Nie widzę pani poseł. To teraz już rzeczywiście lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Zamykam dyskusję. Do głosowania nad projektem uchwały przystąpimy w bloku głosowań.

Stwierdzam kworum. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawiła opinię dotyczącą wniosku w sprawie wyboru kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, druk nr 1987. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tej sprawy. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych, druk nr 2003. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Powracamy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w związku z setną rocznicą urodzin Tadeusza Gajcego. Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały z druku nr 1995. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 1995, zechce nacisnąć przycisk.

456 - za, 1 - przeciw, 1 się wstrzymał. Sejm podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia Tadeusza Gajcego w 100. rocznicę urodzin. Powracamy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1975. Komisje przedstawiają również wnioski mniejszości, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. W 4. wniosku mniejszości do art. 6 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wnioskodawcy proponują dodać ust. 5b. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosków mniejszości 1. i 4., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wnioski mniejszości odrzucił. Wnioski mniejszości 2. i 3. zgłoszone zostały do art. 1 projektu ustawy zawierającego zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1975, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1977-A. Proszę pana posła Jarosława Sachajkę o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Panowie Premierzy! Wysoka Izbo! Dzisiaj o godz. 12 odbyło się drugie czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, druki nr 1611 i 1977. W trakcie drugiego czytania złożono osiem poprawek.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1977. Komisja w dodatkowym sprawozdaniu przedstawia poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Wszystkie poprawki zostały zgłoszone do art. 1 projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Komisja wnosi o ich odrzucenie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 2. i 4., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawki odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Komisja wnosi o jej przyjęcie.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Proszę państwa, mogę prosić troszeczkę ciszej, bo przestaję słyszeć samą siebie.

Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1977, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który poddam pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczać, że Sejm, zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu, skierował ten projekt ustawy do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 1913, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował ten projekt ustawy do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia. Powracamy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacji i Nowoczesnych Technologii o pilnym rządowym projekcie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1996-A. Proszę pana posła Radosława Fogla o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Dzisiaj na posiedzeniu Sejm skierował pilny rządowy projekt ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej ponownie do Komisji Cyfryzacji, Innowacji i Nowoczesnych Technologii.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1996. Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności. Komisja wnosi o odrzucenie tych poprawek. Ich przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 2. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy.